Wysoka Izbo! Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji: - Etyki Poselskiej - godz. 10.30, - Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 10.30, - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 11, - Finansów Publicznych - godz. 11, - Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - godz. 11, - Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 11, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 11, Zdrowia - godz. 11, - Edukacji, Nauki i Młodzieży wspólnie z Komisją Zdrowia - godz. 12, - Kultury i Środków Przekazu - godz. 12, Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach - godz. 12, - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 12.30, - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 12.30, - Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - godz. 13, - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 13, - Finansów Publicznych - godz. 13.30, Infrastruktury wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - bezpośrednio po zakończeniu wspólnego posiedzenia komisji zwołanego na godz. 11, ok. godz. 14, Łączności z Polakami za Granicą - godz. 14, - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 14.30, - Administracji i Spraw Wewnętrznych - godz. 15, - do Spraw Służb Specjalnych - godz. 15, - Infrastruktury - godz. 15, - Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 15, - Gospodarki i Rozwoju - godz. 16, - Obrony Narodowej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych - godz. 16, - Finansów Publicznych - godz. 16.30, - Obrony Narodowej - godz. 17, - Polityki Społecznej i Rodziny - godz. 17, - Spraw Zagranicznych - godz. 17, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - godz. 18, - Finansów Publicznych - godz. 18.30, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 19, Gospodarki i Rozwoju wspólnie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 20. W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia następujących zespołów parlamentarnych: - Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Każdym Rozmiarze - godz. 12, - Parlamentarnego Zespołu ds. uregulowania ustawowego polityki górskiej - godz. 19. W imieniu pani poseł Ewy Kołodziej, przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, oraz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w ramach obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w Sejmie RP zapraszamy państwa do bezpłatnego badania poziomu cukru we krwi. Badania pozwolą poznać poziom glikemii oraz, w razie potrzeby, skorzystać z porady edukacyjnej i pogłębionej diagnostyki.

Dziękuję. Proszę państwa, zanim przystąpimy do wniosków formalnych, bo takie mamy, chciałam państwu przypomnieć, że dzisiaj rano wszyscy posłowie otrzymali SMS-y informujące o tym, że obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek na sali plenarnej w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań, także wśród pracowników naszego parlamentu.

Proszę nie krzyczeć, bo wie pan.

Nie ma zgody na narażanie cudzego zdrowia. Panie pośle, już panu powiedziałam, że decyzją sądu, do którego pan się na mnie skarżył, skarga została uchylona, a właściwie odsunięta, w związku z tym, że Sejm, marszałek ma prawo wydawać takie zarządzenia. Ma zwolnienie lekarskie. Ja widzę, kto ma zwolnienie lekarskie, dlatego tych posłów nie upominam, natomiast pozostali - nie. Mogę prosić? Bardzo proszę, pan poseł Bosak, pan poseł Kulesza, pan poseł Braun, pan poseł Dziambor ma zwolnienie, pan poseł Sośnierz, pan poseł Urbaniak, pan poseł Kamiński też ma zwolnienie, i pan poseł Berkowicz.

Pan poseł Bosak założył, dobrze. Pozostali panowie nie, tak? Zwracam się do panów posłów Kuleszy, Brauna, Sośnierza, Urbaniaka i Berkowicza.

Pan Sośnierz ma zwolnienie lekarskie.

Panowie posłowie Kulesza, Braun, Kamiński i Berkowicz, na podstawie art. 175 ust. 5, w związku z tym, że nadal panowie uniemożliwiają prowadzenie obrad, podejmuję decyzję o wykluczeniu panów z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę panów o opuszczenie sali plenarnej.

Pani poseł Karolina Pawliczak, Lewica.

Wysoka Izbo! Składam wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w sprawie uzupełnienia informacji ministra sprawiedliwości i ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie skandalicznych wydarzeń, tego, co wydarzyło się w naszym mieście - Kaliszu, gdzie nacjonaliści spalili w centrum miasta Statut Kaliski. Działo się to wszystko pod osłoną czy pod parasolem służb, Policji. Prosimy o informację, dlaczego tak się stało. Kaliszanie, mieszkańcy naszego miasta, oczekują dokładnych informacji w tej sprawie. Są tu, na tej sali, posłowie i posłanki z naszego wspólnego okręgu. Oczekujemy szczegółowych informacji w tej sprawie. Szanowni Państwo!

Pani poseł, mówienie, że nic się nie robi w tej sprawie, jest po prostu nieprawdą. Ponieważ padł wniosek formalny o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Jako mieszkaniec Kalisza chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, bardzo stanowczo tutaj zareagować. Osoby, które dopuściły się tego haniebnego czynu, są już zatrzymane. Reakcja ministra spraw wewnętrznych i administracji jest natychmiastowa. Ponieważ padł wniosek o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw?

Sejm wniosek odrzucił. Wniosek formalny - pani poseł Małgorzata Tracz, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Polski rząd nie wykorzystał szansy, by przedstawić krajowe cele klimatyczne na tym szczycie. Zamiast tego dostał tytuł skamieliny dnia za kluczenie w sprawie daty odejścia od węgla. Hańba. A tymczasem w porozumieniu końcowym szczytu są jasne zapisy, że czas węgla w energetyce się kończy, a zaczyna się czas energii ze źródeł odnawialnych. Chcemy jasnej informacji, co poza ośmieszeniem Polski robiła polska delegacja na szczycie klimatycznym. W jaki sposób wdroży porozumienia zawarte w Glasgow? Dziękuję, pani poseł. Ponieważ padł wniosek o odroczenie posiedzenia, poddam ten wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050. Wysoka Izbo! Zakończył się szczyt klimatyczny w Glasgow, a my nadal jesteśmy jedynym krajem w Unii, który nie ogłosił konkretnej daty odejścia od węgla. Przez chwilę wydawało się, że rząd zdecydował się na deklarację odwrotu od paliw kopalnych w jednym terminie z krajami rozwiniętymi, czyli do końca lat 30., jednak wycofaliśmy się rakiem z tych obietnic. Wszyscy czuliśmy jakiś wstyd, kiedy rząd umieścił nas w szeregu krajów rozwijających się, które w podróży ku przyszłości wybrały wagon dla palących i będą w nim siedzieć do 2049 r. A podobno tak świetnie ma się nasza gospodarka.

Wysoka Izbo! W Polsce znowu morduje się księży. Zaczęło się od przypisywania win w ramach odpowiedzialności zbiorowej ogółowi ludzi Kościoła. A potem? Potem zaczęło się szczucie. Agresja słowna - tego byliśmy świadkami. Agresja słowna, potem profanowanie symboli religijnych, szydzenie z tego, co dla Polaków najświętsze, demolowanie miejsc kultu. Potem mieliśmy do czynienia również z dehumanizacją katolików i osób duchownych. Zaczęło się także wzywanie do przemocy, a następnie były same akty przemocy i agresji fizycznej, pobicia.

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałem przedstawić powody wystąpienia z rządową inicjatywą legislacyjną w zakresie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 1729. Ta inicjatywa w postaci nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych spowodowana jest podnoszonymi przez jednostki samorządu terytorialnego postulatami dotyczącymi uszczelnienia systemu zwolnień od podatku od nieruchomości dla nieruchomości kolejowych w związku z wykorzystywaniem gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze, który nie jest związany z kolejnictwem. Zwracam się do państwa posłów o wyciszenie rozmów, ewentualnie przeniesienie ich poza salę sejmową, ponieważ uniemożliwiamy wystąpienie panu ministrowi. Panie senatorze, zapraszamy. Jeszcze chwilkę, panie ministrze. Panie senatorze, proszę zająć miejsce.

Dziękuję bardzo.

W projekcie doprecyzowuje się zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości w obszarze zwolnienia dla nieruchomości kolejowych w celu uszczelnienia systemu zwolnień i kompleksowego uregulowania tego obszaru. Proponowane zwolnienia od podatku od nieruchomości obejmują grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiektu infrastruktury usługowej, w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym, w części zajętej wyłącznie do wykonywania zadań zarządcy infrastruktury lub świadczenia usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej, jeżeli infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są udostępniane przewoźnikom kolejowym lub infrastruktura kolejowa lub obiekt infrastruktury usługowej są wykorzystywane do przewozu osób, lub infrastruktura kolejowa tworzy linie kolejowe szerokotorowe, lub infrastruktura kolejowa stanowi infrastrukturę nieczynną. Drugi punkt w zakresie tego zwolnienia obejmuje grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych. Trzecia część to nieruchomości inne niż określone powyżej, stanowiące obszar kolejowy, z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności innej niż kolejowa. Ten postulat dotyczący uszczelnienia systemu sprowadza się do dookreślenia tego, że dana nieruchomość zwolniona jest z podatku od nieruchomości wyłącznie w takiej części, w jakiej zajęta jest na prowadzenie działalności kolejowej w ramach wskazanych przed chwilą obszarów, poprzez powiązanie zwolnienia z wykonywaniem działalności kolejowej polegającej na zarządzaniu infrastrukturą kolejową, obiektem infrastruktury usługowej, wykonywaniem usług związanych z bezpośrednią obsługą podróżnych, wykorzystywaniem infrastruktury lub obiektu do przewozu osób. Chciałem zwrócić państwa uwagę na to, że przed implementacją w 2016 r. dyrektywy 34 w sprawie ustanowienia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego do polskiego porządku prawnego infrastrukturę kolejową stanowiły wszystkie elementy kolejowe stanowiące całość techniczno-użytkową, umożliwiające przewóz osób lub rzeczy. Wraz z implementacją ww. dyrektywy nastąpiła zmiana nomenklatury, co spowodowało rozróżnienie na infrastrukturę kolejową, obejmującą co do zasady linie i bocznice kolejowe, oraz na obiekty infrastruktury usługowej, obejmujące elementy infrastruktury przeznaczone do m.in. zestawiania składów pociągów lub wykonywania manewrów oraz przeładunków, jak również stanowiące stacje pasażerskie, zaplecza techniczne, tory postojowe i inne instalacje niezbędne do niezakłóconego i bezpiecznego prowadzenia transportu kolejowego. Z tego względu istotne jest, by wszystkie elementy umożliwiające w ujęciu funkcjonalnym transport towarów lub osób były objęte zwolnieniem. Z tego też powodu zwolnieniem od podatku od nieruchomości objęto infrastrukturę kolejową, jak i obiekty infrastruktury usługowej. Zwolnieniem proponuje się objąć również linie kolejowe szerokotorowe, analogicznie do obowiązującego stanu prawnego. Objęcie zwolnieniem podatkowym infrastruktury nieczynnej jest zasadne z uwagi na konieczność zachowania tej infrastruktury, jak również z uwagi na to, że ze zwolnienia podatkowego nie korzystałaby infrastruktura wyłączona z ruchu w celu jej modernizacji. Przez infrastrukturę nieczynną, zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym, należy rozumieć infrastrukturę, na której zarządca infrastruktury nie dopuścił prowadzenia ruchu. Literalnie oznacza to, że będzie to infrastruktura zarządzana przez podmiot, który ma status zarządcy infrastruktury, na której nie jest prowadzony ruch. Zwolnienie dla części nieruchomości przeznaczonych na świadczenie usług bezpośrednio związanych z obsługą podróżnych ma na celu doprecyzowanie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla tych elementów obiektów infrastruktury pasażerskich, których utrzymywanie jest niezbędne z uwagi na oczekiwania społeczne. Po pierwsze, projektowane zwolnienie warunkowane jest świadczeniem usług przez przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej. Po drugie, zwolnienie obejmować będzie jedynie część nieruchomości zajętą na świadczenie usług związanych z bezpośrednią obsługą podróżnych. I po trzecie, pojęcie usług bezpośrednio związanych z obsługą nie budziło do tej pory wątpliwości. Jednak celem uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych w uzasadnieniu projektowanej ustawy wyszczególniono elementy związane z bezpośrednią obsługą podróżnych. Do elementów podlegających zwolnieniu podatkowemu należy zaliczyć ogólnodostępne powierzchnie bezpośrednio związane z obsługą podróżnych przez przewoźnika kolejowego lub operatora stacji pasażerskiej obejmujące: poczekalnie, hole dworcowe i antresole, wydzielone pomieszczenia dostosowane do karmienia i przewijania dzieci, toalety, dostęp do terenów zielonych, np. dla pasażerów podróżujących ze zwierzętami, powierzchnie przed kasami biletowymi, powierzchnie zajęte przez kasy biletowe i inne powierzchnie przeznaczone do sprzedaży biletów, punkty informacyjne, piesze ciągi komunikacyjne, powierzchnie zajęte pod dźwigi osobowe i inne urządzenia służące przemieszczaniu się osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się, pochylnie, kładki dla pieszych, wiaty osłaniające przed czynnikami atmosferycznymi, miejsca parkingowe i postojowe dla pojazdów, powierzchnie stanowiące dostęp z drogi publicznej do peronów, dworca kolejowego lub innej przestrzeni ogólnodostępnej, ciągi dojazdowe do parkingów wraz z infrastrukturą - dźwigi towarowe, elementy najazdowe, pochylnie, wiadukty, tunele - powierzchnie służące do umieszczania dodatkowych informacji dla pasażerów wyznaczone przez operatora stacji pasażerskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, powierzchnie stanowiące zaplecze techniczne w części służącej prawidłowemu funkcjonowaniu ww. elementów stacji pasażerskich.

Przykładem są m.in. miejsca parkingowe i postojowe dla pojazdów udostępniane na potrzeby pasażerów transportu publicznego zbiorowego, takie jak parkingi Park & Ride, stanowiska Bike & Ride, służące do przesiadania się podróżnych z innego środka transportu: samochodu, motocykla, roweru, hulajnogi itd. do pociągu. Rozwiązanie to ma również umożliwić przekształcenie stacji pasażerskich w węzły komunikacyjne łączące różne gałęzie i rodzaje transportu: samochodowego z kolejowym, dalekobieżnego z miejskim, rowerowego z kolejowym - tu można wprowadzać różne elementy. Jeśli chodzi o ostatnią kwestię, którą chciałem poruszyć, czyli zwolnienie dla pozostałych nieruchomości niezajętych na prowadzenie działalności komercyjnej - są to co do zasady nieużytki kolejowe - to objęcie podatkowym zwolnieniem gruntów, budynków i budowli położonych na obszarze kolejowym, które nie są wykorzystywane do innej niż kolejowa działalności, jest uzasadnione dla utrzymania dotychczasowego zwolnienia podatkowego dla m.in. takich gruntów kolejowych, jak międzytorza czy pasy bezpieczeństwa, jak również nieruchomości utrzymywanych jako rezerwa pod przyszłe potrzeby sektora kolejowego, w tym inwestycyjne. Bez wprowadzenia tego przypisu powyższe nieruchomości zostałyby objęte podatkiem od nieruchomości w związku z brzmieniem przepisu uszczelniającego system, ponieważ wcześniej wskazane zwolnienie podatkowe dotyczy jedynie części nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie zadań zarządcy infrastruktury lub operatora obiektu infrastruktury. Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie niniejszego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Bardzo serdecznie witam pana senatora i proszę o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy zawartego w druku nr 919. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Senat proponuje państwu przyjęcie krótkiej ustawy, która likwiduje ewidentną lukę podatkową w podatku od nieruchomości, który to podatek jest dochodem gmin. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniła art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Suma strat, która jest dość trudna do określenia, przez związki samorządowe jest szacowana na ponad 1 mld zł w tym okresie, czyli to są naprawdę znaczące pieniądze. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten podatek nie jest tracony równo przez wszystkie gminy, tylko na bardzo dużą skalę przez nieliczne, to prowadzi to do wniosku, że część gmin znalazła się w bardzo złej sytuacji finansowej.

Podobny zapis jest w projekcie rządowym.

Mianowicie rozszerza zwolnienie, jeśli chodzi o infrastrukturę usługową wykorzystywaną na świadczenie usług dla pasażerów i obsługi ruchu kolejowego, przy czym są też zastrzeżenia związane z tym, że usługa może być związana tylko z zadaniem zarządcy infrastruktury albo ze świadczeniem usług przez operatora w rozumieniu ustawy o transporcie kolejowym. Te zabezpieczenia wydają się wystarczające, ale pozostaje obawa o skuteczność tych zapisów, dlatego że mamy doświadczenia sprzed 5 lat, kiedy też się wydawało, że ustawa, mówiąc kolokwialnie, jest szczelna, a tworzyła lukę podatkową. Drugim rozszerzeniem jest nowe rozszerzenie o infrastrukturę nieczynną ze zwolnieniem bezterminowym z podatku od nieruchomości tej nieczynnej infrastruktury. Uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. W uzasadnieniu jest podane, że powodem tego zwolnienia jest prowadzenie modernizacji i remontów, które z natury mają charakter czasowy, dlatego zwolnienie bezterminowe moim zdaniem jest błędem. Podatek od nieruchomości ma nie tylko funkcję fiskalną, skłania również do aktywnego gospodarowania nieruchomościami. W sytuacji gdy zwolnienie będzie bezterminowe, nie będzie istotnej motywacji do aktywnego gospodarowania tą infrastrukturą i będzie to w jeszcze większym stopniu prowadziło do utrzymywania, często w centrach miast, zaniedbanej infrastruktury, która jest fatalną wizytówką. Od tego powinniśmy odchodzić.

O to wnoszę i bardzo o to proszę, dlatego że, tak jak mówiłem, problem może nie dotyczy bardzo wielu samorządów, ale tych, których dotyczy, dotyczy w sposób dramatycznie mocny. To są często małe gminy, które nie mają zdywersyfikowanych źródeł dochodów, i ubytek w tej dziedzinie jest dla nich wyjątkowo bolesny. Większych gmin też to dotyczy, ale tam ta baza podatkowa jest szersza. Do takich większych miast należy Oświęcim czy Swarzędz.

Mianowicie znane są przypadki scalania gruntów po to, aby na dużym obszarze, na którym tylko mała część jest zajęta pod infrastrukturę kolejową, a prowadzona jest duża działalność gospodarcza spoza branży kolejowej, było zwolnienie z podatku od nieruchomości. To jest nieuzasadniona pomoc publiczna i zupełnie niedopuszczalna strata w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję panu senatorowi. Zachęcam do pozostania i wzięcia udziału w dyskusji, która będzie się toczyła na sali sejmowej. Sejm ustalił, że w łącznej dyskusji nad tymi punktami porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Mariusz Trepka, który przedstawi stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 1729, i wobec senackiego projektu ustawy, druk nr 919. Omawiany projekt dotyczy doprecyzowania zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o grunty kolejowe, w szczególności grunty zajęte na prowadzenie działalności przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów obiektów infrastruktury usługowej. Projektowane rozwiązania uszczelniają system zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem. W konsekwencji projektowane rozwiązania wyeliminują nadużycia interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów przez część przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności zarządcy na rynku kolejowym, wykorzystują przepis do unikania opodatkowania i powodują uszczuplenie wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin. Zwolnienia od podatku od nieruchomości dotyczące infrastruktury kolejowej były wprowadzane od początku obowiązywania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Do dziś zwolnienia od podatku są cały czas tożsame i obejmują grunty kolejowe. Ale z uwagi na wdrożenie do polskiego systemu prawnego prawa Unii Europejskiej zmieniła się nomenklatura. Dlatego to, co jeszcze 6 lat temu było infrastrukturą kolejową, obecnie stanowić może obiekt infrastruktury usługowej funkcjonujący i działający w ramach systemu kolei ujednolicanego przez prawo Unii Europejskiej. Projektowany przepis pozwoli na obciążanie podatkiem części gruntów, budynków lub budowli wykorzystywanych do działalności komercyjnej, tj. np. dzierżawionych, wynajmowanych przez podmioty prowadzące inną działalność niż przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskiej. W projektowanej ustawie dodaje się również nowy punkt, który ma zmniejszać obciążenia podatkiem od nieruchomości za grunty, budynki i budowle, które nie są wykorzystywane do żadnej działalności, a są utrzymywane jako rezerwa gruntów, budynków i budowli na potrzeby rozwoju sektora kolejowego, w tym przyszłych inwestycji. Jednocześnie wprowadza się wyjątek, w którym prowadzenie na takim gruncie działalności gospodarczej innej niż kolejowa będzie skutkowało brakiem zwolnienia od podatku od nieruchomości. Wejście w życie powyższych regulacji powinno skutkować zwiększeniem wpływów podatkowych do części budżetów gmin w związku z uszczelnieniem korzystania ze zwolnień z opodatkowania w obszarze kolejnictwa.

Takie rozwiązanie pozwoli również na zbadanie nowych regulacji i przeprowadzenie odpowiednich procedur w kontekście ewentualnego wystąpienia pomocy publicznej w stosunku do terminali towarowych. Warto zauważyć, że w Sejmie został złożony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk sejmowy nr 919, który problem nadużywania zwolnień od podatku od nieruchomości rozwiązuje ułomnie, powodując ryzyko dalszego wykorzystywania zwolnień przez przedsiębiorców nieprowadzących działalności na rynku kolejowym.

Dlatego też projekt rządowy zasługuje na jak najszybsze uchwalenie, bo z jednej strony uszczelnia system podatkowy, a z drugiej strony promuje transport kolejowy i jego rozwój jako bezpieczny i ekologiczny środek transportu zarówno osób, jak i towarów. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pragnę przekazać, że klub będzie pracował nad oboma projektami ustaw o zmianie ustawy o podatkach i opłatach kolejowych, druki nr 1729 i 919. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi za przedstawienie stanowiska. Teraz w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pani poseł Zofia Czernow. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: senackiego projektu ustawy zawartego w druku nr 919 i rządowego projektu ustawy zawartego w druku nr 1729. Celem wymienionych projektów ustaw jest doprecyzowanie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości określonego w art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w obszarze zwolnienia gruntów kolejowych.

Senacki projekt ustawy doprecyzowuje i zawęża przepisy w art. 7, który to artykuł określa zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości. Projekt wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym zwolnienie nie będzie dotyczyło całej działki ewidencyjnej, jak to jest obecnie, określonej jako działka kolejowa, lecz wyłącznie tej jej części, na której znajdują się elementy infrastruktury kolejowej, które są wykorzystywane do celów określonych w ustawie o transporcie kolejowym. Podkreślić należy, że projekt senacki, uszczelniający podatek od nieruchomości i bardzo oczekiwany przez samorządy, wpłynął do Sejmu równo rok temu i cały rok czekał na procedowanie. Powstaje pytanie: Dlaczego tak długo? Projekt rządowy zawiera przepisy, które również likwidują lukę podatkową. W tej części projekty te są zbieżne i nie budzą wątpliwości. Czym różnią się te projekty? Po pierwsze i najważniejsze, terminem wejścia w życie oczekiwanych zmian. Projekt rządowy proponuje wejście w życie 1 stycznia 2023 r., głównie z powodu uniknięcia zarzutu naruszenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego. Zgodnie bowiem z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego z 2001 r. i 2005 r. zmiany dotyczące podatków, których wymiar podatkowy jest dokonywany za okres roczny, powinny być ogłaszane co najmniej miesiąc przed końcem poprzedniego roku podatkowego. Powstają pytania. Dlaczego rząd tak długo zwlekał ze swoim projektem, aż powstało niebezpieczeństwo przekroczenia terminu jednego miesiąca przed końcem roku podatkowego? A przecież uszczelnianie podatków to priorytet rządu. Wyrażam nadzieję, że rząd i Sejm dobrze wykorzystają ten wprawdzie krótki, ale jeszcze możliwy czas, żeby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2022 r. Projekt rządowy wprowadza dodatkowe ulgi w podatku od nieruchomości, a mianowicie zwolnienie od podatku tzw. infrastruktury usługowej związanej z kolejnictwem, bezterminowe zwolnienie infrastruktury nieczynnej, która jest wyłączona czasowo z uwagi na planowane remonty i modernizację, zwolnienie gruntów, które stanowią rezerwy dla rozwoju kolejnictwa. Te propozycje dodatkowych ulg budzą wątpliwość, a zwłaszcza bezterminowe zwolnienie nieczynnej infrastruktury, która ma być według projektu wyłączona czasowo. W naszym przekonaniu ten czas zwolnienia należy precyzyjnie określić i przyjąć np. najbardziej odpowiedni, 5-letni czas zwolnienia. Do tej pory były to - przypominam - 3 lata. Mając nadzieję na wnikliwe rozpatrzenie wątpliwości dotyczących dodatkowych ulg oraz konstruktywne ustalenie vacatio legis, wnioskuję o skierowanie projektów do dalszych prac legislacyjnych. Proszę teraz pana posła Roberta Obaza o przedstawienie stanowiska klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest wyczekiwana przez gminy w całej Polsce, szczególnie przez te, które spotykały się z nadużywaniem obecnie obowiązujących zapisów ustawy przez część przedsiębiorców, którzy nie prowadząc działalności zarządcy na rynku kolejowym, wykorzystywali przepisy do unikania opodatkowania. Problem, który przyczynił się do uszczuplenia wpływów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin, znany był rządowi od momentu wejścia w życie niefortunnych dla samorządu terytorialnego znowelizowanych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 1 stycznia 2017 r. Opieszałość Ministerstwa Infrastruktury postawiła gminy w Polsce przed koniecznością zwrotu nadpłaty podatku, o czym zresztą ministerstwo wiedziało z ustnych relacji przedstawicieli organizacji samorządowych działających w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a także zespołu ds. infrastruktury oraz rozwoju lokalnego i polityki regionalnej. Także w odpowiedzi na złożone przeze mnie zapytanie poselskie w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury otrzymałem informację potwierdzającą, że ministerstwo świetnie zdawało sobie sprawę z konsekwencji wprowadzonego w życie prawa, które w zasadzie ukarało samorząd terytorialny. Nad poprawką więc można było procedować przynajmniej rok wcześniej, w momencie, w którym ministerstwo opracowało rozwiązania, które problem ten eliminowały. Gminy, wielokrotnie zwracając uwagę na zaistniały problem, prosiły ministerstwo, jak i rząd o przeznaczenie pieniędzy na rekompensaty dla samorządów terytorialnych z tytułu stosowania zwolnień podatkowych w odniesieniu do gruntów, budynków i budowli infrastruktury kolejowej. Zmiany w przepisach okazały się niezwykle niebezpieczne dla budżetów gmin. W konsekwencji wiele z planowanych inwestycji nie zostało zrealizowanych lub ich realizacja uległa opóźnieniu. Przykładem w regionie jeleniogórsko-legnickim mogą być Osiecznica czy Nowogrodziec. Zwrot takiej kwoty dla tak małych gmin mógł mieć skrajnie niebezpieczne konsekwencje finansowe. Odpowiedzialność za ograniczenia możliwości finansowych samorządu nie pierwszy raz spada na obecny rząd, jednak w tym wypadku upływają prawie 4 lata od zaistnienia problemu do jego rozwiązania, co pokazuje niewydolność pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwestiach kluczowych dla wspierania i rozwoju samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę pozytywne opinie gmin w zakresie przepisów, które znalazły się w niniejszej ustawie, i konieczność jak najszybszego rozwiązania zaistniałej sytuacji prawnej, klub Lewicy będzie głosował za przedstawioną przez Ministerstwo Infrastruktury ustawą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę teraz pana posła Krzysztofa Paszyka o przedstawienie stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Bardzo dziękuję. Panie i Panowie Posłowie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści chciałbym przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Nie ukrywam, że analiza obu projektów skłania nas jako klub do tego, by to właśnie w projekcie senackim widzieć lepsze rozwiązania, lepiej dostosowane do sytuacji, która dzisiaj panuje.

Tak być nie powinno. Prawo dobre to powinno być prawo precyzyjne, które jest swoistego rodzaju panaceum na problem. A tu widzimy, znając fantazję i skłonności wielu podmiotów, że niestety dalej będzie swoistego rodzaju szara strefa, jeśli chodzi o wykorzystywanie terenów kolejowych do tego, aby prowadzić działalność i nie odprowadzać podatku od nieruchomości. Panie ministrze, prosty przykład.

Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła Artura Dziambora, który przedstawi stanowisko koła Konfederacja. Chciałem powiedzieć: Prawo i Sprawiedliwość, jak to typowo socjaliści, dzielnie naprawia błędy, które samo popełniło, czyli walczy z problemami, które samo stworzyło. W tym przypadku mamy kwestię podatku od nieruchomości, podatku lokalnego. Z oczywistych względów, gdy wprowadziliście takie prawo, które pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z pewnej ulgi, wiadomo było, że przedsiębiorcy dbający o to, żeby mieć jak najniższe koszty prowadzenia działalności - zresztą chwała im za to - będą robili wszystko, żeby z tej ulgi móc skorzystać.

Wasz rzecznik, pan poseł Fogiel, powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która zajmuje się regularnie obniżaniem podatków.

Nawet w samej tej ustawie, w jej analizie jest napisane jasno, że jedyni, którzy na tym stracą, to są przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje działalności gospodarcze na terenach objętych dotychczasowym wykluczeniem, a którzy nie prowadzą określonych działalności gospodarczych związanych z przeznaczeniem tych terenów. Takich przedsiębiorców są przecież tysiące. Tak właśnie, tymi maleńkimi kroczkami, maleńkimi podateczkami, które wprowadzacie albo podwyższacie, doprowadzacie do sytuacji, w której odechciewa się być przedsiębiorczym, odechciewa się prowadzić w Polsce firmy, odechciewa się tworzyć miejsca pracy. Jesteście po prostu - jak tutaj wielokrotnie można było zauważyć - ludźmi, którzy nie mają zielonego pojęcia o prowadzeniu jakiejkolwiek działalności. Są sprytniejsi od was, którzy potrafią odczytać różne dziwaczne prawa, które wprowadzacie, i chwała im za to, ja im naprawdę gratuluję i ich podziwiam. Natomiast wy zasadziliście się na tych ludzi i kombinujecie, co tu zrobić, żeby im było gorzej, i tutaj hańba wam, ponieważ wy powinniście dbać o to, żeby ludzie, którzy prowadzą swoje działalności, mieli jak najlżej w życiu. Powinniście dbać o to, żeby podatki były jak najniższe. W przypadku podatku od nieruchomości powinniście dbać o to, żeby on ewentualnie był lokalny, ale nigdy nie powinniście przeszkadzać w jakimkolwiek rozwoju. Niestety sytuacja jest inna. Smutne to, przykre to. Konfederacja będzie przeciwko temu. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pana posła Mirosława Suchonia o przedstawienie stanowiska Koła Parlamentarnego Polska 2050. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w łącznej dyskusji nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ujętym w druku nr 919 oraz rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ujętym w druku nr 1729. Wysoka Izbo! Przedstawione projekty ustaw wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zasadniczym celem przedstawionych projektów jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy w części dotyczącej zwolnienia z podatku od gruntów kolejowych. Zaproponowane rozwiązania likwidują lukę podatkową w zakresie podatku od nieruchomości, która skutkuje stosowaniem zwolnienia od podatku od nieruchomości w stosunku do podmiotów, które nie mają de facto nic wspólnego z działalnością w obszarze infrastruktury kolejowej poza faktem wykonywania działalności na gruntach kolejowych. Jest to oczywiście skutek ustawowego przedmiotowego zwolnienia od podatku działek zewidencjonowanych jako tereny kolejowe. Obecne brzmienie przepisów nie rozróżnia bowiem tego, czy na działce istnieją elementy infrastruktury kolejowej, czy też prowadzona jest inna działalność. Taka systematyka ma oczywiście negatywne konsekwencje. Po pierwsze, skutkuje uprzywilejowaniem części przedsiębiorców działających na gruntach kolejowych przez stosowanie zwolnienia od podatku od nieruchomości. To prowadzi do osiągnięcia niczym nieuzasadnionej przewagi konkurencyjnej nad tymi przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoją działalność na innych gruntach i normalnie opłacają podatek od nieruchomości. Po drugie, oznacza to również utratę części dochodów wspólnoty samorządowej, czyli mieszkańców tych miejscowości, w których położone są grunty zwolnione z podatku. Jak zauważył pan senator, suma tych zwolnień mogła osiągnąć już ponad 1 mld zł, czyli to są bardzo duże środki. Odnosząc się do obu projektów, należy zauważyć, że w zakresie doprecyzowania treści przepisu z art. 7 ust 1 projekty Senatu i rządu są podobne, natomiast projekt rządowy niejako rozszerza zwolnienie o te elementy infrastruktury, które służą świadczeniu usług związanych z obsługą podróżnych i o nieczynną infrastrukturę.

W imieniu Koła Parlamentarnego Polska 2050 wnoszę o przekazanie projektu do dalszych prac w komisji. Nie ma żadnego uzasadnienia tego, żeby takie grunty podlegały zwolnieniu. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o przedstawienie stanowiska pana posła Ryszarda Gallę. Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panie Ministrze!

Świadczy o tym także to, że Komisja Finansów Publicznych kilka miesięcy temu bardzo gorąco obradowała nad tym, w jakim zakresie mają być zapisane ustawowe zwolnienia z podatku tego typu nieruchomości. Zaistniał taki zbieg okoliczności, że samorządy kończą w tej chwili - czy też już skończyły - prace nad projektami budżetów.

W związku z tym każdy pieniądz, który jest po stronie dochodowej, jest bardzo istotny. Dobrze, że dzisiaj mamy dwa projekty: rządowy i senacki. Jeśli państwo pozwolicie, chciałbym skoncentrować się na kilku kwestiach. Panie ministrze, czy wiemy, jakie będą efekty tych zmian?

Bardzo dziękuję panu posłowi. Przystępujemy do tury pytań.

Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Bardzo dziękuję. Pytanie zada pan poseł Rafał Adamczyk. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pozwala ona na korzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przez podmioty, które nie prowadzą działalności na rynku kolejowym i wykorzystują nieprecyzyjny przepis do unikania opodatkowania. Rządowy projekt ustawy z druku nr 1729 został skierowany do konsultacji publicznych ze skróconym, 14-dniowym terminem przewidzianym na zgłaszanie uwag.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania pana posła Marka Rutkę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam pytanie o zasady dotyczące naliczania podatku od nieruchomości w przypadku bocznic kolejowych LHS, a więc tzw. linii hutniczej szerokotorowej o rozstawie szyn 1520 mm, tzw. rozstaw rosyjski, oraz pytanie dotyczące infrastruktury kolejowej znajdującej się w terminalu logistycznym Małaszewicze będącej częścią infrastruktury nowego jedwabnego szlaku. Dziękuję. Proszę teraz panią poseł Joannę Fabisiak, Koalicja Obywatelska. W moich pytaniach skoncentruję się na inwentaryzacji gruntów tzw. Kolejowych, wykorzystywanych na ten cel. Otóż jak wiadomo, tylko w części są one istotnie wykorzystywane, jak mówili przedmówcy, część to są tzw. rezerwy, często wieloletnie, właściwie będące nieużytkami.

Kolejne pytanie dotyczy tzw. rezerwy. Przedmówca także przed chwilą mówił o tym, że to są znów wieloletnie. Leżą, bo leżą, bo może kiedyś będą przydatne. Te tereny niewątpliwie należy zinwentaryzować, określić ich funkcje, a te, które nie są wykorzystywane, oddać samorządom. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zakłada, że bocznice kolejowe o statusie infrastruktury prywatnej, czyli prawie wszystkie bocznice kolejowe w Polsce, nie będą mogły uzyskać zwolnienia z podatku od nieruchomości. Może to w efekcie, panie ministrze, doprowadzić do takiej sytuacji, że użytkownicy bocznic zmienią status swojej infrastruktury na infrastrukturę nieczynną, bo infrastruktura nieczynna już podlega zwolnieniu. Przedstawione przepisy mogą obniżyć atrakcyjność utrzymywania setek bocznic kolejowych w Polsce. Pytanie, panie ministrze: Czy ministerstwo przeprowadziło analizy w tym zakresie i wie, jakiej liczby bocznic taka sytuacja może dotyczyć? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę teraz panią poseł Krystynę Skowrońską o zadanie pytania. Panie Senatorze! Panie i Panowie Posłowie! Po pierwsze, chciałabym zapytać pana ministra, czy zrobiono bilans gruntów, od których w tej chwili państwo nie płacicie podatku.

To jest rzecz niezwykle istotna. Druga rzecz dotyczy stanu niektórych nieruchomości, które stanowią własność kolei.

Myślę, że państwo powinniście się trochę pospieszyć z tymi deklaracjami, które składał premier akurat w Mielcu, a nie odwlekać włączenie budowy tego dworca do programu dworcowego. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Przedmiotem dzisiejszych prac są dwa projekty nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pierwszy z nich został złożony przez Senat rok temu, a drugi - przez rząd 5 dni temu. Tak się stanowi prawo? Rząd zapewnia, że uszczelnienie podatku od gruntów kolejowych zagwarantuje gminom dodatkowe pieniądze, więc dlaczego zwlekacie z uchwaleniem tego projektu. Z jednej strony mówicie o rekompensowaniu samorządom strat, które poniosły w związku ze zmianami wprowadzanymi w ciągu ostatnich lat dotyczącymi opodatkowania gruntów kolejowych, a z drugiej strony chcecie zabierać należne im pieniądze, działając w sposób opieszały.

Czy ten przepis zostanie doprecyzowany w trakcie procedowania? Chciałam zapytać, jakie przewiduje się rekompensaty dla jednostek samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję. Proszę teraz pana posła Szymona Pogodę o zadanie pytania. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Rządowy projekt ustawy uszczelnia, doprecyzowuje system zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku gruntów kolejowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem. Kilkukrotnie rozmawiałem z panem ministrem o tym problemie oraz o jego skutkach dla samorządów, dlatego, panie ministrze, dziękuję za ten projekt.

Jako poseł i zarazem mieszkaniec ziemi bolesławieckiej jestem żywo zainteresowany tym problemem, dlatego wierzę również, że termin wejście w życia tej ustawy z dniem 1 stycznia 2022 r. jest możliwy. Przekonuję kolegów i koleżanki z klubu o potrzebie zgłoszenia stosownych zmian. Dziękuję bardzo. Nie widzę. A zatem proszę pana posła Mateusza Bochenka. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W tym przypadku to niemal 95%.

Mnóstwo niezagospodarowanych obiektów, niszczejący dworzec PKP, niszczejąca wieża ciśnień, niszczejące, dzisiaj już niestety wyburzone koszary wojskowe, kilkadziesiąt kolejnych budynków - tak niestety wygląda ta rzeczywistość, w której miasto inwestuje, ponosi konkretne koszty, a PKP jako właściciel nie prowadzi absolutnie żadnych inwestycji (Dzwonek) Kiedy ta sytuacja się zmieni? Kiedy samorządy będą otrzymywały wsparcie finansowe, a właściciel weźmie odpowiedzialność za to, co czyni? Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Polskie samorządy od dawna czekają na zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na mocy której niestety powstała luka prawna i samorządy ponoszą straty finansowe ok. 200 mln zł rocznie. Podczas obrad komisji wspólnej rządu i samorządu pan minister obiecał, że nastąpi doprecyzowanie zapisów tej ustawy, tak żeby samorządy nie ponosiły strat finansowych. Tymczasem w projekcie ustawy znajdujemy wręcz rozszerzenie zakresu zwolnienia, które powiększy straty samorządów.

Dlaczego narażamy samorządy na dalsze straty, nieuzasadnione straty finansowe? Ta ustawa wymaga doprecyzowania. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Artura Łąckiego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie jestem zwolennikiem żadnej ustawy, która zwalnia z podatku jakiekolwiek działalności gospodarcze, nie patrząc na to, czy jest to kolej, czy jakaś inna. Chociaż ta ustawa przynajmniej jakieś pieniądze zostawia w kieszeniach samorządów, ale przecież pamiętamy ustawę o portach lotniczych, która z drugiej strony zabrała samorządom jeszcze większe pieniądze. Więc z jednej strony dajecie parę groszy, z drugiej strony zabieracie; wszystko się zgadza w kasie państwowej, oczywiście w samorządowej się nie zgadza. Ale jest jedna działalność, którą prowadzą i państwo, i samorządy, która moim zdaniem jest najważniejszą rzeczą dla społeczeństwa lub jedną z najważniejszych rzeczy. Szkoły są zwolnione z podatku od nieruchomości, jednostki wojskowe są zwolnione z podatku od nieruchomości - i bardzo dobrze, bo takie instytucje powinny być zwolnione - a szpitale nie są zwolnione z podatku od nieruchomości.

Czy to jest normalne czy to jest nienormalne, że kolej ma nie płacić, porty lotnicze nie będą płaciły, a szpitale muszą płacić podatki od nieruchomości? Prosiłbym rządzących o to, żeby się wreszcie nad tym zastanowili. Bardzo dziękuję. Pytanie zada pani poseł Marta Golbik. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana senatora, przedstawiciela wnioskodawców pierwszego projektu. Czy ma pan senator wiedzę, dlaczego aż rok ten projekt czekał? Z jakiego powodu przez rok samorządy musiały ponosić konsekwencje nieprzyjęcia tego projektu? Ale także interesuje mnie to, co na przyszłość. Jakie są szacowane straty związane z tym, że projekt nie wejdzie na początku 2022 r., tylko w roku kolejnym?

Jeśli mogę prosić, bo jest to ciekawa sprawa, o odniesienie się do tego. Bardzo dziękuję.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tereny kolejowe, tereny wyłączone stanowią bardzo często ogromny obszar, bardzo atrakcyjny gospodarczo, znajdujący się w centrum miast, miejscowości. Kwestia związana z możliwością opodatkowania tych terenów, uzyskania dodatkowych wpływów przez samorządy terytorialne, oczywiście mówimy o tych terenach, które nie służą wprost funkcjonowaniu kolei, jest jak najbardziej właściwa. Czy mogę państwa posłów prosić o wyciszenie rozmów? Bo przeszkadzamy koledze. Ale nie do pani poseł zawsze muszę się zwracać. Dziękuję, panie marszałku. Chodzi o doprecyzowanie tych terenów, które rzeczywiście służą działalności kolejowej, i tych, które nie służą. Dlatego że bardzo często właśnie na tych terenach znajdują się również galerie handlowe, punkty obsługowe i wyłączenie tych obszarów z możliwości pobierania podatku przez gminy jest nieuzasadnione. Chciałbym również zapytać, co stało u podstaw, że dopiero rok po wniesieniu projektu poselskiego, senackiego rząd zajął się tą sprawą? Straciliśmy rok. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Grzegorza Wojciechowskiego. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W gminach, gdzie są przystanki kolejowe, jest infrastruktura oczywiście, zawsze wokół dworca czy na samym dworcu rozwija się działalność, natomiast w gminach, gdzie linia kolejowa przebiega, ale ruch pasażerski został wyłączony albo też nie ma tam w ogóle przystanków, może być taka sytuacja, że infrastruktura, która mogłaby być wykorzystywana, nadal nie będzie wykorzystywana.

Proszę teraz pana posła Krzysztofa Grabczuka. Szanowny Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ma on dwa bardzo ważne elementy.

Pamiętajmy o tym, że to samorząd odpowiada za prawie 90% spraw codziennych (Dzwonek), którymi zajmuje się ludność. Bardzo dziękuję. Proszę teraz panią poseł Zofię Czernow. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Senatorze!

Przecież czas remontu lub modernizacji można określić. Do tej pory takie zwolnienia obejmowały 3-letnie okresy. Czyli te zwolnienia się rozszerza, a nie ogranicza, co tutaj błędnie było przekazane przez przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Chciałam zapytać: Dlaczego rząd tak hojną ręką oddaje pieniądze należne samorządom? Proszę dysponować swoimi pieniędzmi. Bardzo dziękuję, pani poseł. Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Mirosława Suchonia. Panie Ministrze! Panie Senatorze! Panie ministrze, mam pytanie dotyczące przepisu, na podstawie którego zamierzają państwo zwalniać z podatku od nieruchomości w przypadku zajęcia tej nieruchomości na cele związane bezpośrednio z obsługą podróżnych. Otóż zakładam, że tu chodzi o budynki stacji kolejowych. W tych budynkach często prowadzona jest różnego rodzaju działalność komercyjna, począwszy od zwykłych sklepików, które zaopatrują podróżnych, poprzez apteki i inne duże sklepy. Generalnie wiele dworców stało się niejako takimi minigaleriami handlowymi. Czy ten przepis będzie dotyczył zwolnienia od podatku również w przypadku, kiedy jest prowadzona działalność komercyjna? I drugie pytanie: Czy prowadzą państwo jakiekolwiek prace zmierzające do tego, żeby jednak nie likwidować bocznic kolejowych? Mówię tutaj w szczególności o Bielsku Podlaskim.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Artura Dziambora. Wysoka Izbo! Jeżeli wprowadza się jakiś dodatkowy podatek albo, tak jak tutaj niektórzy mówicie, uszczelnia się system, który już jest, to oczywiście zawsze wiąże się to z tym, że jest jakiś pieniążek do zarobienia.

Bardzo dziękuję. Na tym lista osób zapisanych do pytań została wyczerpana. Proszę teraz o ustosunkowanie się do nich pana Andrzeja Bittela, który jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za interesującą dyskusję, która dotyczy tego przedłożenia rządowego. Na początku chciałem powiedzieć, oczywiście nie jestem upoważniony do odnoszenia się do projektu senackiego, ale państwo pozwolą, że wyrażę taką opinię, że on jednak nie uszczelnia tej luki wynikającej z orzecznictwa sądów administracyjnych.

W mojej ocenie przepisy, które obowiązują, pozwalają spokojnie pobierać podatki od podmiotów, które nie prowadzą działalności kolejowej, nie udostępniają infrastruktury kolejowej.

Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że proces, w którym następuje łączenie działań po to, żeby dołączaną działkę zwolnić od opodatkowania, nie jest procesem naturalnym. Występuje z tym podmiot prowadzący działalność gospodarczą, organ ewidencyjny, starosta ten wniosek rozpatruje, dołącza. Skutkiem tego jest zwolnienie od opodatkowania, ponieważ ktoś posiada kawałek infrastruktury kolejowej, której na dodatek nie udostępnia. Jakby linia orzecznicza wzięła pod uwagę fakt udostępniania infrastruktury kolejowej, to takiego problemu w mojej ocenie by nie było. Ale skoro jest i linii orzeczniczej ani ja, ani Wysoki Sejm nie jesteśmy w stanie zmienić, to rzeczywiście trzeba podjąć interwencję i temu celowi służy ta ustawa.

Infrastruktura nieczynna to nie jest infrastruktura zlikwidowana, to jest infrastruktura, dla której nie jest prowadzony ruch pociągów, ale ona nie jest zlikwidowana. To jest ta różnica. Oczywiście czas modernizacji jest określony, bo jest umowa, są terminy.

Chciałem też powiedzieć - to jest odpowiedź na wiele wątpliwości czy pytań - że z całą pewnością w obecnym porządku prawnym i w tym projektowanym infrastruktura komercyjna, powierzchnie komercyjne, galerie handlowe, jak to państwo mówicie, powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Jeśli są one ogólnodostępne, powinny być zwolnione z opodatkowania, jeśli są bocznicami prywatnymi, nie wchodzą w zakres zwolnienia z opodatkowania.

Będzie porządek podatkowy. Ci podatnicy, którzy korzystali z luki wynikającej z orzecznictwa sądów administracyjnych, do czego nie mieli uprawnienia, i ich sąsiedzi z innych miejsc albo podlegający innym sądom administracyjnym właściwym miejscowo zachowają pewną równość wobec stosowania przepisów prawa. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Dziękuję za możliwość zabrania ponownie głosu. Najpierw odniosę się do tego, co najważniejsze w tym projekcie, i odpowiem na zadane pytania. Ja przypomnę tylko, że ustawa, która teraz musi być poprawiana, z 2016 r., co ciekawe, też 16 listopada przyjęta, weszła w życie od 1 stycznia 2017 r. Czyli na pewno się da. Mianowicie istnieje niedopuszczalna pomoc publiczna, nielegalna wręcz. W tej chwili istnieje pewna luka i prowadzi to do nieuczciwej konkurencji, dlatego że podmioty prowadzące działalność na obszarze kolejowym, które podlegają zwolnieniu z podatku od nieruchomości, konkurują z innymi podmiotami, które prowadzą swoją działalność bez tych zwolnień poza terenem kolejowym. Odpowiadając na pytanie, dlaczego ten projekt senacki czekał rok. Odpowiedź prawidłowa brzmi: nie wiem. Przy tym zwracam uwagę, że zdecydowana większość inicjatyw legislacyjnych Senatu tkwi w zamrażarce. Tam są równie ważne projekty jak ten, który teraz jest procedowany. To jest wręcz norma, szkodliwa norma, przy czym Senat wielokrotnie jest poganiany, kiedy dobrze proceduje, i to na czas, nad projektami sejmowymi. Nie ma tutaj żadnej współpracy, partnerstwa czy dbania o sprawy państwowe. Senacki projekt uszczelnia system podatkowy - chodzi o to, co nazywamy luką i o czym dyskutujemy. Zapis proponowany przez Senat jest praktycznie dokładnie taki sam jak zapis w projekcie rządowym, nie wiem więc, skąd to podejrzenie, że nie będzie skuteczny. Pan minister powiedział, że teraz jest możliwość pobierania podatku od tych podmiotów, o których mówimy, że unikają tego opodatkowania. No, te dwie rzeczy są sprzeczne. To, że nie jest ten podatek pobierany, wynika z interpretacji i orzecznictwa. Gdyby samorządy mogły go pobierać, na pewno by to robiły. Jeżeli zostanie wprowadzona ustawa senacka, na pewno będzie bez porównania łatwiej pobierać ten podatek, nawet jeżeli istnieją zagrożenia. Co do zwolnienia infrastruktury nieczynnej, zwracam uwagę, że chyba wszyscy wypowiadający się tutaj nie wnosili o zniesienie możliwości zwolnienia z tego opodatkowania, ale wnosili o to, aby to było zwolnienie czasowe, a nie bezterminowe. Zapis w ustawie proponowanej przez rząd dotyczy zwolnienia bezterminowego.

Bardzo proszę o podjęcie prac nad oboma projektami, wybranie z nich tego, co najlepsze, i o czas, czyli o takie procedowanie - będę o to zabiegał również w Senacie - aby ta ustawa likwidująca lukę podatkową mogła wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Odpowiadając na pytania o straty - każdy rok to jest co najmniej 200 mln zł straty. Ta strata to nie jest tylko ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego, to jest również patologia w działalności gospodarczej. Co więcej, ta strata narasta z roku na rok wskutek rozszerzania się tej, powiedziałbym, działalności kreatywnej przedsiębiorców, którzy np. scalają grunty po to, żeby uzyskać większe zwolnienie podatkowe. No, oczywiście to jest przesadne sformułowanie. Jeżeli wejdzie w życie ten projekt senacki.

Tak że o żadnym zahamowaniu rozwoju transportu kolejowego w Polsce przy tym senackim projekcie nie ma mowy. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zawarty w druku nr 1729, oraz senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zawarty w druku nr 919, do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Marszałek Sejmu proponuje, aby Sejm na podstawie art. 39 ust. 3 regulaminu Sejmu wyznaczył termin przedstawienia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (druki nr 1630 i 1708) Bardzo proszę pana posła Andrzeja Szlachtę o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Sejm na 39. posiedzeniu rozpatrzył i w dniu 14 października skierował rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok do Komisji Finansów Publicznych celem rozpatrzenia. Podczas omawiania przedmiotowego projektu ustawy zgłoszono siedem poprawek. Komisja te poprawki zaopiniowała pozytywnie.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Wiesław Janczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość dotyczące omawianego dokumentu, tj. projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej.

Wydaje się, że te wyjaśnienia, które strona rządowa przedłożyła w zakresie paramentów zapisanych w tym dokumencie. Parametry są dosyć istotne, bo przecież dotyczą zasad wynagrodzeń w sferze publicznej, m.in. dotyczą funkcjonowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczą Funduszu Pracy.

Można przywołać tutaj istotne dane i szczegóły, którymi się wówczas dzieliła i opozycja, i większość parlamentarna. One sprowadzają się do takich wielkości, które oddają obraz sytuacji, troski rządu o nauczanie, troski rządu o nauczycieli.

Przypomnę jeszcze, że nasz rząd wziął na siebie ciężar kosztów reformy administracji i likwidacji gimnazjów, co wiązało się ze znacznym rozproszeniem placówek.

Za chwilę zapewne pani zabierze głos w tej sprawie. Natomiast, proszę państwa, bardzo ważna też była obserwacja, którą pan minister oświaty w kontekście tej dyskusji przywołał. Ja osobiście zwracam zatem uwagę na taki szczegół, że ta duża grupa zawodowa, duża grupa branżowa, która jest liczona w setkach tysięcy osób - nie powiem, że to prawie 1 mln, ale to ok. 700 tys. osób - jest grupą zawodową, która została chyba jako kolejna trochę wystawiona, żeby nie powiedzieć: oszukana przez poprzedni rząd PO-PSL.

Ale potem już ten elektorat był mniej potrzebny, bo wiadomo było, że władza wymyka się z rąk, więc również o tej branży, jako jednej z nielicznych wcześniej zauważonych, zapomniano.

Do dalszego procedowania w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam jeszcze kolejne poprawki do tej ważnej ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa okołobudżetowa, zgodnie ze swoją potoczną nazwą, ma umożliwić realizację ustawy budżetowej. Realizowane jest to zasadniczo dwoma głównymi sposobami: albo poprzez mrożenie określonych środków, czyli utrzymywanie ich na określonym poziomie z jakiegoś okresu, w sytuacji gdy przepisy systemowe gwarantują przeliczanie środków np. według wzrostu wynagrodzeń z roku poprzedniego, albo poprzez finansowanie wydatków budżetowych środkami pochodzącymi z określonych funduszy celowych. Rozwiązania w ustawie okołobudżetowej obowiązują tylko w danym roku. Niestety rząd PiS już od kilku lat w ustawie okołobudżetowej praktycznie zawiesza ustawę o finansach publicznych. Przyjrzyjmy się niektórym szczegółowym rozwiązaniom, jakie rząd PiS proponuje w ustawie na rok 2022. Mimo zapewnień o świetnej kondycji budżetu ograniczone zostały środki np. na doskonalenie zawodowe nauczycieli, na doradztwo metodyczne, a także na nagrody, i to w czasie, kiedy szkoły borykają się z nauczaniem zdalnym, nauczaniem hybrydowym, kiedy uczniowie potrzebują wsparcia nauczycieli jak nigdy dotąd. W ustawie rząd zawiesza przepisy, które ograniczają środki na tworzenie rezerw. Uzasadnia to większą elastycznością, a tak naprawdę tworzy mętną wodę poprzez wykluczenie transparentności, bo tej transparentności, jeśli chodzi o wydatkowanie publicznych środków, PiS bardzo nie lubi.

W tej ustawie rząd właściwie likwiduje tzw. bezpłatne leki dla seniorów, bo te nieliczne, które były dla nich bezpłatne, mają być finansowane ze wspólnego worka NFZ-etu, czyli ze składki zdrowotnej podatników, w tym seniorów właśnie, której seniorzy już od podatku nie odliczą. Idźmy dalej, słynna Agencja Badań Medycznych. Jak podkreślał ówczesny minister zdrowia, ma ona służyć niekomercyjnym badaniom medycznym.

Fundusze celowe. Nie umiecie inwestować, nie potraficie przeprowadzić żadnej inwestycji od początku do końca, więc fundusze celowe, które mnożą się jak grzyby po deszczu, mają taryfę ulgową. Ich dysponenci mogą finansować nimi zupełnie inne inwestycje niż te, do których zostały powołane. Wtedy najłatwiej oszukiwać - poprzez budowę niejasnych, mętnych przepływów pieniędzy. Pieniądze w funduszach, przypomnę, są poza kontrolą parlamentarną, poza kontrolą opinii publicznej. Od kiedy rządzi PiS, powstało prawie 100 nowych funduszy, agencji, instytutów, do których PiS drukuje obligacje. Dziś ok. 350 mld zł jest poza kontrolą Sejmu, poza kontrolą budżetu. Tak jest też w wypadku Funduszu Szerokopasmowego - czy przypadkiem nie będzie nim zarządzał minister Cieszyński? - czy też CEPiK-u. Jedziemy dalej, minister obrony narodowej w roku 2022 r. będzie mógł właściwie wszystko. Dlaczego? Bo ministra obrony narodowej nie obowiązują prawie żadne reguły budżetowe. Dodatkowo bardzo szeroki strumień pieniędzy na obronę narodową z obligacji, czyli też z długu, został zagwarantowany w innej ustawie. Rząd PiS często chwali się zwiększeniem nakładów na badania, ale nie dodaje, że je też finansuje z długu. Podobnie fundusz reprywatyzacyjny, który dostaje już obligacje na obsługę obligacji. Zadłużycie nie tylko nasze dzieci, zadłużycie także nasze wnuki. No i prezydent, prezydent może dowolnie przenosić wydatki na obiekty zabytkowe. Wisienką na torcie jest Narodowy Instytut Wolności, któremu PiS zwiększa limit wydatków, żeby było jeszcze więcej na Bąkiewiczów, chociaż działalność Bąkiewicza ani nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, ani nie ma nic wspólnego z wolnością. Z interesem narodowym Polek i Polaków także nie ma nic wspólnego. Kończąc, pani marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej składam poprawki do rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej.

Dziękujemy bardzo, pani poseł. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Adrian Zandberg, Lewica. Wysoka Izbo! Miesiąc temu rozmawialiśmy tutaj w debacie łącznej o całym pakiecie ustaw budżetowych, i to było rozsądne, bo o technicznej w dużym stopniu ustawie, którą zajmujemy się dzisiaj, trudno rozmawiać na poważnie w oderwaniu od założeń, celów i priorytetów, które sobie postawiliście, a to niestety nie są dobre priorytety. Problem z całym tym pakietem można zamknąć w jednym zdaniu: oszczędzacie państwo nie tam, gdzie trzeba. Jeśli chodzi o dochody państwa, sytuacja nie jest zła, co przyznawał zresztą miesiąc temu rzadko widywany w tym budynku minister finansów. Ale wy tej szansy w tym pakiecie ustaw budżetowych po prostu nie wykorzystujecie. Za rozwojem gospodarczym musi w końcu pójść w Polsce rozwój społeczny.

A wy w tej ustawie dalej ograniczacie środki na edukację. Nie wiadomo, kto ma w przyszłości uczyć polskie dzieci informatyki, matematyki, języków. To jest realna sytuacja kryzysowa i odpowiedzią na ten kryzys powinien być budżet na przyszły rok, cały pakiet ustaw budżetowych. Ale prawica zachowuje się tak, jakby tego nie widziała. Niektórzy złośliwi mówią, że to dlatego, że panowie ministrowie posłali swoje dzieci do szkół prywatnych, tylko że to nie jest rozwiązanie systemowe, bo miliony Polek i Polaków będą wysyłać swoje dzieci do szkół publicznych. Jeśli dalej będziemy wydawać tak mało środków na edukację, to odbierzemy po prostu tym dzieciakom wiele, wiele szans. Czasem jednak niestety mam w tej Izbie smutne wrażenie, że po prawej stronie sceny politycznej nikogo to nie interesuje. Z podobnych powodów sypie nam się w Polsce budżetówka, bo przez lata było bardzo wdzięcznie szczuć na urzędników, wzywać, żeby im zaciskać pasa, i mamy dzisiaj efekty: specjalistów, którzy uciekają, rosnącą liczbę wakatów i niewydolne państwo. Niewiele. Prawda jest taka, że odrzuciliście skromne i naprawdę bardzo niewygórowane propozycje pracowników z OPZZ-etu, a w tym, co proponujecie, nie na nawet realnej osłony pracowników budżetówki przed rosnącymi kosztami życia. Fundusz płac ustawiliście tak, że rosnące koszty życia po prostu go pożrą, i to w ciągu kilku miesięcy. Ja mówiłem o tym miesiąc temu i powtórzę to dzisiaj: to jest naprawdę nie w porządku wobec ludzi, na których pracy stoi polskie państwo. Wreszcie najsłabsi.

Tym bardziej to jest moralnie nie w porządku, zwłaszcza teraz, kiedy będą rosły ceny żywności, kiedy będą rosły koszty życia i dla tych najbiedniejszych rodzin szykuje się ciężki czas.

Przypominam, że to tam właśnie pompujecie miliony złotych, które trafiają do fundamentalistów religijnych, na organizacje powiązane z panem Bąkiewiczem, do środowisk skrajnie prawicowych. To z tych pieniędzy wreszcie finansujecie w praktyce antyszczepionkowców, którzy potem paraliżują walkę z koronawirusem. I teraz bez żadnego sensownego uzasadnienia podnosicie skokowo ten budżet, tak naprawdę względem pierwotnego kształtu ustawy wielokrotnie.

I ktoś mógłby powiedzieć, że te dziesiątki milionów w skali budżetu to są drobniaki. Może tak, pewnie tak, ale niestety to jest symbol tego, jak dzisiaj wyglądają wasze priorytety. Te priorytety są po prostu nieakceptowalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska.

Zabierając głos w imieniu Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, chciałbym nawiązać do pewnej filozofii ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej. Właściwie ta ustawa otwiera boczne ścieżki nie do końca zgodne z zasadami budżetowymi, a na pewno narusza przejrzystość finansów publicznych i budżetu.

Główna uwaga jest taka, że poza kontrolą parlamentu pozostaje szereg obszarów finansowych, które są w bezpośredniej dyspozycji premiera czy ministrów.

Podobnie jest, jeśli chodzi o finansowanie niektórych obszarów w Agencji Badań Medycznych. Do szczegółowej analizy poszczególnych pozycji budżetu przystąpimy w przyszłości, po przeanalizowaniu i przyjęciu uwag, opinii poszczególnych komisji sejmowych, na poziomie Komisji Finansów Publicznych.

Sytuacja jest wyjątkowo złożona. Oczywiście wiemy, jak rośnie inflacja, jak jest ze stabilnością finansów.

Mówiłem też o tym, że duża część tych wydatków jest poza kontrolą parlamentu.

Już nie chcę nawiązywać do problemów związanych ze środkami unijnymi, które przecież są niezbędne dla realizacji naszego rozwoju. Na koniec chciałbym się odnieść do problemów związanych ze wzrostem cen, a więc do drożyzny, rosnącej inflacji.

Oczywiście są tu też czynniki obiektywne, związane z uwarunkowaniami zewnętrznymi, ze wzrostem cen surowców energetycznych, głównie paliw, gazu, ale są także działania, które są wynikiem pewnej niekonsekwencji rządu.

I bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wielce czcigodny towarzysz Adrian Zandberg powiedział przed chwilą, że biednych nie stać na lobbystów. I ma świętą rację, biednych nie stać na lobbystów i trzeba z tego wyciągnąć konsekwencje. Otóż np. miasto Houston w Teksasie przeznaczyło spore pieniądze na pomoc socjalną. Jak się okazało później, 80% tych pieniędzy poszło na budowę wieżowców dla wielkich firm. Bo wielkie firmy mają lobbystów, a biedni lobbystów nie mają. Dlatego też trzeba wszystkie pieniądze trzymać możliwie daleko od lobbystów, czyli trzymać poza rządem. Bo jeżeli trafią do rządu, to niewątpliwie lobbyści się tymi pieniędzmi zajmą i dla swoich klientów to załatwią. Rząd pieniądze wydaje gorzej, po prostu nie zna naszych potrzeb. Nawet gdyby nie kradł, co jest trudne, nawet gdyby nie był niedbały, nawet gdyby chciał jak najlepiej, to i tak nie zrobi tego, co nam jest potrzebne, ponieważ on naszych potrzeb nie zna.

Polska zbiedniała o 400 mln, bo pieniądze trafiły do rządu, zamiast być w kieszeni obywateli. Druga sprawa, bardzo niebezpieczna, to są zmiany.

Otóż niestety to, co widzimy w działalności rządu, to są nieustanne zmiany i poprawki.

Powiem jeszcze raz: jeżeli ludzie wydają swoje pieniądze, to je wydają na ogół rozsądnie i celowo, natomiast rząd te pieniądze na ogół marnuje. Na co marnuje, to ja nie będę mówił, bo koledzy z innych partii bardzo starannie pokazują to wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, Polska 2050.

Wysoka Izbo! Przedkładany projekt ustawy okołobudżetowej zawiera propozycje zarówno dobre, jak i kontrowersyjne. Koło Parlamentarne Polska 2050 z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w tym roku nie ma w niej mowy o zamrożeniu płac dla pracowników budżetówki. Praca wykonywana przez nauczycieli czy pielęgniarki zasługuje na godne zarobki, o które zawsze będziemy się upominać. Mam konkretne pytanie do rządu:

Więcej dostaną też służby mundurowe, choć uważamy, że dalsze zwiększenia tych wydatków powinny odbywać się pod kontrolą Sejmu, ale spod tej kontroli niestety ustawa te wydatki wyjmuje. Mamy nadzieję, że nie zapomnicie o sowitych podwyżkach dla cywilnych pracowników Policji, głównie kobiet, których płace są najniższe w sferze publicznej i nie pozwalają im na utrzymanie rodzin. To jawna dyskryminacja, która powinna się jak najszybciej skończyć. Nie rozumiemy jednak, czemu ta ustawa jest antyklimatyczna. W art. 41 wyłączacie regułę wydatkową, zgodnie z którą 18% z akcyzy od paliw silnikowych wspomagało rozwój kolei, a więc transportu publicznego. Likwidujecie ten zapis, co jest jawną abdykacją zielonych celów, bo teraz wszystko będzie szło na drogi. Tradycyjnie, jak co roku, nasz drogi pan prezydent staje się coraz droższy. Co więcej, kiedy w Polsce wzrasta skala skrajnego ubóstwa, wy wydajecie pieniądze na kolejne remonty rezydencji: Pałacu Prezydenckiego i Belwederu. W tym roku mieliśmy w ustawie okołobudżetowej ujęty remont ośrodka rządowego w Łańsku, gdzie z publicznych pieniędzy zakupiono samospłukujące się, nowoczesne toalety - w kraju, w którym według danych GUS 2 mln obywateli marzy, żeby posiadać w domu jakąkolwiek toaletę. Moglibyśmy cieszyć się, że społeczeństwo obywatelskie dostanie cztery razy więcej, gdyby nie fakt, że Narodowy Instytut Wolności, który zasilacie hojną kwotą 160 mln zł, jest silnie powiązany z osobami z Ordo Iuris i w niejasny sposób przekazuje pieniądze nacjonalistycznym, radykalnym ugrupowaniom, a drugą ręką pompuje środki w - a jakże - obywatelskie dzieła o. Rydzyka. A skoro jesteśmy już przy dziełach, to na Fundusz Kościelny w tym roku mieliśmy wydać 140 mln, wydaliśmy w 2021 r. 156 mln, a w następnym według tej ustawy wydamy prawie 193 mln. To o 36% więcej. Może proporcjonalnie o tyle właśnie ustalimy wzrost płac w budżetówce? Co rząd na taką propozycję?

Dziękuję bardzo, pani poseł. Jeżeli nie, zamykam listę. Jako pierwszy pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Bardzo proszę, panie pośle.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Podczas rozmów z wyborcami na temat tej ustawy każdy z nich formułował jeden wniosek, z którym nie sposób się nie zgodzić. Jeżeli do realizacji ustawy budżetowej potrzeba całego szeregu szczególnych rozwiązań, które wymagają formy ustawowej, to mamy do czynienia ze złym budżetem, niemożliwym do realizacji w warunkach prawnych, w których został on ustalony. Projekt ten jest przyznaniem się rządu do nierzetelnego przygotowania budżetu i przepchnięcia go przez Sejm dzięki posiadanej większości głosów z pełną świadomością, że jest on niewykonalny. Dlaczego rząd, mając pełną świadomość funkcjonujących ustawowych ograniczeń, przepycha przez Sejm kolejną ustawę, która jest niewykonalna? Dlaczego rząd stara się wstecznie dopasować realia prawne, aby dzięki takim zabiegom umożliwić realizację budżetu uchwalonego z naruszeniem obowiązujących przepisów? Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rządowy projekt ustawy z druku nr 1630 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 jest ściśle związany z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2022. W projekcie przewidziano możliwość przekazania przez ministra właściwego do spraw budżetu skarbowych papierów wartościowych dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna wartość zobowiązań z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty 4 mld zł. Panie Ministrze! Czym tak naprawdę spowodowana jest konieczność zwiększenia kapitałów będących w dyspozycji funduszu? Bardzo proszę o pisemną odpowiedź. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Wysoka Izbo! Rozpędzona inflacja, rekordowy wzrost cen, kryzys na granicy polsko-białoruskiej to sprawy, o których mówimy codziennie i którymi z pewnością zajmować się będziemy jeszcze bardzo długo. W związku z tym informacja o planowanych wydatkach na remonty prezydenckich rezydencji w Juracie, w Wiśle, w Klarysewie, w Promniku, Belwederu, Pałacu Prezydenckiego, opiewające na kwotę 25 mln, to chyba jakiś żart. Żeby tego było mało i premierowi nie było przykro, premierówka Stynka też przechodzi metamorfozę wartą 1600 tys. Kiedy pomyślicie w końcu o osobach z niepełnosprawnościami, o tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy? Czy będą pieniądze na kontynuację tego programu? Ile będzie tych środków? Kiedy zwiększycie dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych, do sprzętu rehabilitacyjnego? Na stronach i formach dla osób niepełnosprawnych w ostatnim czasie można przeczytać głównie o obawach dotyczących braku pieniędzy na leczenie (Dzwonek), na rehabilitację, na wózki, protezy, środki higieny, które z dnia na dzień drożeją.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pani poseł. Wysoka Izbo! Rozumiem, że waszą rolą przy rozpatrywaniu tego punktu jest uspokojenie nastrojów i zapewnienie obywateli, że ustawa ma ograniczyć wydatki budżetu państwa, ale wasze czyny w tej materii świadczą o czymś zgoła odmiennym. Fakty są takie, że regularnie zmniejszacie przejrzystość finansów państwa. Wypychanie przez was wydatków poza budżet przybrało niespotykaną dotąd skalę. Nie wykorzystywaliście dobrej koniunktury gospodarczej do oszczędzania, w efekcie czego szukacie pieniędzy, gdzie się da, nakładając kolejne podatki na obywateli. Polakom żyje się coraz trudniej. Mamy inflację najwyższą od 20 lat. To wszystko przy najmniejszej liczbie urodzeń od II wojny światowej i największej liczbie zgonów w powojennej historii Polski. Kiedy w końcu przedstawicie rzetelną i przejrzystą analizę i strategię prowadzenia polityki finansowej? Polacy mają prawo wiedzieć, czy finanse państwa są bezpieczne. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jedne podstawy są zamrażane, drugie są odmrażane i właściwie ma się wrażenie, że to wszystko ma tylko jeden cel: ukrycie inflacji.

Myślę o dzieciach. Galopująca inflacja i drożyzna powodują, że znów docierają do nas coraz liczniejsze sygnały o dzieciach po prostu głodnych, o rodzinach, które już sobie nie radzą, a co będzie od stycznia, jak będą wzrosty cen energii i gazu, trudno powiedzieć.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałem spytać, czy wielce czcigodny towarzysz Adrian Zandberg, który mówił o tym, że ministrowie swoje dzieci mają w szkołach prywatnych, a biedni to muszą posyłać do szkół państwowych. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z wybitnym przedstawicielem Lewicy w radiu i ten człowiek powiedział, zgodnie z prawdą zresztą, że bogaci to nie płacą podatków w gruncie rzeczy, unikają podatków, wielkie firmy unikają podatków, przede wszystkim podatki płacą biedni. No i dobrze. I on powiedział, że oczywiście edukacja nie może być prywatna, musi być finansowana z budżetu, z podatków, na co odpowiedziałem, że to znaczy, że biedni mają płacić na tę edukację, bo bogaci podobno podatków unikają. W radiu zapanowała minutowa cisza. Otóż, proszę państwa, trzeba by tak naprawdę skasować z podatków wszystkie pieniądze na edukację - to jest chyba, o ile pamiętam, 1300 zł na jedno dziecko miesięcznie - i dać te pieniądze rodzicom. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wydaje się, że dzisiaj. Inflacji, która zżera dochody, która powoduje, że ceny towarów, żywności, usług, nośników energii są coraz wyższe. I to zagraża bezpieczeństwu ekonomicznemu obywateli.

Dlaczego rząd nie chce pomóc obywatelom, panie ministrze? Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa o budżecie i ustawy okołobudżetowe to jedne z najważniejszych ustaw.

Rząd chwali się, że jest dobra sytuacja w budżecie. Tam wynagrodzenia są wyjątkowo niskie. Drugi gigantyczny dział, służba zdrowia. Zadłużenie szpitali za czasów PiS-u wzrosło o ok. 60%. Tysiące wakatów.

Zróbcie wszystko, żeby symbolem PiS-u nie były inflacja i drożyzna. Pani Marszałek!

Niewątpliwie w przyszłym roku będzie duża inflacja i niewątpliwie z tego tytułu do budżetu państwa wpłynie bardzo dużo środków. W związku z tym aż prosiłoby się, żeby zmniejszyć dług publiczny. Jeżeli przekroczymy budżet, a przekroczymy, to nie rozdawajmy tego np. na remonty instytucji państwowych, tylko spróbujmy ten dług zlikwidować czy zmniejszyć, ponieważ następne pokolenia będą go spłacać. Moje pytanie (Dzwonek): Czy rząd planuje zmniejszenie długu publicznego poprzez większy wpływ do budżetu państwa z powodu inflacji? Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Dyskusję o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 należy postrzegać w kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej Polski, a więc najwyższej od ponad 30 lat inflacji, szalejącej drożyzny. W tym sensie tworzenie budżetu na nowy rok powinno być oparte w jeszcze większym stopniu na dbałości o środki publiczne. Tymczasem co obserwujemy? Kolejną emisję obligacji. Miliardy obligacji, z których finansowane będą obronność czy badania naukowe. Widzimy tworzenie kolejnych funduszy, które poza kontrolą parlamentu będą wydatkowały miliony złotych. Za to widzimy liczne remonty rezydencji prezydenckich i rządowych. Nie tak powinien wyglądać budżet na rok 2022. Wysoka Izbo! Bez wątpienia sytuacja jest poważna i wymaga poważnych, bardzo odpowiedzialnych, racjonalnych decyzji.

Ten wzrost powinien nastąpić czym prędzej. Podobna sytuacja ma miejsce chociażby w przypadku pracowników cywilnych Policji. Przed kilkoma dniami spotkałem się z przedstawicielami tej grupy społecznej.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Czesław Siekierski, Koalicja Polska. Najlepszą inwestycją w nasz rozwój, w przyszłość, jest wspieranie obszaru edukacji. Samorządy muszą dokładać poważne kwoty do finansowania pensji nauczycieli, a to ogranicza realizację innych zobowiązań wobec mieszkańców. Sytuacja się zmieni, i to na gorsze, po wprowadzeniu rozwiązań podatkowych, które są w Polskim Ładzie. Ile trzeba będzie dokładać z budżetów samorządów na rzecz finansowania pensji nauczycieli? To jest jeden obszar. Mówimy o nauce, o innowacjach, nowych technologiach, badaniach.

Ostatnie pytanie, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Dlaczego będę mówiła? Dlatego że kosztowny jest dług. Kiedyś przyjdzie za to zapłacić. Przy niskich stopach procentowych to nie kosztuje tak wiele, ale zgodnie z założeniami Narodowego Banku Polskiego będzie to coraz droższe. To jest pierwszy wyrzut sumienia - drogość. Drugi. Przed kancelarią premiera od września trwa strajk pracowników ochrony zdrowia.

Brak rekompensat za prąd.

To jest test na szacunek dla obywateli. Dziękuję bardzo, pani poseł. To było ostatnie pytanie. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów pana ministra Sebastiana Skuzę o odpowiedzi na pytania.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa okołobudżetowa stanowi szczególne rozwiązanie i jest elementem powszechnie obowiązującego prawa, gdyż ma formę ustawy, czyli źródła prawa konstytucyjnego.

Pojawiały się pytania o pakiet dla osób niepełnosprawnych. Przypomnę, że omawiając tutaj nowelizację ustawy budżetowej na rok 2021, mówiłem o 1 mld zł dla osób z niepełnosprawnościami jeszcze w tym roku.

W zakresie transparentności finansów publicznych obowiązują nas przepisy unijne i zestawienie całego sektora finansów publicznych, również funduszy, które są umiejscowione w Banku Gospodarstwa Krajowego, jako tzw. sektor general government. Pojawiały się również pytania dotyczące inflacji. Polityka pieniężna to głównie narzędzia Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego.

Jakie narzędzia powinny być wprowadzone do walki z inflacją w ustawie okołobudżetowej?

Pojawiało się również pytanie o system oświaty. Uważam, że w naszym kraju jest miejsce zarówno dla publicznej, jak i dla prywatnej oświaty.

Również przypominam o utworzeniu jeszcze w tym roku, z możliwością wykorzystania w roku przyszłym, 6-procentowego funduszu motywacyjnego. Jeżeli chodzi o służby MSWiA, to kierownictwo podpisało porozumienie ze związkami zawodowymi. Ma być kontynuowany program modernizacji służb mundurowych, w tym również w obszarze wynagrodzeń. Co do państwowego długu publicznego, to strategia zarządzania długiem zakłada spadek tego długu w relacji do produktu krajowego brutto. W latach 90. obligacje Skarbu Państwa były wykorzystywane do restrukturyzacji sektora bankowego. W latach dwutysięcznych, od 2009 r. obligacjami może być dokapitalizowany Bank Gospodarstwa Krajowego, co jest kontynuowane. A jeżeli chodzi o sektor nauki i szkolnictwa wyższego, wprowadzenie takiej możliwości dokapitalizowania obligacjami zostało bardzo dobrze przyjęte przez sektor uczelni. Chciałbym zauważyć, że środki, o których jest mowa w ustawie okołobudżetowej, w obligacjach dla jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego to jest, można powiedzieć, coś dodatkowego, gdyż z algorytmu opartego na inflacji i produkcie krajowym brutto wynika jakaś minimalna kwota dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, a obligacje nie wchodzą w tę kwotę, czyli są czymś jeszcze ponad ten minimalny wymóg.

Padło również pytanie o kwestie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Chciałbym zwrócić uwagę, że po trzech kwartałach tego roku nadwyżka operacyjna, czyli dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, w sektorze samorządu wynosi ponad 30 mld i jest rekordowa, a jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymały jeszcze, czyli w tej kwocie nie jest to uwzględniane, 8 mld z tytułu subwencji rekompensującej i 4 mld z tytułu subwencji na kwestie związane z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Tu padło pytanie, właściwie stwierdzenie, że 2 mln Polaków chciało... ich marzeniem jest posiadanie łazienki. Zauważam, że 4 mld zł jeszcze w tym roku zostanie przekazane do jednostek samorządu terytorialnego, w których nasycenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną jest najniższe.

W zakresie leków i ich finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia chciałbym zauważyć, że taka operacja miała już miejsce i absolutnie nie ma tu jakiejkolwiek likwidacji przywilejów. To jest tylko zmiana w finansowaniu organizacyjnym. Wzrost nakładów na służbę zdrowia w przyszłym roku jest zauważalny.

Bardzo proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Andrzeja Szlachtę.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! My w tej chwili omawiamy rządowy projekt ustawy okołobudżetowej, a nie dyskutujemy o budżecie państwa. Chciałem mimo wszystko podziękować członkom Komisji Finansów Publicznych, którzy przy tym projekcie pracowali kilka godzin. To była w większości debata merytoryczna, troska o budżet polskiego państwa, o wydatki, ale sytuacja została stworzona przecież nie przez władze, ale przez zjawiska zewnętrzne, takie jak pandemia, skutki pandemii, sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie. Jesteśmy krajem, który żyje w warunkach polityki globalnej, i zjawiska inflacyjne nie są ewenementem tylko polskim.

Proszę państwa, no nie siejmy paniki. Każda ustawa, tak jak pan minister powiedział, ma charakter konstytucyjny i ustawy, które Sejm przyjmuje, są realizowane.

To jest rzecz normalna.

To są setki miliardów złotych kierowane do polskich rodzin, do dzieci.

Jeżeli chodzi natomiast o subwencję, to porównajmy dochody kierowane. Pani ma taką manierę przeszkadzania zawsze i w każdym miejscu. Proszę nad tym panować.

Proszę państwa, 13 mld zł na subwencję.

Dziękuję bardzo. Chciałabym też przypomnieć, że jest pan sprawozdawcą komisji.

Wysoka Izbo!

Wedle tych danych rośnie stopa ubóstwa, w tym rośną także ubóstwo rodzin i bieda dzieci. Wobec powyższego, wobec danych GUS-u, spytałam tylko o to, jakie są środki zaradcze, bo dalej tego procederu nie możemy przecież utrzymywać ani akceptować. Dziękuję bardzo. Pani poseł Krystyna Skowrońska. Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Szanowny Panie Pośle Sprawozdawco! Jakoś trudno wytrzymać, jeżeli państwo opowiadacie rzeczy nieprawdziwe.

Niestety, panie ministrze, pan również mnie źle zrozumiał. Jest pan znany z bardzo dużej dokładności, szanuję ją, ale jednak pomimo wszystko leki dla osób starszych państwo wyrzucacie z budżetu. Już drugi raz niesławetne 75+ jest wyrzucone. My będziemy płacić, bo Narodowy Fundusz Zdrowia to są nasze pieniądze, które pracujący Polacy wpłacili.

Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druki nr 1672 i 1745) Bardzo proszę panią poseł Danutę Nowicką o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, druki nr 1672 i 1745. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 21 października 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania.

Celem omawianej regulacji jest rozszerzenie katalogu przesłanek zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy z odpłatności za jego pobyt w tym domu i wynika ze społecznej potrzeby zagwarantowania większej ochrony członkom rodzin pensjonariuszy tych instytucji. Projekt ma na celu wyeliminowanie poczucia niesprawiedliwości w stosunku do członków rodzin osób, które w sposób rażący nie wywiązywały się z obowiązków rodzicielskich.

Izby o przyjęcie ustawy zgodnie z drukiem nr 1672. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, druki nr 1672 oraz 1745. Wysoka Izbo!

Celem projektowanej regulacji jest rozszerzenie katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodzin mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w tym domu. O wprowadzenie zmian w zakresie rozszerzenia katalogu przesłanek umożliwiających zwolnienie członków rodziny mieszkańca DPS-u z odpłatności za jego pobyt postulował m.in. rzecznik praw obywatelskich.

uwzględniając wyjątkowe okoliczności, odstąpić od ustalenia opłaty. Problem będący przedmiotem projektowanej regulacji sygnalizowali również rzecznik praw dziecka oraz sami pracownicy DPS-u za pośrednictwem Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Zwrócili oni uwagę na zaporowe warunki, jakie muszą wypełnić dorosłe dzieci, ofiary wcześniejszych nadużyć ze strony rodziców, by nie były zobowiązane do pokrywania kosztów związanych z pobytem rodziców w domu pomocy społecznej. Skierowali oni postulaty, by instytucja zwolnienia z odpłatności objęła również przypadki dotyczące postępowań rodziców określonych mianem sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, które to pojęcie na gruncie prawa posiada również swoje precyzyjne odniesienie i interpretacje.

Obecne przepisy pomijają kwestię braku więzi rodzinnych między osobą zobowiązaną do ponoszenia opłaty a pensjonariuszem domu pomocy społecznej.

Wysoka Izbo! Mając na uwadze powyższe, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o przyjęcie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu komisji z druku nr 1745. Bardzo proszę, pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicja Obywatelska w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, druki nr 1672 i 1745. Celem projektowanej regulacji jest zagwarantowanie większej ochrony rodzinom, których osoby spokrewnione przebywają w domach pomocy społecznej, poprzez rozszerzenie katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia rodzin tych mieszkańców DPS-ów z odpłatności za ich pobyt w jednostkach pomocy społecznej. Zgodnie z aktualnymi przepisami w pierwszej kolejności za pobyt w DPS-ie powinien zapłacić sam mieszkaniec. Jeżeli nie jest to możliwe, to odpłatność ponosi małżonek, spokrewnieni zstępni przed wstępnymi, a jeżeli nie ma krewnych lub nie można wyegzekwować od nich należnych środków, pobyt opłaca gmina, z której osoba została skierowana do DPS-u. O zwolnieniu z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej stanowi art. 64 ustawy o pomocy społecznej. W artykule tym wskazano, iż zwolniona z odpłatności może być osoba, która przebywała w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do DPS-u lub mieszkańcowi domu. Zmiany te wprowadzone kilka lat temu są jak najbardziej sprawiedliwe i w praktyce się sprawdzają. Jednak jak wynika z uzasadnienia, a także z konsultacji, które przeprowadziłam z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej oraz przedstawicielami domów pomocy społecznej, problem pojawia się w sytuacji, gdy rodzic nie został w odpowiednim czasie pozbawiony praw rodzicielskich. Dzieje się tak wtedy, gdy w najtrudniejszym momencie braku opieki i realizowania podstawowych potrzeb dziecka drugi z rodziców czy opiekun, który sam doświadcza przemocy, chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa dzieciom, nie doprowadzi do końca procedury pozbawienia praw rodzicielskich, nie dopilnuje tego. Tym samym nie otrzyma prawomocnego orzeczenia o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Na domiar złego zdarza się, że drugi z rodziców nie żyje, co w praktyce eliminuje możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej jedynego opiekuna dopuszczającego się nadużyć. Środowisko pomocy społecznej jest zgodne co do tego, że właśnie te kwestie należy doprecyzować, tak aby instytucja zwolnienia z odpłatności objęła również przypadki postępowań rodziców określone mianem sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Wprowadzenie do ustawy o pomocy społecznej wyraźnej regulacji prawnej umożliwiającej właściwemu organowi odstąpienie od obciążania odpłatnością za pobyt w domu pomocy społecznej jest oczekiwane i uzasadnione. W projekcie, nad którym dzisiaj procedujemy, przewidziano możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt mieszkańca DPS-u osoby, wobec której pensjonariusz ten w przeszłości rażąco zaniedbywał obowiązki rodzicielskie, doprowadzając do ustania więzi rodzinnych, oraz gdy było to rażące naruszenie przez pensjonariusza obowiązku alimentacyjnego względem dziecka lub zaniedbywanie innych obowiązków rodzinnych, np. obowiązku opieki, wychowania czy utrzymania.

Na dorosłych dzieciach spoczywa obowiązek troski o rodziców. Dla wielu z nas jest to oczywiste i nie wyobrażamy sobie, aby mogło być inaczej. Jednak zasada ta nie może być wykorzystywana i nadużywana przez osoby, które jedynie formalnie są rodzicami, a w rzeczywistości nigdy nie zajmowały się swoimi dziećmi i nie były finansowo zaangażowane w ich utrzymanie. Często słyszy się o przypadkach dorosłych już dzieci, które po kilkudziesięciu latach dowiadują się, że ojciec, który był przemocowcem, lub matka, która porzuciła dzieci, przypomnieli sobie o ich istnieniu i wymagana jest od nich alimentacja za ich pobyt w placówce pomocy społecznej. Myślę, że wielu z nas zna różne historie, chociażby taką jak ta opisana przez pewną kobietę. Dostałam odpowiedź z SKO o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji o odpłatności za ojca, który przebywał w DPS-ie. Nie wiem, co powinnam teraz zrobić. Jakiś czas temu dostałam decyzję z OPS-u o konieczności wnoszenia opłat, od której się odwołałam. W międzyczasie ojciec zmarł. Nie płacił alimentów. Byłam w rodzinie zastępczej, ale przez to, że mama chorowała na schizofrenię, nie była w stanie pozbawić go praw rodzicielskich. SKO twierdzi, że nie mają znaczenia negatywne więzi emocjonalne z ojcem, a strona ma obowiązek prawny uiszczać opłatę. Ponadto napisano, że postępowanie w sprawie zwolnienia może być wszczęte dopiero, gdy decyzja ustalająca wysokość opłaty stanie się ostateczna. Nie mam pojęcia, co mam w tej sytuacji zrobić. Takie sprawy to ludzkie dramaty i powrót myślami do traumatycznych przeżyć z okresu dzieciństwa. Dlatego zgodnie z nowymi przepisami dorosłe dzieci osób, które w społecznie nieakceptowalny sposób podchodziły do rodzicielstwa, powinny zostać zwolnione z opłaty bez względu na to, w jakiej sytuacji finansowej się znajdują. Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni (Dzwonek) będzie głosował za proponowanymi zmianami w ustawie o pomocy społecznej. Mamy jednak wątpliwości dotyczące kwestii weryfikacji składanych wniosków, panie ministrze. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy przygotowany przez rząd uwzględnia wiele sygnałów i wystąpień rzecznika praw obywatelskich i rzecznika praw dziecka. Jest też wynikiem analizy orzeczeń sądów, orzeczeń instytucji w procesie postępowania o wydanie decyzji administracyjnych. Uwzględnia również opinię wyrażoną już wtedy, kiedy trafił do parlamentu, do Biura Analiz Sejmowych. Celem projektowanej regulacji jest rozszerzenie katalogu przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt. Dzisiejsze regulacje, zwłaszcza art. 64a ustawy o pomocy społecznej, wskazują, że osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona, albo jest prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej małoletniego rodzeństwa lub rodzica. Te rozwiązania jednak nie wytrzymały próby czasu. Są sytuacje, z którymi mamy często do czynienia również w naszych biurach poselskich, są prośby o interwencję. Jednak bez tej interwencji prawnej, którą przygotował rząd, trudno byłoby wyjść naprzeciw tymże oczekiwaniom. Dlatego też Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy będzie popierał te rozwiązania, które przewidują oprócz przesłanek fakultatywnych również obligatoryjne. Jeśli chodzi o wyłączenie z obowiązku opłacania przez dzieci, rodzinę pobytu rodziców wtedy, kiedy naruszane są zasady współżycia społecznego, zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny czy wychowanie dzieci, jest to w pełni uzasadnione. Jest także ta przesłanka mogąca wyłączyć obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt pensjonariusza w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do opłaty wykaże na podstawie tych dokumentów rażące naruszenie przez osobę kierowaną do DPS-u lub mieszkańca DPS-u obowiązku alimentacyjnego, obowiązku wnoszenia opłaty, obowiązku związanego z wychowaniem i utrzymaniem, dbałością o rozwój intelektualny swojego dziecka. Wszystkie te rozwiązania uszczelniają, można powiedzieć, tę kwestię wzajemnych relacji.

Konkludując, chciałbym poinformować, że klub udziela wsparcia temu projektowi, będzie głosował za przyjęciem zmiany ustawy o pomocy społecznej zawartej w druku nr 1672. Dziękuję.

Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów mam przyjemność przedstawić państwu stanowisko klubu dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z druku nr 1672. Często w naszej pracy, wcześniej społecznej, a teraz poselskiej, spotykamy się z problemami społecznymi, z problemami rodzinnymi. Niejednokrotnie, jak sami państwo wiecie, są to dramaty ludzkie.

Tak, ta ustawa, choć nie jest doskonała, pozwoli rozwiązać szereg takich problemów. W uzasadnieniu ustawy nowelizującej wskazano, że wprowadzenie nowej regulacji w art. 64 ma na celu przeciwdziałanie poczuciu niesprawiedliwości w stosunku do dzieci zobowiązanych do ponoszenia odpłatności w domu pomocy społecznej za pobyt rodzica, wobec którego zostało wydane orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej. W nowelizacji ten katalog został rozszerzony o następne dwie przesłanki. W tej kwestii niejednokrotnie zabierał również głos rzecznik praw obywatelskich, w którego ocenie dorosłe dzieci rodziców, którzy względem nich w sposób rażący zaniedbywali obowiązki rodzicielskie lub byli sprawcami przemocy wobec dziecka, zasługują na ochronę państwa i powinny zostać objęte obligatoryjnym zwolnieniem z opłat bez względu na ich sytuację materialną. Omawiany problem był również przedmiotem analiz rzecznika praw dziecka. W ocenie rzecznika praw dziecka prawo powinno chronić dorosłe dzieci rodziców w przypadku braku wykonywania przez tych rodziców obowiązków rodzicielskich czy popełniania na szkodę małoletnich dzieci przestępstw.

Dotychczas dorosłe dziecko mogło zostać zwolnione z takich opłat tylko pod warunkiem, że rodzic był pozbawiony praw rodzicielskich wyrokiem sądu. Nowelizacja proponuje dodanie nowych przesłanek mogących wyłączyć obowiązek ponoszenia opłaty za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej, tj. sytuację, w której osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku rażące naruszenie przez osobę kierowaną do DPS-u lub mieszkańca domu pomocy społecznej obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty. Tutaj nasuwa się pytanie, jakie to mają być dokumenty, bo nowela wyraźnie tego nie wskazuje, i czy ich weryfikacja przez pracowników domu pomocy społecznej będzie wystarczająca i rzetelna. W wielu przypadkach, jeżeli zostaną uznane powyższe przesłanki i rodzina nie zechce łożyć na pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej, ten obowiązek będzie spoczywał, jak wiemy, na barkach samorządu. Mam zatem pytanie do strony rządowej: Czy samorządy będą mogły liczyć na rekompensatę w tym zakresie? Klub Koalicji Polskiej - Polskiego Stronnictwa Ludowego, Unii Europejskich Demokratów i Konserwatystów poprze rozwiązania zawarte w nowelizacji tej ustawy.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przede wszystkim chciałbym wyrazić pewne zdziwienie, że w dyskusji nad rzeczą bardzo skomplikowaną, jaką jest budżet, mieliśmy po 3 minuty, a w dyskusji nad drobną poprawką do jednej ustawy mamy po 5 minut. Po drugie, chciałem zwrócić uwagę, że to nie jest dyskusja o pomocy społecznej, tylko o pomocy państwowej. Zbieramy pod przymusem podatki i te pieniądze są potem rozdawane. Powinien to być dom pomocy państwowej, a nie dom pomocy społecznej. Po trzecie, doskonale rozumiemy, że urzędnicy państwowi chcieliby zrobić jak najlepiej. Obecna sytuacja prawna jest zła i po tym jest trochę lepsza być może. Natomiast chciałbym zwrócić uprzejmie uwagę, że są dwa podstawowe zastrzeżenia do tej ustawy. Pierwsze jest takie, że ona jest oczywiście nieprecyzyjna i będą dalej dyskusje, czy rzeczywiście są dostateczne przesłanki, czy nie. O wiele prościej byłoby powiedzieć po prostu: niech sąd to ustali, czy jest słuszne, żeby płacić, czy nie, i to by było o wiele prościej, nie byłoby długiej ustawy, tylko byśmy to powierzyli sędziemu, który robi to na miejscu, w gminie czy w powiecie. I to jest znacznie lepsze rozwiązanie.

Takie rzeczy niestety będą bardzo powszechne, chcę o tym ostrzec ustawodawców, którzy potem chcą jak najlepiej.

To jest złe w ogóle podejście do rzeczy, ale rozumiem, że na inne podejście nas nie stać, bo mamy prawo rzymskie, a nie prawo angielskie, w związku z czym musimy dawać dużo prawnych wytycznych, wskazówek sędziemu, żeby wiedział, jaką podjąć decyzję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Joanna Mucha, Polska 2050.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! W pierwszych słowach od razu powiem, że oczywiście zagłosujemy za tą ustawą, bo to jest ustawa, która przywraca trochę elementarną sprawiedliwość społeczną. Oczywiście rozmawiamy dzisiaj o ustawie, która dotyczy wyłącznie dramatów ludzkich, i to dramatów, naprawdę, których pewnie nie chcielibyśmy rozstrzygać. Nie chcę powtarzać argumentacji, która tutaj już padała, bo oczywiście wszyscy wiemy, że to jest ustawa o rozszerzeniu katalogu przesłanek obligatoryjnego lub fakultatywnego zwolnienia z opłat za pobyt w DPS-ach, to jest główna treść tej ustawy, i że oczywiście tego typu rozstrzygnięcie prawne było potrzebne i było oczekiwane. Każda z tych sytuacji, czy to jest zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czy to jest brak więzi społecznych, czy to jest rażące zaniedbanie obowiązków rodzicielskich, czy nawet brak alimentacji - to zawsze jest jakieś kontinuum. Bo przecież i brak alimentacji może być czasowy, może być tak, że alimenty wpływają tylko częściowo, nie w pełnej kwocie. Więc za każdym razem albo bardzo często mamy do czynienia nie z zerojedynkowymi sytuacjami, tylko z sytuacjami, które są ocenne. Z tego powodu mój apel do pana ministra, żeby spróbować jednak w jakiś sposób ułatwić sytuację osób, które będą musiały dokonywać oceny, i by jak najbardziej zbliżyć tę ustawę czy może przepisy z nią powiązane, do tego, żeby jak najbardziej ułatwić pracownikom ocenę, weryfikację np. właśnie poprzez dokładne określenie, jakiego typu dokumenty mogą być brane pod uwagę, bo tego trochę brakuje w tej ustawie. Brakuje też przepisów przejściowych, na co chciałabym zwrócić uwagę. Więc, tak jak w innych okolicznościach istnieje coś takiego jak katalog dobrych praktyk, tak tutaj możemy pomyśleć o jakimś katalogu interpretacyjnym, który będzie pomagał w ocenie każdej tego typu sytuacji. Bo tak jak mówię, tak jak rozpoczęłam moją wypowiedź - my tu za każdym razem będziemy mieli do czynienia z sytuacją jakiegoś dramatu, dramatu rodziny lub części tej rodziny. Obciążeni tą sytuacją będą pracownicy, którzy będą musieli podejmować decyzje. W ostatnich słowach apel o to, żeby środki, które nie wpłyną w ten sposób do samorządów, zostały (Dzwonek) uzupełnione przez rząd. Dziękuję bardzo. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oczywiście, panie ministrze, kierunek słuszny: niweluje pewną niesprawiedliwość społeczną, o której wszyscy przedmówcy tutaj mówili. Jeżeli ktoś jest dorosłą osobą, a w życiu musiał sobie poradzić sam, bo jego rodzice nie wywiązywali się z obowiązków, to jest bardzo sprawiedliwe, że w takim wypadku nie będzie ponosić kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej.

Oczywiście ta sprawa w wielu ośrodkach pomocy społecznej bardzo często spędza sen z powiek pracownikom socjalnym, którzy pracując w swoim środowisku, znają rodziny od podstaw i wiedzą, że muszą wydać decyzje - czy dyrektorzy, czy kierownicy - które są po prostu niesprawiedliwe wobec ludzi, którzy nie mieli kontaktu ze swoimi rodzicami przez wiele lat, ale nie mają dowodów prawnych w postaci wyroku i to nie jest ich wina, ponieważ o te wyroki musiałaby zadbać druga strona, czyli drugi rodzic albo w jakiś sposób ktoś inny, kto sprawował opiekę, ale tak się nie działo. Chcę tylko nawiązać do tego, że to jest kolejna zmiana ustawy o pomocy społecznej. Takich sytuacji będziemy mieć wiele, gdzie trzeba będzie ją poprawiać w różnych elementach, dlatego że zmienia się struktura społeczna, struktura problemów społecznych i światowe podejście do rozwiązywania problemów rodziny, bo osoba nigdy nie jest sama, tylko istnieje w rodzinie, na zasadach bardzo holistycznego podejścia. Warto, żeby przeprowadzić poważną reformę pomocy społecznej właśnie w takim kierunku, aby wykorzystać już bardzo dobrze zgromadzony potencjał pracowników socjalnych, dobrze wykształconych, dobrze przygotowanych, ponieważ przez lata stawiano im wysokie wymagania, aby trochę zdać się na zindywidualizowane podejście, czyli żeby pracownik socjalny, nie sąd, tak jak mówił tu mój przedmówca pan Korwin-Mikke, tylko pracownik socjalny, wysokiej klasy specjalista mógł razem z rodziną opracować plan pomocy dotyczącej wyjścia z kryzysu. To jest naprawdę poważna zmiana systemowa, ale myślę, że trzeba jej dokonać. A druga moja sugestia i prośba, od paru lat składana właśnie do pana ministra sprawiedliwości, w przypadku której wielokrotnie się zobowiązywał, po części powiązana z tym problemem, z którym mamy do czynienia, dotyczy pracy nad zmianą instytucji ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie, dlatego że nadal ta instytucja jest bardzo nadużywana. Dwukrotnie składałam projekt poparty przez wiele organizacji pozarządowych i dwukrotnie słyszałam od ministra sprawiedliwości, że projekt być może miał wady prawne, powinien znaleźć się w komisji kodyfikacyjnej i Prawo i Sprawiedliwość taki poprawny prawnie projekt przygotuje. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zgłosić się do zadania pytania? Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ta regulacja ustawowa rozszerza katalog przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w domu pomocy społecznej. Rzeczywiście rozwiązuje i reguluje niesprawiedliwość społeczną, która do tej pory w sprawie tej odpłatności była. Natomiast mam takie pytanie. Ustawa przewiduje, że wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. A pytanie jest takie: Czy zaproponowany termin wejścia w życie ustawy jest wystarczający z punktu widzenia możliwości przygotowania się adresatów norm, których dotyczą projektowane przepisy? Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Wysoka Izbo! Mówimy dzisiaj o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Projekt rozszerza katalog przesłanek obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia członków rodziny mieszkańca domu pomocy społecznej z odpłatności za jego pobyt w tym domu. Czy w związku z rozszerzeniem i zwiększeniem wsparcia dla osób potrzebujących Skarb Państwa przekaże większe środki do samorządów lokalnych na wspieranie obywateli? Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! I kolejne pytania, panie ministrze. Moje wątpliwości budzą rozwiązania związane z wejściem procedowanych przepisów w życie i objęciem tą regulacją spraw zakończonych. Art. 2 stanowi, że regulacja będzie miała zastosowane do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy. Wprowadza to nierówność prawną osób, których obowiązki zostały już uregulowane dotychczasowymi przepisami. Istnieje zagrożenie, że sytuacja osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS-ie do chwili wejścia w życie nowelizacji pozostanie niezmienna i nie będą oni mogli skorzystać z regulacji korzystniejszych. I pytanie: Czy nowa regulacja będzie podstawą do wszczęcia postępowania dotyczącego zwolnienia rodziny z odpłatności w przypadkach wskazanych w nowelizowanych przepisach? Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Ta ustawa jest dobra, ale może być martwa, i to w sposób bardzo prosty.

Niedobrze dlatego, że nie wymeldowali jej, a więc gdy osiągnęła pełnoletność, a rodzice się zapili, jedno poszło do DPS-u, drugie zmarło, to ona musiała spłacać długi, bo nie można było umorzyć, nie było podstawy prawnej. A do tego zażądano także od niej, żeby weszła w system alimentacyjny tegoż ojca, który był w DPS-ie. Otóż ustawa jest bardzo dobra, ale jeśli pieniędzy nie otrzyma samorząd, to nie będzie miał z czego finansować tej różnicy, której nie zapłaci rodzina. Jeśli tak będzie, to kierownictwo DPS-u nie będzie (Dzwonek) podejmowało decyzji korzystnych dla tych osób, bo nie będzie miało na to pieniędzy. A zatem tylko wtedy, kiedy państwo przekonacie nas, jakie środki pójdą w ślad za ustawą, będzie można za nią głosować, chociaż jest ona oczywiście - podkreślam po raz trzeci - dobra i potrzebna. Bardzo proszę, pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Mamy stary portfel, czyli osoby, w przypadku których są dopłaty z budżetu za miejsce w domu pomocy społecznej. To i dobrze. Swobodna ocena dowodów czy wszystkich dokumentów moim zdaniem jest rzeczą zasadną, ale trzeci problem, którego nie rozwiązujemy po nowemu, to problem podwyższenia opłaty za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej w stosunku do zmieniających się kosztów utrzymania.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Katalog przesłanek, które umożliwiają zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pensjonariusza domu pomocy społecznej, powinien zostać poszerzony już dawno temu. Od kilku lat problem ten poruszany był przez samych zainteresowanych, ale także stanowił temat wielu spraw sądowych, gdzie niestety częstym przypadkiem było niejednolite orzecznictwo. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, że nanoszenie tych poprawek jest tylko kosmetyką ze strony rządu. Tak naprawdę cały system odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wymaga głębokiej reformy, która powinna odbyć się po konsultacjach ze środowiskiem. W domach pomocy społecznej przebywa obecnie ok. 80 tys. osób. Jak rząd zakłada, ile takich wniosków o zwolnienie po zmianie przepisów wpłynie (Dzwonek) i jak obciąży to budżety gmin? Czy w związku z tym przewidziane są rekompensaty dla samorządów w tym zakresie? Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Chodzi mi o proponowane zmiany art. 6 ustawy z 2004 r., a konkretnie o sytuacje, kiedy dziecko wyparło czasami z pamięci fakt, że ma rodzica, bo był tak obojętny lub toksyczny, że nieraz dopiero wtedy, gdy już samo jest dorosłe, po dziesięcioleciach, przypomina mu o tym MOPS, domagając się uiszczenia opłaty za tego rodzica przebywającego w domu pomocy społecznej. Są przesłanki, żeby automatycznie ten mechanizm przerwać. Ale mam pytanie do pana ministra: Czemu nie wprowadzono również obligatoryjności zwolnienia w tych sytuacjach z opłat, jeżeli dziecko takie przedstawi dokumenty (Dzwonek) poświadczające rażące naruszenie przez rodzica obowiązków alimentacyjnych lub innych obowiązków rodzinnych? To też powinno być obligatoryjne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska.

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Ustawa przewiduje rozszerzenie katalogu podstaw zwolnienia z opłaty o wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, a nie, tak jak obecnie, przestępstwa z użyciem przemocy. Czy rząd, przygotowując ten projekt ustawy, miał informacje, ile było tych zwolnień, jeśli chodzi o wnoszone opłaty, z tytułu przestępstwa z użyciem przemocy, i czy teraz - to rozszerzenie o wszystkie przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego uważam za zasadne - też badano, o jaką grupę osób może chodzić? Słabością tego projektu ustawy jest to, że nie umiemy przewidzieć skutków finansowych dla samorządów, bo jednak na końcu za obywatela, który mieszka w danej gminie, opłatę będzie musiała ponieść (Dzwonek) gmina. Czy wobec powyższego w przyszłości będą brane pod uwagę różne formy wsparcia samorządów w tej sprawie? Bardzo proszę, pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Myślę, że nikogo na tej sali nie muszę przekonywać do tego, jak ważne są domy pomocy społecznej, które świadczą usługi opiekuńcze, bytowe. One w naszych gminach, miastach odgrywają bardzo istotną rolę. Jednocześnie też widzimy, obserwujemy, jak potrzebne jest powstawanie kolejnych miejsc w domach pomocy społecznej, jak ważna tutaj jest współpraca pomiędzy rządem i samorządem terytorialnym. Stąd też moje pytanie do pana ministra dotyczące kwestii wsparcia ze strony rządu w zakresie powstawania nowych miejsc, nowych obiektów, domów pomocy społecznej, a także kwestii wsparcia finansowego w utrzymaniu mieszkańców. Jak wiemy, te koszty z roku na rok, a w zasadzie z miesiąca na miesiąc rosną i tutaj niezbędne jest wsparcie i ścisła współpraca. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Omawiany projekt ustawy zmieniający ustawę o pomocy społecznej w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej rozszerza ten katalog, i bardzo dobrze. Te zmiany są zgodne z zasadami współżycia społecznego. Natomiast są takie sytuacje jak chociażby te związane z utratą więzi rodzicielskich, kiedy ta odpłatność nie powinna być pobierana. I tutaj mamy pewną swobodę w zakresie podejmowania decyzji. Ale mam pytanie do przedstawicieli ministerstwa: No właśnie, na jakich kryteriach można się oprzeć?

Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Nie ma pana posła. Pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Wierzę w to, że 460 posłów za nią zagłosuje, bo tak właśnie wygląda solidarna Polska, tak wygląda solidarne państwo, że o sprawach ważnych dla ludzi, o likwidacji tych niesprawiedliwości społecznych rozmawiamy w sposób absolutnie profesjonalny, transparentny. Bardzo serdecznie dziękuję za tę ustawę, tym bardziej że jest to w dniu szóstej rocznicy powołania rządu pani premier Beaty Szydło, która pokazała, jak solidarna Polska, jak solidarne państwo powinno działać. Bardzo proszę, pani poseł Urszula Rusecka, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

A drugie pytanie dotyczy skali zjawiska. Rozumiem, że od dawna to jest postulat i rzecznika praw obywatelskich, i rzecznika praw dziecka, pracowników socjalnych, instytucji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Czy w przypadku kiedy sprawa została już zakończona, ale osoba zainteresowana ponownie zwróci się o rozpatrzenie swojej sprawy, to czy to prawo będzie wtedy obowiązywać i będziemy mogli to traktować jako sprawę w toku oraz w oparciu o ten przepis zwolnić tę osobę.

Dziękuję. Ostatnie pytanie zada pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Nie, rezygnuje pan poseł z pytania. Bardzo proszę, na pytania odpowie minister

Pani Marszałek! Pani Minister! Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję za tę rzeczową, jak powiedział pan poseł Janusz Kowalski, bardzo profesjonalną dyskusję dotyczącą tego ważnego społecznie projektu. Chciałbym podziękować ministerstwu rodziny. Bardzo serdecznie dziękuję za współpracę pani przewodniczącej i całej komisji. Dziękuję wszystkim państwu parlamentarzystom zarówno obozu rządzącego, jak i opozycji.

Bo czy uznać za sprawiedliwe to, że rodzic dziecka, które nie miało z nim więzi przez kilkadziesiąt lat, którym rodzic się nie interesował, z którym nie miał ochoty mieć jakichkolwiek więzi, jakichkolwiek relacji, nawet nie płacił, nie wywiązywał się ze swoich obowiązków alimentacyjnych, po wielu latach, kiedy trafia do domu pomocy społecznej jako pensjonariusz, nagle oczekuje, że jego dziecko pokryje koszty jego pobytu w takim domu pomocy społecznej? Otóż to nie jest uczciwe ani to nie jest sprawiedliwe. A sprawa w praktyce wygląda tak, że nie jest łatwo ekskulpować się, szanowni państwo, od pokrycia takich kosztów. Oczywiście w pierwszej kolejności pracownik socjalny ocenia sytuację, dalej jest ewentualnie samorządowe kolegium odwoławcze, dalej jest ewentualnie sąd, ale przesłanki, które są zawarte w obecnej ustawie o pomocy społecznej, są na tyle ogólne, że nie pozwalają w sposób jednoznaczny rozstrzygnąć pewnych kwestii. My przygotowując ten projekt, zastanawialiśmy się, jaką drogę wybrać.

W kuluarach rozmawiałem także z posłami opozycji, którzy mówili, że to jest dobre rozwiązanie. Dziękuję za te dzisiejsze głosy. Można było przyjąć drogę, którą proponował wspominany tutaj przez państwa rzecznik praw obywatelskich czy rzecznik praw dziecka, czyli zastosować klauzulę zasad współżycia społecznego.

My przyjęliśmy rozwiązanie, że trzeba wskazać konkretne sytuacje.

Mam nadzieję, że ją zupełnie wyeliminujemy. Moim zdaniem tylko w ten sposób mogliśmy to zrobić.

To prawda, pracownik socjalny jest tym, który w pierwszej kolejności bada sytuację. Jest wywiad środowiskowy, który jest przeprowadzany. Szanowni państwo, oto pismo z 2017 r. Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Tym pismem dysponuję i na poszczególnych etapach legislacyjnych przekazywałem treść tego pisma.

Otóż w żadnym razie nie mogę się zgodzić. Może ona jest 1-stronicowa, ale jest istotna, niesie daleko idące konsekwencje.

Dlaczego tak musi być? Życie niesie różne sytuacje za sobą, więc czasami osoba nie jest zainteresowana, żeby występować na drogę sądową o takie orzeczenie.

Rażący - to jest zdefiniowane.

Dziecko musi mieć zapewniony właściwy rozwój, jeżeli chodzi o edukację, kulturę, sport, duchowość. Wiadomo, rodzice zajmują się, bo to też wynika z konstytucji, wychowaniem dziecka. Więc ten katalog.

Dlaczego?

Pan poseł musi wiedzieć, że są także prywatne domy pomocy społecznej. Mam nadzieję, że to nie zaburza jego wolnościowego sposobu patrzenia na funkcjonowanie państwa. Czy będzie wsparcie finansowe? W wielu miejscach pojawiło się to pytanie ze strony państwa parlamentarzystów. Otóż szanowni państwo, my dyskutowaliśmy z komisją wspólną rządu i samorządu, i to była jedyna uwaga do tego projektu zgłoszona przez tę komisję. Nie będzie takiego wsparcia, to będzie robione w ramach limitu, który przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego.

Jeżeli będzie takie oczekiwanie, to ja je podam. Musi to być przeprowadzone w ramach limitu. Bo jak to określić, szanowni państwo? Państwo pytacie mnie, czy jeżeli były takie sytuacje, to czy możemy powrócić do nich, sprawdzić, jeszcze raz przeprowadzić wywiad środowiskowy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie ma takiej możliwości, nikt nie ma.

Czy będą nadużycia?

Jest, art. 2 jest przepisem przejściowym i mówi, że do spraw, które były wszczęte, a niezakończone, kiedy wejdzie w życie ta regulacja, stosowana będzie nowa regulacja. Ale niezależnie od tego zawsze, szanowni państwo, będzie możliwość aktualizacji, niezależnie od wszystkiego. Sprawa przesłanek. Jakie są przesłanki, które będzie brał pod uwagę pracownik socjalny? One są, szanowni państwo, określone w ustawie o pomocy społecznej w art. 107 ust. 5b.

Czy były więzi, jeżeli ktoś wysyłał korespondencję do swojego rodzica, a rodzic nie odpowiadał przez całe lata, nie interesował się, nie było kontaktu, nie odwiedzał, to wyjdzie podczas wywiadu środowiskowego, szanowni państwo. Pracownicy socjalni nie powinni mieć z tym większych problemów, a jeżeli będą mieli, to zawsze jest droga odwoławcza. Tak jak mówię, również na drodze administracyjnej będzie to badane przez sąd. Jeżeli chodzi o kwestię aktualizacji, to już mówiłem. Będzie możliwość aktualizacji sytuacji, ponowne badanie, czy dalej taka osoba musi płacić na pensjonariusza czy nie.

Nie. Nie wchodzimy w ogóle w te kwestie. My tak naprawdę tworzymy mechanizm. Nie ingerujemy w to, w jaki sposób jednostka samorządu terytorialnego sobie to ustala. To już jest kwestia, która leży poza naszym zakresem. Pytanie, czy były konsultacje.

Ale to już wyjaśniałem i mówię, że w orzecznictwie także jest to dosyć szczegółowo określone. Jak najbardziej.

Ten wywiad będzie również sprawdzany ewentualnie przez samorządowe kolegium odwoławcze oraz ewentualnie sąd administracyjny. Czy były badania, ile może być takich przypadków? Nie ma takich badań, staraliśmy się to wyciągnąć, nie były one nigdy prowadzone w tym zakresie.

Nie, szanowni państwo, to, co przygotowaliśmy, jest w naszym przekonaniu wystarczające do tego, żeby zmienić niesprawiedliwą sytuację osób, które czasami przez lata muszą płacić za to, żeby ktoś mógł przebywać w domu pomocy społecznej, a nie miały z nim żadnej więzi.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 5. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku (druki nr 1727 i 1748) Bardzo proszę pana posła Dariusza Olszewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu w dniu 15 listopada br. połączone Komisje: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły sprawozdanie o projekcie rządowym z druku nr 1727, tj. o projekcie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Założeniem projektu jest dostarczenie odpowiednich podstaw prawnych w celu stworzenia warunków właściwym jednostkom samorządu terytorialnego do terminowej realizacji przedsięwzięć i właściwej organizacji planowanych na 2023 r. igrzysk europejskich, które mają odbywać się na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Po merytorycznej dyskusji z udziałem przedstawicieli samorządów ww. województw oraz przedstawicieli prezydenta miasta Krakowa komisje zakończyły pierwsze czytanie projektu i podjęły decyzję o przystąpieniu do jego niezwłocznego rozpatrzenia. W trakcie szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje wprowadziły do niego cztery poprawki, które m.in. usprawniły tryb transferowania środków na inwestycje realizowane w związku z organizacją igrzysk, a także zmieniły proponowany skład rady nadzorczej spółki celowej powołanej w celu realizacji przedsięwzięć związanych z tymi igrzyskami. Wysoka Izbo!

Za to bardzo serdecznie chciałbym tym posłankom i posłom podziękować. Komisje w sprawozdaniu wnoszą o przyjęcie załączonego projektu ustawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Igrzyska europejskie będą wielką promocją dla sportu polskiego. To sztandarowa impreza sportowa, rozgrywana co 4 lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich. Najlepsi sportowcy Starego Kontynentu będą rywalizować w 23 dyscyplinach. Polska na pewno sprosta temu wyzwaniu - mamy duże doświadczenie w organizowaniu dużych imprez sportowych. Igrzyska będą miały ogromne wsparcie rządu polskiego, będą świetną okazją, aby pokazać nasze możliwości, i będą wielką promocją Polski. Projekt ustawy dotyczy umożliwienia województwu małopolskiemu, województwu śląskiemu oraz miastu Kraków terminowego wykonania przedsięwzięć oraz stworzenia warunków dla właściwej organizacji igrzysk oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy Host City Contract. Na wspólnym posiedzeniu w dniu 15 listopada br. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadziły pierwsze czytanie oraz rozpatrzyły powyższy projekt ustawy. Uprzejmie informuję Wysoką Izbę, że ww. projekt ustawy nie budzi zastrzeżeń i zapewni umożliwienie województwu małopolskiemu, województwu śląskiemu oraz miastu Kraków terminowego wykonania przedsięwzięć związanych z organizacją III Igrzysk Europejskich, letnich, w 2023 r. W związku z tym w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość rekomenduję jego przyjęcie, zgodnie ze sprawozdaniem z druku nr 1748. Jednocześnie składam cztery poprawki, aby projekt był jeszcze lepszy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 30 miesięcy minęło od momentu przyznania organizacji igrzysk europejskich Małopolsce. I co przez ten okres się stało? Nic. Ja się dzisiaj nie dziwię, że na sali nie ma ani jednego posła, ani jednej posłanki ze strony PiS-u z Małopolski, bo to, co państwo zaproponowaliście nam w tej specustawie, nie jest warte poparcia. A przypomnę, jak przebiegały ostatnie miesiące. Nie brakowało zapewnień: miliard na krakowskie inwestycje. Budżet państwa weźmie na siebie koszty organizacji igrzysk w Krakowie. Ustawa będzie do końca kwietnia, do końca czerwca, do końca września - to wszystko zapewnienia głównie ministra Sasina, który jest pełnomocnikiem rządu i wielkim nieobecnym dzisiaj. Ale pamiętajmy - Sasinowi nic przez ostatnie 6 lat jeszcze się nie udało zrobić, i to jest największe zagrożenie dla tych igrzysk.

160 mln zł na opłatę licencyjną i na opłaty dla europejskich federacji sportowych. Nic więcej. A gdzie inwestycje sportowe? Gdzie inwestycje infrastrukturalne? Kto ma za to zapłacić? Kto weźmie na siebie odpowiedzialność za poniesienie wszystkich kosztów? Cała nadzieja w tym, że obecny minister Rabenda niewiele wie o tym projekcie i być może wczoraj się pomylił, mówiąc, że 160 i koniec, ani złotówki więcej.

Składamy trzy poprawki. Niewiele.

Od jej poparcia, uwzględnienia zależy to, czy poprzemy tę ustawę, czy nie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Miszalski. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście idea organizacji igrzysk europejskich brzmi pięknie.

Pierwsza kwestia to wymiar sportowy i promocyjny tej imprezy. Wymiar promocyjny wcale nie jest tak wielki, jak by się mogło wydawać. Wymiar sportowy pewnie będzie trochę większy, ale jednak Kraków był jedynym starającym się o tę imprezę. Ano dlatego, że często koszty organizacji takiej imprezy przekraczają korzyści z niej płynące. Przypomnijmy sobie igrzyska zimowe w Krakowie. 2014 r., referendum, 70% krakowian było przeciwnych tej imprezie, która miała dużo większy i sportowy, i promocyjny wymiar. Zresztą Rada Miasta Krakowa 1 września podjęła uchwałę o rekomendacji wycofania się z igrzysk, jeżeli nie będzie gwarancji finansowych. Trudno się dziwić, ponieważ od 2 lat zapewniacie, że te finanse i te gwarancje będą, ale do tej pory nic, żadnych konkretów nie przedstawiliście i w tej ustawie również tych gwarancji nie ma. A gdzie są pieniądze na transport, na bezpieczeństwo, na ochronę zdrowia, na zakwaterowanie, na utrzymanie czystości podczas tej imprezy?

Rada miasta wnioskowała jeszcze o stadiony Hutnika, Wieczystej - załącznika brak. Co więcej, minister Bortniczuk obiecywał specjalny program dedykowany igrzyskom, który powinien być w tej ustawie.

Dziękuję bardzo. Pani poseł Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Panie Ministrze! Jestem tu w imieniu swoich wyborców i wyborczyń. Jestem tu jako mieszkanka Krakowa i zabieram głos w imieniu tych, którzy w 2014 r. już raz powiedzieli: nie igrzyskom, kiedy 70% osób biorących udział w referendum sprzeciwiło się tej kosztownej imprezie. Natomiast teraz miasto, województwo i rząd uparły się, aby realizować drogie i niepotrzebne igrzyska, kiedy w Krakowie wciąż brakuje naprawdę potrzebnych rzeczy takich jak przedszkola, żłobki czy nawet chodniki. Rząd i samorządy chcą wydać miliony. Ile? Nie wiemy, dlatego że w ciągu 30 miesięcy, jakie upłynęły od dnia złożenia wniosku aplikacyjnego, nie przedstawiono budżetu imprezy. Bardzo chciałabym to wyliczyć, ale nie wiem dokładnie, bo nadal nie przedstawiono listy inwestycji innych niż sportowe. Ta lista jest największą tajemnicą skrywaną, nie wiem gdzie, w którym ministerstwie. Jeśli chcemy podnosić jakość życia, to mam wiadomość: to robi się zupełnie inaczej, niż organizując imprezę, która do tej pory służyła wschodnim satrapom, dyktatorowi Azerbejdżanu i dyktatorowi Białorusi, do organizacji której nie zgłosiło się żadne inne państwo europejskie i która swój żywot najprawdopodobniej zakończy w Krakowie, bo nie ma kandydatów do organizowania kolejnych edycji. Chciałam też zapytać, jak te mgliście obiecane - właściwie w jakim trybie? - inwestycje mają podnieść jakość życia, skoro mówi się np. o budowie Trasy Balickiej, która jak alarmują specjaliści od transportu i ekolodzy, jest przeskalowanym obiektem z lat 70., w ogóle nieprzystającym do współczesnej myśli o tym, jak powinien być organizowany transport w miastach, i która zniszczy cenne tereny przyrodnicze. Potrzebujemy czystego powietrza, potrzebujemy terenów zielonych, potrzebujemy rozsądnej polityki transportowej, potrzebujemy rozwoju miast, a nie tej imprezy, która naprawdę niczemu się nie przysłuży. Z powodu własnych i nietrafionych ambicji chcecie państwo organizować niepotrzebną imprezę, której kosztami i uciążliwościami zostaną obarczeni mieszkańcy i mieszkanki Krakowa. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! My w tej kadencji funkcjonujemy coraz częściej w logice stanu wyjątkowego. Tak się dzieje ze względu na zewnętrzne okoliczności. To jest uzasadnione, kiedy mamy do czynienia z pandemią. Ale nie możemy zapominać, że podczas takich realnych albo wykreowanych sytuacji zdarzają się rzeczy karygodne. Podczas pandemii mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi nadużyciami. Wciąż nie są wyjaśnione zakupy respiratorów, maseczek, testów. To są realne rzeczy, które się wydarzyły właśnie dlatego, że działamy w sytuacji stanu wyjątkowego, trzeba na gwałt, szybko wydawać pieniądze, szybko realizować projekty. I z tego względu ten projekt, który państwo przedstawili obecnie, dotyczący igrzysk europejskich, wydaje nam się wątpliwy. On w wielu miejscach wprowadza właśnie tę logikę stanu wyjątkowego, kiedy ją rozumiemy szeroko, tzn. upraszcza np. procedury związane z planowaniem przestrzennym, upraszcza czy zawiesza mechanizm zamówień publicznych, ogranicza przepisy prawa restrukturyzacyjnego. W tych okolicznościach, kiedy mamy na razie do czynienia z tak bardzo słabym przygotowaniem tej imprezy, kiedy decyzje, umowy nie są podpisane, decyzje się wloką, wszystko ma być załatwione w ciągu kilkunastu miesięcy, naszym zdaniem jest to mieszanka wybuchowa i ona będzie prowadziła do wadliwych decyzji, może prowadzić do korupcji. Dlatego mamy głębokie przeświadczenie, żeby tej ustawy nie popierać. Zgłosimy poprawkę związaną z lepszą kontrolą wydawania tych środków, bo to jakoś, mamy nadzieję, ograniczy negatywne aspekty tej ustawy, jeżeli w ogóle dojdzie do jej przyjęcia, jeżeli w ogóle dojdzie do tych igrzysk, bo na razie wszystko wygląda na to, że te igrzyska się nie odbędą. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie!

Panie Ministrze! Od lat przyglądam się przygotowaniu tego projektu.

Dlaczego? O czym nie mówią przedstawiciele innych klubów parlamentarnych, które krytykują ten projekt? Dziś mamy czas wielkiego zamieszania. Zawsze Karta Olimpijska, wielkie wydarzenia sportowe mówiły o wartościach. Te igrzyska europejskie, które rzeczywiście są nowym projektem, po raz trzeci będą organizowane, są oparte na wartościach Karty Olimpijskiej, które szczególnie w czasach zamętu trzeba przypominać. Myślę, że ten czas igrzysk w Krakowie - mam nadzieję, że te igrzyska dojdą do skutku - będzie dobrym czasem na to, żeby o tych wartościach mówić. Po drugie, to będą pierwsze igrzyska w Unii Europejskiej. Wiem, że europejski komitet olimpijski stara się, żeby była to impreza pod patronatem Brukseli. To byłby też wymowny sygnał do tego, że ta impreza wzrasta i ma większe znaczenie. Od tych igrzysk w Krakowie rzeczywiście kategoria sportowców, którzy będą brać w nich udział, zupełnie się zmieni, z drugiej na pierwszą kategorię, ponieważ, jak to było wczoraj tłumaczone, będą to również kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu. A więc tutaj pojawią się sportowcy, którzy będą chcieli w tych dyscyplinach walczyć o tę przepustkę do igrzysk. To tytułem takiego prawdziwego pokazania, co to za impreza. Oczywiście uważam, że po pandemii ponowienie promocji Polski w oparciu o dużą imprezę, która zgromadzi sportowców z różnych stron Europy, może być dobrze wykorzystane. Ale czy będzie?

Dzisiaj pod presją czasu musimy poprawić to, co państwo wczoraj przedłożyliście w komisji, o poprawki, które zgłaszam, nie wchodząc w szczegóły.

Natomiast chciałbym złożyć pięć poprawek w imieniu klubu.

Wysoka Izbo! Igrzysk i chleba. Praktyka organizowania publicznych rozgrywek i rozdawnictwa miała na celu łagodzenie napięć społecznych i zyskiwanie popularności niezbędnej w działalności politycznej oraz odwracanie uwagi społeczeństwa od działań polityków. Służyły prewencyjnej polityce zapobiegania rozruchom i przejawom niezadowolenia.

Gratuluję planu marketingowego. Oczywiście są to pieniądze nie tyle wyrzucone w błoto, co zwyczajnie przepalane najprawdopodobniej tylko dlatego, żebyście wy na tym coś zyskali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Igrzyska europejskie nie mają dużego sportowego znaczenia. Być może w przyszłości będzie inaczej, ale to nie będzie, jak zapowiadał wicepremier Jacek Sasin, największa sportowa impreza organizowana w Polsce w 2023 r. Nie trąbmy więc, panie pośle Matuszewski, w fanfary, nie ruszajmy dział propagandowych w tej sprawie, choć pewnie ktoś chciałby już bić monety albo drukować okolicznościowe banknoty właśnie z tej okazji. To zdumiewające, że dopiero dzisiaj rozpoczynamy procedowanie nad ustawą, a przecież minęło prawie 30 miesięcy od dnia, kiedy Kraków został organizatorem igrzysk. Czy został? Oto jest pytanie. Rządzący mówią o wielkiej imprezie, a organizacyjnie wszystko jest w powijakach. Podobnie powinno być z organizacją tej imprezy. Do końca października Kraków miał otrzymać gwarancje rządowe. Nie otrzymał. Kraków jest wielką marką. Nie występował o organizację igrzysk, o czym mało kto wie. Kraków został o tę organizację poproszony. Kraków słusznie nie chce wydać ani jednej zbędnej złotówki.

To kwota, którą trzeba wpłacić Stowarzyszeniu Europejskich Komitetów Olimpijskich, a na organizację igrzysk potrzeba grubo ponad 300 mln zł. Na to gwarancji nie ma. Kraków wyraźnie określił listę inwestycji, które powinny być sfinansowane z budżetu państwa.

Drodzy Rządzący! Nie marnujcie czasu na zastanawianie się, kto i przez kogo ma być powołany, by zasiadać w spółce celowej i radzie nadzorczej. Jeśli nie wiecie, jak zabrać się do organizacji tak dużej imprezy, to zapraszam w sobotę do Łazisk Górnych na charytatywny turniej piłki nożnej. Młodzi zawodnicy zagrają dla ciężko chorej Dorotki Dąbrowskiej. Będzie okazja, żeby porozmawiać z wolontariuszami z Polski 2050, a Dorotkę zaprosić na igrzyska do Krakowa. Tylko do kogo ja to mówię? Wicepremiera Sasina nie ma. Nowego ministra sportu Kamila Bortniczuka także nie ma dzisiaj z nami. Bardzo proszę, pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dwie sprawy. Po pierwsze, po co kolejna specustawa o kolejnych igrzyskach? Dlaczego? To jest cytat z uzasadnienia: Projektowana ustawa ma stworzyć warunki umożliwiające właściwą organizację igrzysk. Czyli państwo przyznajecie, że koszmarne prawo, które tutaj od lat wytwarzacie, nie zapewnia warunków do właściwej organizacji igrzysk. Dlaczego nasze prawo nie zapewnia warunków do np. właściwej organizacji igrzysk, mistrzostw, Światowego Forum Miejskiego, budowy płotu na granicy czy Pałacu Saskiego? Może to jest właśnie moment na taką refleksję, że chyba robicie to źle. Może to jest sygnał, jaki natura dyskretnie wam wysyła, jakim natura wam podpowiada, żebyście przestali uchwalać kolejne regulacje, skoro sami potem potrzebujecie specustawy, żeby każde większe przedsięwzięcie dokończyć, żeby tą specustawą te regulacje uchylić czy ominąć. Może to znaczy, że produkujecie tu buble prawne, których nie chce się wam potem przestrzegać, ale oczekujecie jednocześnie, że obywatele będą do ostatniego papierka musieli to robić, i to nawet w sprawach ważniejszych niż jakieś tam skoki na igelicie czy gra w badmintona, bo mieszkania czy sklepy są ważniejsze od rozrywek. Po drugie, dlaczego niby w ogóle państwo bierze się za jakieś igrzyska, za jakieś kolejne sasinalia? Jeśli są chętni, żeby oglądać, jak inni grają w badmintona czy odbijają piłkę na piasku, to super, niech tę rozrywkę sfinansują od początku do końca z własnych pieniędzy.

Uczciwe jest tylko takie rozwiązanie, kiedy każdy finansuje swoją zabawę i swoje rozrywki. Głosowanie portfelami jest bardziej uczciwe niż sondaże. Oczywiście taktyka chleba i igrzysk sprawdza się od dawna, ale cesarze przynajmniej nie potrzebowali specustawy do każdych igrzysk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Stanisław Bukowiec, Porozumienie. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 30 maja 2019 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków 2023 r. W uchwale zadeklarowano poparcie dla zgłoszenia kandydatury miasta Krakowa i województwa małopolskiego jako gospodarza imprezy. Igrzyska europejskie są szansą na promocję Polski, ale przede wszystkim promocję Małopolski, Śląska i Krakowa. Według zapowiedzi organizatorów w różnych dyscyplinach sportowych ma wziąć udział 4 tys. zawodników z 50 krajów.

Mam pytanie do pana ministra Sasina. Skąd takie opóźnienie w przygotowaniu tej imprezy?

O konieczne środki na te inwestycje zabiegają prezydenci i burmistrzowie małopolskich miast, przede wszystkim Krakowa i Tarnowa. Niestety deklarowana przez rząd kwota jest niewystarczająca, aby można było odpowiednio przygotować infrastrukturę tych miast, by dobrze i godnie przyjąć sportowców z całej Europy. Trzeba powiedzieć jasno: bez dodatkowych środków dla samorządów nie jest możliwe przeprowadzenie igrzysk europejskich, a organizacja imprezy bez udziału np. miasta Krakowa jest bezzasadna. W obecnej trudnej sytuacji gospodarczej samorządów nie stać na kolejne wydatki, dlatego gwarancje finansowe państwa są konieczne. Apelujemy do rządu o zwiększenie dotacji dla małopolskich samorządów Krakowa, Tarnowa, Krynicy i Zakopanego o 300 mln zł po to, aby igrzyska europejskie mogły być zrealizowane. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Agnieszka Ścigaj, Polskie Sprawy. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Mówię: potencjalnie, ponieważ wcale nie jest powiedziane, że te igrzyska się odbędą.

Samemu miastu Kraków promocja za kilkaset milionów, które ono samo miałoby wydać, nie jest potrzebna. Miasto Kraków jest marką samą w sobie i jest znaną marką.

Ale oby w 2023 r., kiedy zbiegną się wybory, nie była to tylko i wyłącznie promocja polityków, którzy bardzo chętnie będą wieszać medale w świetle jupiterów. Szanowni Państwo!

Wydaje się, że w momencie kiedy miasto potrzebuje impulsu gospodarczego - tak jak każde miasto w Polsce, każdy samorząd po pandemii, ale też z uwagi na wprowadzenie zapisów Nowego Ładu potrzebuje impulsu gospodarczego - będą tylko wydatki. Jak z tego wynika, 160 mln zaplanowane w tej ustawie to jest tylko składka do europejskich organizacji sportowych, to nie są żadne pieniądze na inwestycje.

Bez środków finansowych to nie będzie żadna promocja.

Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Czy widzimy pana ministra sportu? Czy widzimy pana premiera?

A czy impreza się odbędzie, czy nie odbędzie, to już nas po prostu nie interesuje.

Bardzo proszę, pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Wysoka Izbo! Z projektu umowy Host City Contract wynika, że w ramach poniesionych kosztów za prawo do zorganizowania III Igrzysk Europejskich oraz za przyznanie praw komercyjnych spółka celowa przekaże świadczenie pieniężne w wysokości do 160 mln zł.

Jakie środki będą przeznaczone w przypadku wsparcia finansowego na infrastrukturę sportową? Pan poseł Marek Rutka, Lewica. Wysoka Izbo! Dwie pierwsze edycje europejskich igrzysk zorganizowali dyktatorzy z Azerbejdżanu i Białorusi. Do organizacji III edycji igrzysk nie zgłosił się żaden kraj oprócz Polski. Zarówno Ilham Alijew, jak i Aleksander Łukaszenka wykorzystali sport do legitymizowania swoich autorytarnych rządów. Jednym z orędowników tej kosztownej imprezy jest minister Sasin znany z tego, że był w stanie wydać 70 mln zł na wybory, które nigdy się nie odbyły.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Aleksander Miszalski, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Teoretycznie fajny projekt, teoretycznie fajna impreza, może nie wybitna, ale jednak. Minęło 30 miesięcy, zostało jeszcze 18, a dalej jesteście w lesie. Trasa Balicka, węzeł opatkowicki, przebudowa Okulickiego i Buszka. Jest ustawa, brak jest inwestycji. Brak kosztów organizacji, brak kwot w rozporządzeniach w sprawie inwestycji sportowych - o nie również proszę.

Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze!

Mówienie o tym, że to jest niska ranga (Dzwonek), nie jest właściwe. Chciałem zapytać pana ministra, czy Kraków ma już całą wizję związaną z obiektami sportowymi poza tą dwunastką, która jest wykazana w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Dariusz Olszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek!

Nie chcę się licytować, kto zrobił ich więcej, ale zapraszam na każdy mecz Polskiego Związku Rugby, już w najbliższą sobotę na stadionie Polonii Polska będzie grała ze Szwajcarią. Również pan się przekona, że organizacja imprez jest na najwyższym poziomie. Ale przechodząc do ustawy o wsparciu do przygotowań do III Igrzysk Europejskich, chciałbym poprosić o informację - chociaż tutaj już mój przedmówca w części o tym mówił - dotyczącą ilości dyscyplin, które będą rozgrywane podczas III Igrzysk Europejskich. Ile z tych dyscyplin, panie ministrze, będzie jednocześnie eliminacjami do igrzysk letnich Paryż 2024? Pani poseł Elżbieta Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam takie pytanie. Ponieważ igrzyska europejskie będą doskonałą promocją regionu województwa małopolskiego, śląskiego, a przede wszystkim miasta Krakowa, ale także szansą na pokazanie sprawności państwa. Dobrze, że powstała proponowana lista rozwiązań prawnych - czy sposobu finansowania, czy zasady tworzenia i działania spółki celowej, czy warunków umowy. Jak wiemy, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa to 103 mln zł. W związku z tym mam dwa pytania do pana ministra. Jaki będzie zakres działań ministra właściwego do spraw monitorowania wydatków? I czy w przypadku przekroczenia limitu na dany rok mechanizm korygujący będzie polegał na ograniczeniu dalszego finansowania przedsięwzięć na rok kolejny? Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Mam uprzejmą prośbę do Platformy Obywatelskiej, do etatowych malkontentów i psujów. Igrzyska europejskie są ważną imprezą dla Polski. To, że dzisiaj z tej strony atakujecie pana ministra Sasina, krytykujecie rozwiązania polskiego rządu. Jesteście przeciwko obronie polskiej granicy, jesteście przeciwko Pałacowi Saskiemu, jesteście przeciwko każdej polskiej imprezie. Chyba że to by były igrzyska dla aktywistów LGBT, to wtedy byście się zgodzili. Bardzo proszę, pan poseł Patryk Wicher, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo! Słyszę tylko, że Małopolska to Kraków. Kraków jest przepięknym miastem, ale jako mieszkaniec Małopolski mieszkający w Nowym Sączu i na południu tego pięknego województwa w To jest Krynica, to jest Tarnów, to jest Nowy Sącz.

Ponadto, moi drodzy państwo, zwróćmy uwagę na to, że te wydarzenia organizują federacje europejskie, federacje sportowe wszystkich krajów Unii Europejskiej, całej Europy, a nie jacyś dyktatorzy. A więc proszę się troszeczkę douczyć, moi drodzy państwo, i nie obrażać imprez na poziomie europejskim. I taka jest różnica między nami a wami. Pytanie, panie ministrze, czy te wszystkie dyscypliny sportowe, które będą realizowane, mogą liczyć na dodatkową promocję w czasie tej imprezy, po tej imprezie (Dzwonek) i czy to wpłynie na rozwój tych dyscyplin. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Oczywiście sport, rywalizacja, karta olimpijska - sam byłem zawodowym sportowcem, wiem, że to są ważne przesłania. Natomiast igrzyska europejskie, trzeba wspomnieć, to jednak nie są te główne, najważniejsze igrzyska światowe, które cieszą się największą popularnością. Państwa retoryka, że to wspaniała promocja - troszeczkę bym się z tym jednak wstrzymał, patrząc po tym, co się działo i w Azerbejdżanie, i na Białorusi, że to taka wspaniała promocja regionu czy też miasta.

Przypomnę, ok. 4 tys. sportowców, koszty są szacowane na ok. 300 mln zł (Dzwonek), czyli transport, nocleg, wyżywienie, opieka medyczna, bezpieczeństwo w tym trudnym czasie COVID-owym. Kto za to zapłaci? Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Chciałoby się powiedzieć: jaki rząd, takie imprezy. Przypominam Euro 2012 - wspaniała impreza i to była rzeczywiście piękna promocja kraju, a wy w tej chwili rzeczywiście, jeżeli mówicie o sprawności działania, to to jest na razie pasmo porażek, szanowni państwo. 30 miesięcy nie zrobiono nic i to jest wielki problem. Myślę, że panie ministrze, jako poseł z Wielkopolski, ale myślę, że tutaj przede wszystkim Małopolska oczekuje jasnej deklaracji, czy pieniądze, dodatkowe pieniądze na organizację się znajdą, bo wczoraj podczas prac w komisji usłyszeliśmy z pana ust, że tych dodatkowych pieniędzy na organizację nie będzie. Mówimy tutaj o blisko 400 mln zł. To jest teraz ten czas, aby stanąć i jasno to wszystko powiedzieć. A jeżeli posłowie PiS-u mówią, że jest to szansa na wielką promocję Polski. W takim towarzystwie, z panem Łukaszenką obok, biorąc pod uwagę szczególnie sytuację, która jest w tej chwili (Dzwonek) na polskiej granicy - nie jestem tego pewny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo!

Dlatego że od momentu, kiedy rząd zdecydował, że w Polsce odbędą się takie igrzyska, minęło już 2,5 roku, 30 miesięcy, a my nadal mamy wrażenie, że w zasadzie rząd nie jest kompletnie dogadany z samorządami - czy to miejskimi, czy wojewódzkimi - w zakresie organizacji i podziału zadań. Impreza będzie kosztować ponad 400 mln zł. Wiemy, że samorządy nie zadeklarowały wsparcia w tym zakresie, uznając, że są pilniejsze wydatki. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Tych terminów podawanych przez was było już bardzo wiele, do dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Kto w rządzie zajmuje się organizacją i przygotowaniem igrzysk europejskich? Z jednej strony ustawa jest przygotowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale z drugiej strony jako płatnik jest wskazane ministerstwo kultury fizycznej i sportu. Pytam: Gdzie jest minister sportu? Gdzie są jego deklaracje? Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest jego zdanie i jakie środki, bo to od niego zależy, będą przeznaczone na konkretne inwestycje. Tych odpowiedzi po prostu nie ma. Zaangażowanie posłów i polityków PiS-u też skończyło się tak naprawdę w ubiegłym roku. W tym roku nie macie państwo nic do powiedzenia, [[Dzwonek]] bo wszyscy wiemy doskonale, że ta sprawa jest spóźniona, a w tym projekcie ustawy nie dajecie złotówki na organizację igrzysk i na inwestycje. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tutaj jeden z panów posłów z Prawa i Sprawiedliwości twierdził, że wszyscy czekają i cieszą się na te igrzyska. Panie Pośle! Naprawdę, wystarczy kontakt z wyborcami i pan zrozumie, że większość wyborców, większość Polaków w ogóle nie wie, że takie igrzyska są. Już nie mówię o tym, że miałby ktoś wiedzieć, że są one organizowane w Polsce. To jest oczywiście też wynik nieudolności rządu Prawa i Sprawiedliwości, który de facto nic w tej sprawie nie robi.

Bez środków centralnych z pewnością nie uda się tego zrobić. Ma zostać powołana spółka celowa. Bardzo bym prosił (Dzwonek) o informację, czy członkowie rady nadzorczej będą pobierali wynagrodzenie, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Bardzo proszę, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Wierzę w to, że te igrzyska odbędą się, zostaną sprawnie zorganizowane, nie tak jak zapowiadane przez działaczy Platformy zimowe igrzyska olimpijskie, na które województwo małopolskie zarządzane przez Platformę Obywatelską wydało 20 mln zł, a igrzyska się nie odbyły. Być może Kraków nie potrzebuje takiej promocji, chociaż wydaje mi się (Dzwonek), że nie ma miejsca na mapie, które by nie wymagało promocji.

Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Grabczuk, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jestem wielkim zwolennikiem organizacji różnych imprez sportowych na terenie naszego kraju, bowiem sport potrafi łączyć, sport potrafi być ponad podziałami politycznymi, partyjnymi, ale przede wszystkim sport dzisiaj to niezwykle piękna promocja regionów, miast i poszczególnych państw. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co do tej pory robiliście? Dzisiaj wprowadzacie specustawę, żeby zdążyć. Każdy, kto organizował ważną imprezę o zasięgu europejskim czy światowym, wie, że dzisiaj powinna być wielka promocja tej imprezy w Europie i na świecie, chociaż to są igrzyska europejskie. Zawodniczka z mojego klubu Katarzyna Krawczyk zdobyła na nich kiedyś tytuł wicemistrzyni. To będą eliminacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu i to jest również dla nas wielka szansa. Bardzo proszę, pan poseł Ireneusz Raś, Koalicja Polska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Po pierwsze, chciałem prosić o to, aby te poprawki, których złożyłem pięć, rozważyć nie politycznie, tylko merytorycznie, bo one są głęboko skonsultowane również z samorządem i będą służyć lepszej realizacji tych zadań, które w krótkim czasie muszą być wykonane przez spółkę celową. A z drugiej strony chciałem pana zapytać, panie ministrze, i zaapelować do pana, żeby pan przy okazji udzielania odpowiedzi wyszedł i powiedział, jakie konkretne cele Polska może osiągnąć. Jakie chcecie osiągnąć cele, zyski z tej imprezy? Bo tutaj jest skakanie po tej imprezie. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Ile potrzeba czasu na stworzenie ustawy? Jeśli weźmiemy pod uwagę ten projekt, to wychodzi na to, że 2,5 roku. Szanowni Państwo! 2,5 roku to dziecko zdąży się nauczyć chodzić, jeść i w satysfakcjonującym stopniu obsługiwać smartfona, a wy nie potrafiliście w tym czasie stworzyć dobrej ustawy, już nie mówiąc o tym, że powstała ona dopiero po 30 miesiącach od decyzji. Skoro politycy Prawa i Sprawiedliwości mówili o tym, że jest to bardzo ważny projekt, bardzo ważna impreza, to dlaczego w ten sposób do tej imprezy nie podeszli politycy i ludzie odpowiedzialni w ministerstwie sportu? Dziękuję, panie pośle. Pan poseł Marek Matuszewski, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Myślałem, że na tej sali są wszyscy za sportem, za tym, żeby organizować tę wielką imprezę w Polsce, ale niestety jest ta wielka krytyka ze strony szczególnie Platformy Obywatelskiej, która wydaje mi się, że jest przeciwna organizacji tej imprezy, tego wielkiego wydarzenia sportowego w Polsce. Wczoraj na posiedzeniu połączonych Komisji: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej słyszałem z ust gospodarzy, samorządowców, z ust przedstawicieli Krakowa, że są za, że są zadowoleni. Ja mogę powiedzieć, że przygotowania, wyczerpująca informacja złożona przez Ministerstwo Aktywów Państwowych kierowane przez premiera Jacka Sasina, to wszystko zasługuje na wielkie podziękowania, bo wiem doskonale. Tak, opozycja nie chciałaby pokazywać światu sukcesów Polski (Dzwonek), sukcesów organizacyjnych. Dziękuję, panie pośle.

Chciałem powiedzieć, biorąc pod uwagę liczbę wiceministrów, ministrów, że 160 mln to jest 1 mln z kawałkiem na głowę. Chciałbym dostać listę ministrów, którzy już wpłacili swoją składkę, swoją zrzutkę, bo skoro rząd bierze na siebie, to znaczy, że rząd bierze na siebie, a nie Polacy, a nie nasz budżet, nie dyskutujmy tutaj o tym, że to z podatków będzie zrobiona ta wasza impreza. Drugie. W związku z tym, że powstanie spółka celowa, która będzie to robiła, a ustawa antysitwowa jeszcze nie będzie funkcjonowała, bo się zabezpieczyliście i zrobiliście ją dopiero od nowej kadencji, chciałem się zapytać, jaki będzie stosunek ludzi, którzy będą mieli partyjną legitymację oraz nazwiska podobne do nazwisk polityków PiS-u, jaki będzie stosunek tych ludzi do ludzi, którzy znają się na sporcie i organizacji imprez masowych w tej spółce. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Ja proponowałem wizytę w Łaziskach Górnych po to, by zobaczyć, jak organizuje się mały turniej, jak to pan powiedział, charytatywny, by zobaczyć, że to nie jest sprawa do załatwienia w ciągu jednego dnia. Panie Pośle Matuszewski! Prosiłem bez tub propagandowych. Nie ma już posła z Nowego Sącza. Chciałbym go zapytać, czy on w ogóle wie, jakie dyscypliny będą organizowane w ramach igrzysk europejskich. Podobnie czy pani posłanka z Tarnowa wie, czy w Tarnowie w ogóle odbędą się te igrzyska? Nawet w takiej sprawie polaryzujecie scenę polityczną, nawet w takiej sprawie sportowej. Panie Pośle Matuszewski! Do pana nie dociera, że brakuje 400 mln Krakowowi na zorganizowanie tych igrzysk. Pan przyjmuje (Dzwonek) tylko propagandę i tylko to, co jest najważniejsze właśnie dla was, rządzących. Jedno pytanie, panie ministrze: Do kiedy jest ostateczny termin na podpisanie umowy z Krakowem? Wczoraj przedstawiciele Krakowa powiedzieli, że tą ostateczną datą jest 15 stycznia. Czy pan to potwierdza, czy będzie szybciej podpisana umowa? Czy rzeczywiście te igrzyska w Krakowie się odbędą? Bardzo dziękuję. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pana ministra Karola Rabendę o zabranie głosu. Zapraszam, panie ministrze.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Może na początek przypomnę, że mówimy o ustawie o wsparciu organizacji igrzysk, a nie o organizacji igrzysk. Organizatorami tej imprezy są samorządy Krakowa i województwa małopolskiego.

III Igrzyska Europejskie będą pierwszą w Polsce multidyscyplinarną imprezą sportową rozgrywaną na terenie Unii Europejskiej, bo to jest coś, czego jeszcze w Unii nie było. Słusznie tu ktoś zwrócił uwagę, że były poza obszarem europejskim, więc mierzymy się z czymś zupełnie nowym. Rząd polski w swojej uchwale podjął decyzję o wsparciu tej imprezy i to wsparcie będzie realizowane. Powierzenie Polsce organizacji igrzysk stanowi nobilitację i szansę rozwojowa dla regionu, ale też dla całej Polski.

To będzie szansa dla samorządów, jeśli chodzi o sytuację post-COVID-ową, na przywrócenie rozwoju turystycznego. Jesteśmy w rzeczywistości po-COVID-owej, jeszcze nie mamy końca epidemii, ale gospodarka wraca na normalne tory. Wszystkie bodźce, które mają skierować nas na prawidłowe tory rozwoju, są istotne. Projektowana ustawa ma stworzyć warunki umożliwiające właściwą organizację igrzysk oraz wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy host city contract. Konieczne jest zatem opracowanie rozwiązań prawnych zapewniających efektywne działanie organizatorów, czyli samorządów. Kierujecie pytania, które nie są do strony rządowej, bo organizatorami są samorządy. Określenie warunków realizacji przedsięwzięć w zakresie projektowania budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia igrzysk oraz wskazanych podmiotów, które będą mogły je realizować. Określenie sposobu finansowania lub dofinansowania niektórych kosztów organizacji igrzysk oraz przygotowania i realizacji przedsięwzięć. Określenie zasad udzielania i realizacji zamówień publicznych przedmiotom realizującym przedsięwzięcia związane z organizacją igrzysk. Określenie zasad tworzenia i działania spółki celowej oraz warunków umowy o powierzeniu tej spółce realizacji zadań związanych z przygotowaniem igrzysk. Określenie zasad w postępowaniu administracyjnym dotyczącym realizacji przedsięwzięć. O tym jest ta ustawa, ona nie jest o organizacji imprezy, bo rząd nie organizuje tej imprezy, tylko samorząd, a rząd wspiera tę imprezę, tę organizację. Tak jak wspomniałem na początku, ta ustawa powstała we współpracy z samorządami, na ich prośbę. Są tu zapisy, o które one zabiegały, żeby ta impreza mogła się odbyć. Apeluję zwłaszcza do posłów z komisji. Wczoraj przedstawiciele samorządów - za co im dziękuję, za obecność, ale też za współpracę - wyjaśnili państwu, co do tej pory zostało zrobione w kwestii przygotowania igrzysk. Mówienie, że samorządy nic nie zrobiły przez ten okres, jest obrażaniem samorządów. Wiem, że politykę można robić na wszystkim, ale nie róbmy jej na sporcie, na czymś, co służy obywatelom, wszystkim obywatelom, bo te obiekty, które zostaną wyremontowane, zbudowane przy okazji igrzysk olimpijskich, będą służyły mieszkańcom Małopolski, ale też będą służyły promocji sportu, a w dzisiejszym świecie sport jest istotny, biorąc pod uwagę różnego rodzaju problemy z chorobami cywilizacyjnymi itd.

Infrastruktura, która będzie zbudowana, przebudowana, w oczywisty sposób będzie służyła rozwojowi tych dyscyplin.

Tak jak wspomniałem, sport jest czymś, co powinno nas wszystkich łączyć. Wiem, że walka polityczna może być sprowadzona do każdego tematu, ale mówimy o organizacji imprezy, która przyniesie tylko korzyści, nie tylko Małopolsce, nie tylko Krakowowi, ale także całej Polsce. Wczoraj na posiedzeniu komisji byliśmy świadkami naprawdę skandalicznego zachowania. Kiedy wasze pytania zostały sprostowane przez przedstawicieli samorządów, postanowiliście zrywać kworum na posiedzeniu tej komisji. Ale o czym to świadczy? Wy chcecie, żeby ona się nie udała. A tak jak wspominałem wcześniej, organizatorem nie jest rząd polski, tylko samorząd. Szkodzicie samorządowi Krakowa, szkodzicie samorządowi Małopolski takimi zachowaniami nie wszystkich członków opozycji.

No po co? Po co to było? Jeśli nie chcecie pomagać, nie przeszkadzajcie.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie mogę nie zareagować, jeżeli słyszę, że to posłowie PiS-u chcieli wczoraj zerwać posiedzenie komisji albo że posłów PiS-u było za mało. Chciałem powiedzieć, że właśnie większość posłów, którzy wczoraj uczestniczyli w posiedzeniu komisji.

Liczę na to, że również te poprawki, których jeszcze nie zdążyłem przeczytać, do tego dążą - poprawki wszystkich klubów, bo praktycznie rzecz biorąc, wszystkie kluby te poprawki zgłosiły. Natomiast proszę nie mówić takich rzeczy, że to posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości wczoraj zrobili rewoltę, bo to akurat nie ci posłowie.

Zapraszam na posiedzenie komisji. Dziękuję serdecznie. Nie słyszę.

Dziękuję za tę błyskotliwą uwagę. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1631 i 1741) Proszę panią poseł Józefę Szczurek-Żelazko o przedstawienie sprawozdania komisji. A państwu ministrom dziękuję serdecznie za przybycie. Jednych żegnam, a drugich witam. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1631.

Komisja Zdrowia wczoraj rozpatrzyła powyższy projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, co ma zagwarantować skoncentrowanie realizacji działań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej jako państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi zdrowia. Centrum powstanie na bazie połączonych dwóch instytucji, które w tej chwili realizowały podobne zadania, ale w różnych zakresach, tj. Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja w trakcie prac przyjęła 10 poprawek, polegających m.in. na dodaniu do Rady do spraw Zdrowia Publicznego przedstawiciela Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Do tej pory w Radzie do spraw Zdrowia Publicznego pracowali przedstawiciele pozostałych zawodów medycznych, natomiast brakowało w jej składzie przedstawiciela fizjoterapeutów.

W trakcie prac uwzględniono także poprawkę dotyczącą uzupełnienia przepisów części wspólnej projektu o specjalizację w dziedzinie psychoterapii uzależnień. W tej chwili te zapisy będą miały charakter ujednolicający i doprecyzowujący. W trakcie prac pojawiły się inne poprawki, które zostały przez komisję odrzucone, ale zostały zgłoszone jako wnioski mniejszości. Te poprawki dotyczyły m.in. zmian w składzie Rady do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. W projekcie ustawy mamy wpisane instytucje, które mogą delegować do prac w Radzie do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. Natomiast część posłów zgłosiła poprawkę mającą na celu wykreślenie z tego projektu chociażby przedstawicieli poszczególnych ministerstw, a na to miejsce wpisanie przedstawicieli różnych organizacji. Przedstawiono również poprawkę dotyczącą umożliwienia wiceprzewodniczącemu rady zapraszania specjalistów zajmujących się problematyką uzależnień oraz powoływania zespołów roboczych. Chcę zaznaczyć, że przewodniczącym rady jest członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, a wiceprzewodniczącym jest członek kierownictwa innego ministerstwa.

Ta poprawka nie znalazła uznania komisji, ponieważ taki zapis byłby wbrew przepisom ustawy o specjalizacjach, które mogą być realizowane w ochronie zdrowia. Tam dokładnie został unormowany sposób, czy ścieżka, zdobywania specjalizacji w dziedzinach z zakresu ochrony zdrowia. W związku z powyższym komisja po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy na posiedzeniu 15 listopada wnosi, aby Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Zgodnie z regulaminem komisja przedstawia na żądanie wnioskodawców 10 wniosków mniejszości. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę panią poseł Katarzynę Sójkę z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość o zabranie głosu.

Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1631 i 1741. Proponowane zmiany mają na celu utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poprzez połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Projektowane zmiany mają na celu skupienie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w kierunku profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z różnymi rodzajami uzależnień w jednej jednostce organizacyjnej jako państwowej jednostce budżetowej podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Skoncentrowanie działań w jednym podmiocie decyzyjnym, jakim będzie to centrum, pozwoli na połączenie tematyki różnych uzależnień - czynnościowych, chemicznych, uzależnień od substancji legalnych, od substancji nielegalnych - na różnych etapach działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Obecnie funkcjonujące jednostki działają osobno w odniesieniu do problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z pominięciem innych uzależnień, które w tym zakresie pozostają poza regulacjami prawa powszechnie obowiązującego. Aktualnie każda z tych jednostek realizuje swoje zadania ustawowe i zadania „Narodowego programu zdrowia” związane z odrębnymi rodzajami uzależnień, mimo że w wielu przypadkach ich połączenie byłoby zasadne i korzystne, ponieważ oba podmioty realizują zadania o zbliżonym zakresie przedmiotowym. Zadania tych podmiotów odnoszą się wspólnie do profilaktyki, do leczenia uzależnień, do edukacji publicznej oraz wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań dotyczących odpowiednio profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Czynnikiem różnicującym zakres zadań obu tych podmiotów nie są obszary problemowe czy formy oddziaływania społecznego, a jedynie podział na substancje, których używanie powoduje szkody i problemy społeczne. Centrum zajmujące się w sposób kompleksowy problematyką uzależnień umożliwi prowadzenie profilaktyki państwa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w sposób skoordynowany, spójny, co przyczyni się do bardziej skutecznego niż dotychczas osiągania planowanych celów. Wprowadzenie proponowanych zmian zwiększy efektywność działań, zmniejszy obciążenie administracyjne, pozwoli na poprawę obecnie funkcjonującego rozwiązania organizacyjnego i lepsze wykorzystanie środków z budżetu państwa, a przede wszystkim poprawi efektywność prowadzonych działań i zadań. Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość ocenia pozytywnie projekt ustawy i rekomenduje kontynuowanie prac legislacyjnych nad omawianym projektem. Dziękuję bardzo. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w ramach drugiego czytania chciałby złożyć dwie poprawki, które usprawnią ten projekt. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, pan poseł Rajmund Miller, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu KO - PO wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1631 i 1741. Projekt ustawy wprowadza połączenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku tego utworzone zostanie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Celem powołania centrum jest skoncentrowanie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w jednej jednostce organizacyjnej jako państwowej jednostce budżetowej utworzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia. W miejsce Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powołana zostanie Rada do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. W skład rady będą wchodzili przedstawiciele organów i podmiotów, które są obecnie reprezentowane w Radzie do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Zakładane są również zmiany dotyczące ustanawiania wojewódzkich i gminnych programów w zakresie profilaktyki uzależnień. Projekt oddziałuje na Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, populacje osób uzależnionych i współuzależnionych, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Chociaż sama idea połączenia tych instytucji wydaje się uzasadniona, to jednak szczegółowe zapisy zawarte w ustawie budzą poważne zastrzeżenia. Po pierwsze, chodzi o sposób powoływania i skład Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. To nie jest stworzenie merytorycznego ośrodka, a utworzenie kolejnego ciała politycznego, czego zresztą przedstawiciele ministerstwa nie ukrywali, mówiąc o takim celu w czasie posiedzenia komisji, co nas bardzo zdziwiło. Taki polityczny sposób powoływania krajowego centrum budzi poważne wątpliwości co do skuteczności realizacji zakładanych celów. W związku z tym opozycja wspólnie z przedstawicielami strony społecznej złożyła poprawki do ustawy. W miejsce przedstawicieli resortów, które mają najmniej wspólnego z polityką dotyczącą problemów uzależnień, proponuje się wprowadzenie przedstawiciela ministra właściwego do spraw edukacji i nauki, specjalistów w dziedzinie uzależnień, samorządu terytorialnego i przedstawiciela rzecznika praw obywatelskich.

Tam też zostali powołani przedstawiciele na analogicznych zasadach, czyli ciało polityczne.

Obawiamy się, że podobnie będzie wyglądało działanie tego, który dzisiaj zostaje powołany.

Mamy powód do obaw? Jak najbardziej.

Chciałem państwu powiedzieć, że w Polsce jest 290 tys. osób uzależnionych. W przeliczeniu ze współuzależnionymi to 870 tys. osób wymagających takiego leczenia.

Tam mamy jeszcze więcej zastrzeżeń co do tego, o czym mówiła pani minister. Zmusza się osoby, które mają zdany egzamin państwowy, do ponownego zdawania egzaminu państwowego po to, żeby uzyskały stopień specjalizacji. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej - Platformy Obywatelskiej składam 10 poprawek do tej ustawy. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Wysoka Izbo! Rozpoczęliśmy drugą dyskusję na posiedzeniu plenarnym na temat ustawy. Wczoraj Komisja Zdrowia zajmowała się nią przez 3 godziny. Bo oczywiście ustawa w swej istocie polegająca na tym.

Jest tyle zapisów w tym projekcie nawet wewnętrznie niejasnych, nie mówiąc o tym, że niezgodnych z innymi ustawami. Doszło przecież do sytuacji, pani poseł, że po tej 5-minutowej przerwie, która się wydłużyła, zgodnie z propozycją przewodniczącego Latosa, bardzo racjonalną, umówiliśmy się z panem ministrem, że po posiedzeniu komisji, może w nocy, w każdym razie do dzisiaj, przedstawi nam swoje stanowisko. Czy te bałaganiarskie zapisy dotyczące specjalistów, przy okazji także rehabilitacji uzależnień, zostaną, czy będą nowe rozwiązania? Jakoś nie słyszymy, żeby były zmienione, patrzę na pana ministra. Usterek jest wiele. Są to opisowo zachowania o charakterze nałogowym związane z zażywaniem jakiejś substancji, które wiążą się z odczuwaniem przymusu wykonywania określonych czynności i powtarzaniem ich pomimo negatywnego sensu dla siebie i otoczenia, ale w tej ustawie powinna być definicja uzależnienia behawioralnego. Tego typu niejasności jest dużo. Nawet w tej ustawie ta centralizacja zarządzania, to, że wszystko jest w rękach ministra zdrowia, jest wręcz niesmaczna. I z uporem nie pozwalacie, żeby do tej krajowej rady tworzonej przez premiera dokooptować kogoś innego, np. rzecznika praw obywatelskich czy rzecznika praw pacjenta. Mnóstwo rzeczy jest tam albo bałaganiarskich, albo złych.

Chciałbym w imieniu naszego klubu, klubu Lewica, zapytać, jaki jest faktyczny podział środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie uzależnień. Jakie środki konsumowane są przez terenowe placówki specjalistyczne zajmujące się tymi zagadnieniami od strony praktycznej, a w końcu jakie środki wydaje się obecnie oraz jaki będzie łączny budżet wszystkich jednostek centralnych, łącznie z nowo utworzonymi podmiotami? Jednocześnie na ręce pana marszałka chciałbym złożyć w imieniu mojego klubu poprawki do projektu o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, wraz z uzasadnieniem. Od rozpatrzenia tych poprawek warunkujemy nasze głosowanie nad przyjęciem całości projektu tej ustawy. Dziękuję serdecznie. A przedstawiał to stanowisko pan poseł Jan Szopiński. Wysoka Izbo! Pierwotnie wydawało się, że podstawowym celem ustawy jest techniczne połączenie Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i utworzenia jednej, nowej instytucji: Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Warto dodać, że nawet zmiany, które nie dotyczą głównego zakresu projektu ustawy, a które mają charakter teoretycznie porządkujący czy upraszczający określone przepisy, wywołały krytyczną dyskusję np. w środowisku psychoterapeutów. Rządowy projekt ustawy stawia szereg celów, szczególnie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi. Niestety brakuje określenia narzędzi oraz tworzenia jasnych mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie tych celów.

Mam na myśli tutaj przede wszystkim synergię działania kilku resortów, które mają największy wpływ na walkę z uzależnieniami. Bo ustawa, jeżeli już ingeruje w działania samorządów terytorialnych, ich strategię walki z uzależnieniami, to mogłaby, a raczej powinna zacząć od wskazania niezbędnych i obligatoryjnych działań wspólnych poszczególnych ministerstw, a najlepiej określonych działów administracji.

Tego brakuje. Uważam, że tego typu ustawy, z którymi wiele osób, specjalistów w tej dziedzinie, wiąże naprawdę bardzo duże nadzieje, powinny być staranniej przygotowane, powinny określać nowe narzędzia, mechanizmy, nowe sposoby rozwiązywania problemów.

Dziękuję serdecznie. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Omawiamy, wydawałoby się, jeden z najmniej kontrowersyjnych rządowych projektów.

Zasługuje to na uwagę i na to, żeby pozwolić przeprowadzić tego typu działanie. Niewątpliwie są przesłanki, żeby uznać, że jest to dobry pomysł nie tylko ze względów oszczędnościowych, ale także ze względu na kwestie koordynacji i podniesienia rangi w ogóle problemów uzależnień.

Takie jest stanowisko naszego koła, które będzie generalnie popierać te rozwiązania. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Zamykam listę. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Podczas pierwszego czytania tego projektu pytałem o zasadność utworzenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sytuacji, gdy w kraju funkcjonuje obecnie bliźniacza jednostka: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Pytałem również o celowość centralnych instytucji w obszarze zwalczania uzależnień, które w praktyce nie mają żadnego kontaktu z osobami uzależnionymi, a ich działalność polega m.in. na zlecaniu kampanii agencjom reklamowym oraz opracowywaniu sprawozdań uzasadniających ich istnienie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Panie ministrze, proszę odpowiedzieć, dlaczego nie są doprecyzowane zasady współpracy z sądami powszechnymi w sprawach nieletnich i rodzinnych i czy ewentualnie te poprawki zostaną wprowadzone do tego projektu ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W państwie Prawa i Sprawiedliwości, jak wszyscy doskonale wiemy, unika się za wszelką cenę transparentności, jawności i sprawiedliwości. Są to pojęcia, mam nadzieję, znane posłankom i posłom znajdującym się po mojej prawej stronie, jednak zupełnie niepasujące do ich polityki, a pewnie w niektórych przypadkach i do charakteru. Dlaczego o tym mówię? Dla samego pojęcia nie jest istotne to, czy chodzi o sprawę wagi państwowej, czy o usprawnienie życia codziennego Polek i Polaków. Dlatego chciałabym zadać pytanie. Jakie jest wytłumaczenie tego, że dyrektor centrum powoływanego w tej ustawie nie może być wyłaniany w jawnym, rzetelnym konkursie? Czy wszędzie musicie mieć swoich wiernych aparatczyków, którzy służą nie dobru państwa, ale tylko waszym politycznym interesom? Dziękuję serdecznie. Pan poseł Zdzisław Wolski, Lewica. Nowe centrum będzie zajmowało się uzależnieniami. Wiadomo, to jest wielki, bolesny problem, również społeczny, problem osób uzależnionych i ich rodzin, dzieci.

A przecież będą tam dane tzw. wrażliwe, których wypłynięcie może doprowadzić np. do stygmatyzacji dzieci i nie tylko.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym zapytać o kwestię finansowania zadań nowej agencji. Otóż wydawałoby się, że kluczową kwestią jest zwiększenie tego finansowania, nie są zaś wyłącznie czynności, powiedziałbym, administracyjno-techniczne, które w istocie nie przyniosą zbyt wielu korzyści poza, być może, likwidacją części etatów administracyjnych. Chciałbym zapytać o to, dlaczego, z jakich powodów nie przewidziano dodatkowych źródeł, dodatkowych środków finansowych na realizację zadań przez nową agencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mówi się, że od mieszania herbata nie jest słodsza, i to jest prawda. Od mieszania w tym garnku uzależnień też nie będzie lepiej, jak się powoła nową radę i nową agencję.

Nie znajdujemy żadnych merytorycznych wskazówek co do tego, że nowa agencja będzie rozwiązywała także nowe problemy. To bardzo niedobrze. No to po co to wszystko? PARPA działa od lat i działa skutecznie. Tak jak mówią specjaliści, ta ustawa przyniesie nie rozwój, a raczej regres. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze!

Chciałem wobec powyższego zapytać: Kto zawalił, że w ustawie właściwej, czyli w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych z 29 października 2021 r., ta kwestia nie została uregulowana?

Dziękuję. Zapraszam. Kontynuuję wystąpienie pana posła Tomaszewskiego, panie marszałku.

Jesteśmy temu przeciwni, bo jeżeli składacie ustawę, to róbcie to porządnie. Po drugie, pokazaliśmy, że mamy uwagi do tego, tak jak i strona społeczna, w zakresie powołania Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, w stosunku do analogicznie funkcjonującego „Narodowego programu zdrowia”

Jak połączenie obu agencji pozwoli na uzyskanie lepszego efektu walki z uzależnieniami? Bo tego niestety państwo nam nie powiedzieli. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Przez to w ostatnich latach dosyć silnie to zjawisko dawało znać o sobie. W związku z tym mam pytanie: W jaki sposób to połączenie - wydaje mi się, że zbliżenie - zwalczania wszelkich uzależnień właśnie w mniejszych gminach pomoże w zatrzymaniu tego bardzo niekorzystnego zjawiska? Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam podstawowe pytanie dotyczące finansów, ponieważ bardzo dużo mówiliśmy o nowej jakości, jaką ma dać nowa instytucja po połączeniu dwóch poprzednich, ale bardzo mało mówi się o tym, co jest niezwykle ważne przy funkcjonowaniu tego typu mechanizmów, czyli o dodatkowym finansowaniu. Z uzasadnienia i z dyskusji, którą toczyliśmy, wynika, że tak naprawdę będą oszczędności wynikające z połączenia tych dwóch instytucji. Chyba nie tego oczekują ludzie, którzy mają wykonywać te same zadania. Druga sprawa to pytanie o ochronę danych osobowych. To niezwykle ważna kwestia, o którą upominał się w swoich uwagach przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prosiłbym o dodatkowe wyjaśnienie tej kwestii tutaj, z mównicy sejmowej. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W obecnym czasie mamy do czynienia z nasilonym zjawiskiem uzależnień połączonych, współuzależnień. W związku z tym te działania mające na celu profilaktykę dotyczącą tych zjawisk są niezwykle ważne. Te dwie instytucje, które do tej pory działały, prowadziły równolegle pewne działania, mając swoje programy, swoje metody profilaktyki. Chcę również podkreślić, że na poziomie gminy zgodnie z ustawą powstawały dwa programy: profilaktyki uzależnień od alkoholu i profilaktyki uzależnień od narkotyków. W związku z tym połączenie tych instytucji i wprowadzenie nowych regulacji powoduje, że te działania będą skoncentrowane, będą wieloaspektowe, ale koordynowane przez jedną instytucję. To jest niezwykle ważne.

Dziękuję bardzo. Zapraszam podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Macieja Miłkowskiego do zabrania głosu. Czy pani sprawozdawca komisji będzie chciała jeszcze zabrać głos? Pani poseł, tutaj jestem. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, panie ministrze. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo serdecznie za przedstawione stanowiska oraz przedstawione pytania. Po pierwsze, pytanie pana posła Szopińskiego: Dlaczego połączenie i po co formalne? Ponieważ było zapytanie, jeszcze przygotowujemy odpowiedź, która będzie wysłana do pana posła. Wszyscy się zgodzili, że właściwie to jest niby sprawa techniczna, ale jest tu bardzo istotny element, czyli w jednej instytucji zorganizowanie pracy i zadań, które są związane z uzależnieniami.

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie uzależnień zgodnie z koszykiem świadczeń gwarantowanych, który jest określony w ramach koszyka świadczeń psychiatryczno-uzależnieniowych.

Te środki będą wykorzystane.

Wielokrotne padło pytanie, dlaczego nie zostały uwzględnione uwagi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Tak jak powiedziałem, te środki na konkretną realizację zadań już są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i NPZ-etu przedstawione i wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne będą te środki przeznaczane. Widzimy, że jest zasadność kontynuacji wzrostu środków finansowych w tym zakresie, ponieważ mamy problemy z kolejnymi uzależnieniami. Kolejny pilotaż, na razie dla dzieci, które nałogowo używają urządzeń cyfrowych, pilotaż celem zweryfikowania metod leczenia. Planujemy, że po etapie pilotażu to świadczenie wejdzie do świadczeń gwarantowanych, bo widzimy, tak jak mówiłem, problemy z innymi uzależnieniami, w szczególności również cyfrowymi, i to w tej populacji naszych dzieci. Na tym będziemy musieli się skupić.

Mniej osób będzie musiało te zadania realizować, lepiej będą one przygotowywane. W związku z tym uważamy, że lepsze wykorzystanie zasobów, lepsze wykorzystanie i lepsze efekty będą w tym zakresie.

Jeden to ta rada do spraw przeciwdziałania uzależnieniom, skład rady, możliwość kompromisu we współpracy, pomiędzy przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego, co było bardzo istotnym elementem w dyskusji. Tak że z tego, co widzimy, te osoby, które współpracują, które są w radzie, nie mają problemów komunikacyjnych. Nigdy nie zdarzyło się, żeby jakiś wniosek, nie tylko wiceprzewodniczącego, ale też zastępcy czy nawet członka, nie został uwzględniony.

Zresztą ta rada powołuje ciała doradcze, zespoły. Aktualnie jest zespół, jak mówiłem, do spraw reformy lecznictwa uzależnień i ta praca jest na dosyć zaawansowanym etapie. Pan Zdzisław Wolski mówił, że bardzo wiele osób utraci uprawnienia do leczenia osób właśnie z uzależnieniami.

W związku z tym te wszystkie osoby, które są tam wymienione, mogą realizować te przepisy. Ale wiemy, żeby była jasność, żeby to było zagwarantowane w ustawie, wiem, że takie poprawki zostały przedstawione. Ponieważ ten problem był zgłoszony w Komisji Zdrowia, to takie uprawnienia będą nie tylko dla specjalisty psychoterapii uzależnień, ale również dla instruktorów terapii uzależnień, żeby jednakowo potraktować te dwie grupy zawodowe.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Zdrowia w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1731 i 1737) Bardzo proszę pana posła Jerzego Maternę o przedstawienie sprawozdania komisji. A państwu ministrom dziękuję serdecznie za przybycie i zabranie głosu. Proszę bardzo, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1731 i 1737. Pani marszałek Sejmu, zgodnie z regulaminem, skierowała w dniu 8 listopada powyższy projekt do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do pierwszego czytania. W ramach pierwszego czytania posłowie zgłosili trzy poprawki poprawiające funkcjonowanie ustawy. Biuro Legislacyjne zgłosiło poprawkę o charakterze doprecyzowującym ustawę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projektowana ustawa stanowi jeden z elementów tzw. tarczy antykryzysowej wprowadzającej szereg rozwiązań regulacyjnych minimalizujących negatywne skutki dla gospodarki i społeczeństwa w wyniku stanu epidemicznego powstałego na skutek COVID-19. Projekt ustawy wprowadza zmianę do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. poz. 1842, z późn. zm., zwanej dalej ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19, przez dodanie art. 15zzzt, , który umożliwi zachowanie ważności dokumentów marynarskich – dyplom, świadectwo przeszkolenia, świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej – do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. Proponowana zmiana związana z zachowaniem ważności dokumentów marynarskich wynika z pogarszającej się sytuacji marynarzy, którzy z uwagi na ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw mają trudności z powrotem do kraju i nie mogą odnowić dyplomu, świadectw, przeszkolenia lub świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie morskiej albo nie mogą odbyć odpowiedniego szkolenia lub zdać egzaminu niezbędnego do odnowienia dokumentów z uwagi na wprowadzone ograniczenia. Zgodnie z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht muszą one być odnawiane w okresach 5-letnich przez ukończenie przeszkolenia uaktualniającego lub zdanie egzaminu. Szkolenia takie odbywają się w morskich jednostkach edukacyjnych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, MJE, i składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Brak możliwości prowadzenia szkolenia w sposób stacjonarny uniemożliwia przeprowadzenie przeszkolenia przez MJE, a tym samym odnowienie świadectw przez marynarzy. Brak takich świadectw uniemożliwia zaokrętowanie marynarzy na statek i powoduje zerwanie kontraktu za niedopełnienie przez marynarza obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów kwalifikacyjnych.

Prawo telekomunikacyjne, upływa w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 13 marca 2020 r., termin ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. Rekomendowane rozwiązanie uwzględnia wytyczne określone w piśmie okólnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej nr 4204 z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącym wytycznych w zakresie certyfikacji marynarzy i rybaków.

Projekt zawiera propozycję zmian w zakresie spraw przyporządkowanych działowi gospodarka wodna. Zakłada się przejęcie przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zadań w zakresie melioracji od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Przedmiotowa zmiana ma na celu zapewnienie stworzenia spójnego systemu melioracji wodnej zrządzanego przez organ właściwy w sprawach gospodarki wodnej. Melioracja wodna polega na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Działanie to stanowi jeden z sposobów wykorzystania zasobów wodnych. Dlatego też działania podejmowane w obszarze melioracji przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powinny być prowadzone w ścisłej współpracy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, który jest właściwy w sprawach dotyczących izb rolniczych, związków zawodowych rolników i organizacji społeczno-zawodowych rolników, czyli przedstawicieli bezpośrednio zainteresowanych poprawą warunków wodnych na potrzeby rolnictwa.

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Komisja przyjęła projektowaną ustawę bez głosu sprzeciwu. Rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie projektowanej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Otwieram dyskusję. Pan poseł Kacper Płażyński, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Staram się, chociaż jak pan wie, różnie to jest oceniane. Bardzo proszę.

Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Tych zmian jest bardzo wiele. Nie będę powtarzał po pośle sprawozdawcy, ale podobnie jak pozostali członkowie komisji gospodarki morskiej, rekomenduję w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwość głosowanie za tym projektem.

Są ważne gesty i ta ustawa jest jednym z nich, wychodzi naprzeciw bardzo wielu potrzebom społecznym i ekonomicznym w tym dla nas w dalszym ciągu niełatwym czasie post-COVID-owym czy COVID-owym.

Pozwolę je sobie od pana odebrać, panie pośle. Pan poseł Tadeusz Aziewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jak już wspomniano, ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz niektórych innych ustaw jest jednym z elementów tzw. tarczy antykryzysowej, która wprowadza rozwiązania regulacyjne minimalizujące negatywne skutki powstałe w wyniku stanu epidemicznego wywołanego COVID-19. Proponowane rozwiązania dotyczą przedłużenia ważności dokumentów marynarskich, które z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii nie mogły być odnowione w obowiązujących terminach, dotacji dla Agencji Żeglugi Powietrznej - chodzi tu o zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID, m.in. operacji bezzałogowych statków powietrznych - wsparcia finansowego dla pasażerskich przewoźników kolejowych, przejęcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej zadań z zakresu melioracji od ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Tutaj chciałem tylko podkreślić, że opozycja zasadniczo nie chce ingerować w podział kompetencji pomiędzy resortami, będziemy oceniać rząd za efekty, natomiast wieść gminna niesie, że poprawki, które zostały złożone przez pana posła Płażyńskiego, niejako odwracają rozwiązanie, które zostało przyjęte na forum komisji. Myślę, że jutro na kolejnym posiedzeniu komisji wyjaśnimy to do końca. Propozycje zmian dotyczą także odroczenia w czasie wejścia w życie zmian w systemie opłat za usługi wodne zakładających wprowadzenie uzależniania wysokości opłaty stałej za usługi wodne, za pobór wód podziemnych oraz wód powierzchniowych od dostępności zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia. Według projektodawców z powodu pandemii nie udało się zebrać z terenu danych niezbędnych do wyliczeń, co kwestionuje w materiale przesłanym wysokiej komisji Związek Powiatów Polskich. Dalej propozycje zmian dotyczą zmiany terminu zachowania mocy aktualnie obowiązujących planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, zwolnienia z obowiązku wnoszenia należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych, dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na przewozie ładunków, pasażerów i wykonywaniu prac technicznych oraz osób fizycznych uprawiających żeglugę śródlądową na drogach wodnych. Rząd proponuje także przekazanie spółce Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście skarbowych papierów wartościowych w wysokości 360 mln zł. Proponuje wsparcie organów prowadzących jednostki systemu oświaty w zakresie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wysoki Sejmie!

Poprawki te były konsekwencją proponowanych rozwiązań. W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej rekomenduję przyjęcie tego projektu. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam, panie pośle. Czekamy z panią sekretarz z niecierpliwością na ten głos. Panie Marszałku! Panie Ministrze! W imieniu klubu Lewicy mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec tego projektu ustawy, projektu zmieniającego w sumie sześć ustaw obowiązujących w naszym kraju. Można powiedzieć, że pierwsza generalna uwaga jest taka, że mamy wrażenie, że dzisiaj COVID jest wykorzystywany przez polski rząd nie do poprawiania polskiego prawa, ale raczej do psucia polskiego prawa. Mamy wrażenie, że chodzi tutaj o to, że rozsyłana jest po ministerstwach informacja, że szykujemy zmianę ustaw COVID-owych z 2 marca, z 30 marca, co tam macie w tych ministerstwach, to może jeszcze wrzucimy do jednego projektu ustawy i będziemy nad tym spokojnie procedować.

Tak jak wspomniałem, wrzucacie państwo tutaj kilka spraw, z których jedne nie budzą kontrowersji, ale kilka niestety te kontrowersje budzi. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z bezpieczeństwem morskim, pewnie to jest powód. Pewnie dlatego, że ktoś przeczytał pierwszy punkt, a tam rzeczywiście jest kwestia dotycząca przesunięcia terminów ważności tych wszystkich uprawnień, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo morskie. Pewnie dlatego trafiło to do naszej komisji. Ale co Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma wspólnego z działami administracji rządowej i z waszymi problemami w rządzie, żeby się dogadać, to tego nie wiem.

Jeżeli chodzi o ustawę - Prawo wodne, to ewidentnie znowu mamy do czynienia z funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa, czyli Wód Polskich, które nie zdążyło wykonać wszystkich zadań, oczywiście po części przez COVID, ale niestety po części też przez takie, a nie inne zarządzanie. Dzisiaj przesuwamy to wszystko do 2023 r., powodując, że opłaty za wodę będą dużo wyższe, niż wynikałoby to z obecnie obowiązującego prawa, od roku 2022. Uśmiecham się do pana ministra, ale z drugiej strony rodzi się pytanie, po co to wszystko znowu tak psuć, w sensie prawodawstwa. Wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Znowu idzie to poza budżetem, a przecież pan minister wie i ja doskonale wiem, że te 360 mln zł nie mają nic wspólnego z COVID-em, bo to jest po prostu inwestycja w rozbudowę portów, która rzeczywiście jest bardzo potrzebna i powinna być, ale znajduje się w ustawie COVID-owej. Oczywiście to jest kwestia dotycząca przesunięcia terminów i pewnie bardzo dobrze, że tak się stało, ale pomoc dla szkół za granicą znowu znajduje się w ustawie COVID-owej. Rozumiem, że trzeba pomagać szkołom zagranicznym, które prowadzą naukę w języku polskim, ale od tego jest inna ustawa i można to było zmienić normalną ścieżką, a nie ścieżką COVID-ową.

Dziękujemy za tę zapowiedź. Pan poseł Marek Sawicki, Koalicja Polska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zabierając głos w imieniu klubu Koalicji Polskiej, oczywiście tak jak przy ustawach dotyczących chociażby stanu wyjątkowego czy przy wcześniejszych ustawach COVID-owych, nie będziemy przeszkadzać rządowi w realizacji jego zadań.

W tej chwili odgrzebano je i próbuje się uczynić zadość w związku z kryzysem COVID-owym.

Z jednej strony - powiem to szczerze - gratuluję panu siły. Jako wiceminister pokonał pan w tym rządzie nowo powołanego wicepremiera, ministra rolnictwa Kowalczyka. Co ciekawe, pytałem dzisiaj pana premiera, czy to było uzgodnione i czy on jest świadom, że sprawa melioracji przechodzi do ministra infrastruktury. Był zdziwiony i powiedział, że jeszcze do wieczora to wyjaśni.

Dobrze, że nie odświeżyliście ponownie swojego projektu dotyczącego łamania prawa w imię walki z COVID-19 i niekarania za to.

Znalazłem w projekcie też odniesienia właśnie do melioracji, do ruchu lotniczego - ciekawe rzeczy jak na tak krótką ustawę.

A jednak trochę nasz, więc się tym interesujemy.

Szanowni państwo, to nie jest poważne procedowanie, ale skoro tak, to wy weźmiecie za to odpowiedzialność. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Uprzejmie dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Szanowni Państwo! Ten projekt ustawy zawiera szereg zmian, które można podzielić w zasadzie na takie trzy duże grupy. Pierwsza grupa dotyczy w naszej ocenie rzeczywiście potrzebnych zmian. Do tych zmian, które są potrzebne, możemy zaliczyć np. kwestie związane z przedłużeniem terminu ważności dokumentów marynarskich.

W związku z tym wyjście naprzeciw oczekiwaniom marynarzy jest jak najbardziej zasadne. Do takich zmian, które oceniamy pozytywnie, na pewno można zaliczyć przedłużenie do końca tego roku okresu, za który mogą być przekazywane rekompensaty za świadczenie zleconych przez organizatorów usług publicznego transportu zbiorowego ze środków budżetu państwa przewidzianych na honorowanie ustawowych uprawnień do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

To są takie zmiany, które można uznać za zasadne. Wśród tych zmian, które uznajemy za zasadne, jest też część zmian, które wynikają z potrzeby naprawienia błędów, które popełnił rząd i większość parlamentarna na etapie legislacyjnym, czyli w parlamencie. Tu widzimy, że przepychanie przepisów kolanem się mści. Okazało się, że przepisy przepchnięte przez rząd i przez większość skutkują tym, że PAŻP nie może otrzymać tego dofinansowania. Oczywiście jest to konieczne, natomiast pokazuje ten bezład w działaniach większości. Zresztą podobnie jest, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy. Oczywiście częściowo (Dzwonek) to nie zostało zrobione z powodu warunków COVID-owych, ale w dużej części jest to wynik nieudolności resortu.

To jest coś, co wykracza poza ramy, powiedziałbym, COVID-owe, zresztą podobnie jak zmiana dotycząca przejęcia. Już kończę, panie marszałku. spraw z zakresu melioracji. Nie wiemy, co będzie w poprawkach, które zostały zgłoszone przez większość rządzącą, w związku z czym na temat tego projektu wypowiemy się, po przeanalizowaniu tych poprawek, w głosowaniu. Dziękuję serdecznie, dziękuję. Proszę państwa, otwieram listę pytań. Dziewięć osób się zgłosiło. Zamykam tę listę w związku z tym. Poproszę pana posła Jana Szopińskiego z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy dotyczy rozwiązywania spraw związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zaczynam się zastanawiać, do kiedy rząd będzie w ustawę dotyczącą zwalczania COVID-u wrzucał wszystko, natomiast nie będzie tego realizował w normalnie pojmowanych ustawach. Bardzo proszę o pisemną odpowiedź na pytanie: Jaki związek mają proponowane zmiany z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19? Chodzi zwłaszcza o zmiany, które są w ustawie, a które mówią, że podstawą potwierdzenia poniesionych kosztów w obrocie gospodarczym może być oświadczenie. Pan poseł Rafał Adamczyk, klub parlamentarny Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projekt dotyczy umożliwienia zaokrętowania marynarzy na statek, którzy za względu na stan epidemii mają trudności z powrotem do kraju, oraz odnowienia im posiadanych dokumentów i utrzymania ważności dokumentów marynarskich do dnia upływu 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Panie Ministrze! Proszę o informację, ile jest takich przypadków, które przytoczyłem wcześniej, z uwagi na to, że ten zapis znalazł się projekcie ustawy. Dziękuję i proszę o pisemną odpowiedź. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jego celem, jak wiemy, jest wsparcie z jednej strony rodzin, z drugiej strony firm pokrzywdzonych przez pandemię COVID. Natomiast chciałbym w związku z tym zapytać, po pierwsze, jaki jest obecnie stopień wykorzystania tych bonów, ile się udało wykorzystać, po drugie, ile przedsiębiorstw do tej pory skorzystało z bonu turystycznego. Ponieważ, przypomnę, w zeszłym roku w zimie branża narciarska, kurorty górskie napotkały dosyć duże problemy ze względu na to, że z jednej strony nie było przygotowanych wytycznych, zamykaliście, otwieraliście stoki. W związku z tym może warto by przedłużyć to jednak o cały pełny rok, tak żeby branża, która w zeszłym roku dosyć mocno ucierpiała, w tej chwili mogła się jeszcze bardziej w odkuć sezonie zimowym. A skoro już jestem przy branży zimowej, narciarskiej, to chciałem spytać, kiedy będą jakieś wytyczne odnośnie do obostrzeń na stokach, bo z jednej strony bardzo fajnie (Dzwonek), że stoki będą mogły być otwarte, ale z drugiej strony dobrze by było wiedzieć, i branża o to już dopytuje, czy będzie jakiś reżim sanitarny. Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałem zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza dotyczy bonu turystycznego. Chciałem zapytać, ponieważ jest to kolejne przedłużenie, z jakich powodów rząd upiera się przy tym, że te bony, że te środki muszą być ograniczone w czasie? Wydaje się, myślę, że wszyscy, którzy mieszkamy w regionach turystycznych, zdajemy sobie sprawę, że epidemia odcisnęła bardzo poważne piętno na przedsiębiorcach, na wielu firmach: wiele firm upadło, wiele firm nadal przeżywa kłopoty.

Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Mam pytanie do pana ministra Gróbarczyka, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą inwestycji w morskim porcie Szczecin-Świnoujście, a konkretnie inwestycji dotyczącej portu kontenerowego w Świnoujściu. Jest wpisana kwota 360 mln zł, więc pytanie jest takie, czy to jest kwota, która już została zweryfikowana w kontekście rosnącej inflacji, kosztów budowy. Czy została zweryfikowana i czy to jest kwota, która uwzględnia te wszystkie czynniki zewnętrzne? Rzecz druga, jeżeli chodzi o tę inwestycję, o port kontenerowy: rok czy 2 lata temu były duże napięcia społeczne, jeżeli chodzi o samo miasto Świnoujście i mieszkańców Świnoujścia, w związku z czym moje pytanie jest takie, czy w tej sprawie z władzami Świnoujścia jest już porozumienie i czy wszystkie szczegóły dotyczące budowy portu kontenerowego są uzgodnione z prezydentem i Radą (Dzwonek) Miasta Świnoujście. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dobromir Sośnierz, koło Konfederacja. Zapraszam, panie pośle.

Pan minister Dworczyk nawet chciał się na to zgodzić, żeby po pół roku ponownie te wszystkie przepisy przemyśleć i uchwalić w normalnym trybie, z konsultacjami, ze wszystkim.

To, jeśli ma sens, żeby miały termin ważności (Dzwonek), to po co je przedłużać? Domagamy się uchylenia tej ustawy w całości. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski z Klubu Parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Wody Polskie ustalają wysokość opłat za usługi wodne, nie uwzględniając średniego niskiego przepływu z wielolecia. Wczoraj na łamach „Rzeczypospolitej”

Były trzykrotnie wyższe niż w kolejnym kraju, jakim była Rumunia. W związku z powyższym czy te przepisy, czy niewykonanie tych pomiarów będzie miało wpływ na wzrost cen wody (Dzwonek) dla odbiorców indywidualnych? Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Czasami w stercie śmieci można znaleźć małą perełkę albo diamencik.

Panie ministrze, czy my - bo wiemy, że jak się robi biznes, to trzeba pozyskać pieniądze, a później dobrze je wydać, to jest najważniejsze - mamy zrobiony jakiś biznesplan? Czy jest jakiś biznesplan, czy dopiero będziemy go robili i dopiero będziemy szukali wykonawcy? To jest dla mnie ważne.

Dziękuję, panie pośle, za te perełki i diamenciki. które postara się pozbierać sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Marek Gróbarczyk. Zapraszam serdecznie. Panie Marszałku! Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować państwu za wszystkie uwagi, te konstruktywne oraz te niekonstruktywne. One mają bardzo duże znaczenie w ostatecznym kształcie, ponieważ większość tej Izby popiera tę ustawę, za co państwu bardzo serdecznie dziękuję.

Jeśli chodzi o pytania, które państwo zadaliście, to pierwszym, podstawowym jest to przewijające się przez Izbę, kierowane przede wszystkim przez pana posła Wieczorka, który z jednej strony te rozwiązania popiera, a z drugiej strony ich nie popiera.

Dlatego w takim trybie, bo w innym nie moglibyśmy. W związku z tym, że Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie nr 651, dotyczące właśnie przeciwdziałania skutkom COVID, umożliwiające emisję obligacji w ramach budżetu państwa, skorzystaliśmy z tej okazji i przygotowaliśmy rozwiązanie, które wsparło tak port w Gdyni w zeszłym roku, jak i port w Szczecinie, który już dostał 328 mln. Natomiast aby dokończyć falochron - bo cena tego falochronu będzie oscylowała w granicach 700 mln - kolejne 360 mln zostało przygotowane w ramach obligacji właśnie poprzez tę ustawę.

Potrzeba realizacji terminala kontenerowego - tego już nie będę tłumaczył, panie pośle. Dziękuję bardzo w takim razie.

Oceniamy, że ok. 30 tys. marynarzy jest narodowości polskiej.

A to umożliwia właśnie ta ustawa - przedłużenie tych uprawnień. Oczywiście nowelizacja Prawa wodnego nie ma nic wspólnego z cenami wody. Ceny wody są ustalane przez samorządy i akceptowane przez Wody Polskie. Wody Polskie jako regulator nie dopuszczają do wzrostu cen wody ponad ustawowe rozwiązania. Więc pragnę zapewnić, że nie będzie miało to żadnego wpływu na wzrost cen wody. Na resztę pytań, na które nie odpowiedziałem, pozwolę sobie odpowiedzieć na piśmie. Dziękuję bardzo. Zarzucił pan polski Sejm perełkami i diamencikami. Pomykamy dalej. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 1736. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1681 i 1740) Bardzo proszę pana posła Zdzisława Sipierę o przedstawienie sprawozdania komisji. Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Marszałek Sejmu skierowała powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania, które odbyło się w dniu wczorajszym, czyli 15 listopada. Cała ustawa zawiera tylko albo aż 17 artykułów, natomiast niektóre są bardzo rozbudowane.

Mam nadzieję, że również podczas drugiego czytania - były takie zapowiedzi - będą zgłoszone wnioski do pana marszałka. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Pan poseł Piotr Kaleta z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałby powiedzieć kilka słów. Proszę bardzo, panie pośle.

Pragnę także podkreślić, że jest to ustawa nam w tej chwili niezwykle potrzebna, która powinna jak najszybciej zostać wdrożona do polskiego systemu prawnego. Tak, to są rzeczy, których powinniśmy dokonać w pierwszej kolejności, jak najszybciej. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że odbywa się posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zostało przerwane, byśmy mogli zabrać głos w imieniu komisji, w imieniu klubu, a dotyczy ono również sytuacji na polskiej granicy. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Proszę, Piotrze. Miło cię widzieć. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koalicji Obywatelskiej chciałbym wyrazić opinię w sprawie ustawy, która jest niezwykle istotna.

Rekordziści czekają czasem kilka lat, nawet 5 lat, na wydanie stosownych decyzji. Obiektywnie sprawa jest trudna.

Dlatego ta ustawa zmierza w dobrym kierunku, starano się zrobić wszystko, aby pomóc wszystkim tym, którzy chcą pracować w Polsce.

W związku z tym polscy pracodawcy powinni mieć w dużej części ogrom ułatwień wynikających ze stosownych decyzji dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium naszego kraju, w tym szczególnie na pobyt czasowy i pracę.

Będziemy mieli tylko stosowną uwagę, aby zachować proporcjonalność, bo w przedmiotowym art. 114 pkt 5 mówi się o wysokości minimalnego wynagrodzenia niezależnie od czasu i wymiaru pracy.

Wiemy, że ustawa porządkuje szereg innych elementów wynikających z uznania wyroków Trybunału Sprawiedliwości, także w kontekście dyrektywy o łączeniu rodzin, kwestii małoletności.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Wiesław Szczepański, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. W imieniu klubu parlamentarnego Lewica mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Polska od lat mierzy się z trudną sytuacją demograficzną, a problem ten może narastać w następnych latach. Obecnie brak odpowiedniej liczby pracowników na rynku pracy sprawia, że nasza gospodarka potrzebuje wsparcia cudzoziemców. Uważamy, że polska polityka imigracyjna winna opierać się na systemie kwotowym i przewidywać łatwą ścieżkę nabywania tytułu do stałego pobytu oraz legalnego zatrudnienia.

Wypełniają oni braki na rynku pracy, przyczyniają się do wzrostu PKB oraz wpłat do systemu ubezpieczeń społecznych. Niestety wydaje się, że Polska kopiuje model niemiecki, francuski z lat 50. i 60., gdy państwa zachodnie korzystały z pracy cudzoziemców bez osiedlania ich u siebie na stałe, czyli stosowały tzw. model gastarbeiterski. Możemy za to zapłacić w przyszłości.

Rząd, dostrzegając problemy przedsiębiorców, a jednocześnie starając się wesprzeć ich w uzupełnieniu braków kadrowych pracownikami ze Wschodu, przedłożył zmianę ustawy o cudzoziemcach. Obecnie polskie firmy mogą ściągać na uproszczonych zasadach pracowników z dawnego Związku Radzieckiego, z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, ale tylko na okres 6 miesięcy. Okres ten zostanie wydłużony do 2 lat.

Ma to odciążyć pracę urzędów wojewódzkich.

Uchylony zostanie wymóg przedstawiania przez cudzoziemca adresu zamieszkania w Polsce jako koniecznego do wydania zezwolenia na pobyt i pracę w naszym kraju. Nowela zawiera także przepis mówiący o tym, że obcokrajowiec będzie musiał otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie bez względu na etat pracy, na jakim jest zatrudniony. Ustawa znosi tryb modyfikacji zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonanie pracy. Zezwolenie to nie będzie określało podmiotu powierzającego wykonanie pracy ani warunków jej wykonywania. Te zostaną określone po dostarczeniu decyzji o udzieleniu zezwolenia przez cudzoziemca, który złoży do wojewody oświadczenie przedsiębiorcy powierzającego mu pracę. Poszerzony zostaje katalog okoliczności, które nie wymagają zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Podmioty o szczególnym znaczeniu strategicznym dla naszej gospodarki szybciej uzyskają zezwolenie na pracę i pobyt czasowy cudzoziemca. Zniknąć ma 12-miesięczny okres rozliczeniowy, co umożliwi przedłużenie pracownikowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. W myśl nowelizacji obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego zostanie uznany za spełniony, gdy będzie wynikał z zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Przedsiębiorcy liczą na to, że ministerstwo rodziny skorzysta po zmianach z możliwości rozszerzenia listy państw, z których można ściągnąć tych pracowników, czy też określi zasady, dzięki którym będzie można skorzystać z uproszczonej procedury przy ściąganiu specjalistów do Polski. Mój klub popiera przyjęte rozwiązania, przy czym składa jedną poprawkę. Chcieliśmy również zwrócić, panie ministrze, uwagę na fakt, iż jednak bardzo wiele wiz nie jest (Dzwonek) wydawanych m.in. dla Hindusów czy Nepalczyków. Prosimy o jakieś rozwiązania dla tych osób, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które czekają na to, żeby w Polsce znaleźć pracę. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję za poprawkę. Zapraszam pana posła Marka Biernackiego, Klub Parlamentarny Koalicja Polska. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Klub popiera ten projekt, ponieważ nowelizacja ta zawiera uproszczenia dotyczące prowadzenia postępowań administracyjnych, jeśli chodzi o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce, w szczególności w przypadku łącznych zezwoleń na pobyt i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy.

Wprowadzono natomiast wymóg otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Możliwe będzie przyspieszenie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemcom zamierzającym wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Polski. Projekt ustawy jest dla nas o tyle istotny, że był oczekiwany przez pracodawców, polskich przedsiębiorców. Polscy pracodawcy od lat zwracali uwagę na to, że zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym wymaganiom rynku pracy jest czynnikiem zapewniającym możliwość rozwoju poszczególnych podmiotów gospodarczych oraz regionów Polski. Niedobory rąk do pracy odczuwalne są szczególnie w branży teleinformatycznej, handlu, produkcji czy budownictwie.

I tak wprowadzenie rozwiązań, zgodnie z którymi wymiana informacji między wojewodą lub szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informację, czy wjazd cudzoziemcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jest bardzo istotne, bo służby zawsze lubią robić wszystko na papierze, co bardzo wydłuża bieg, a komunikacja elektroniczna spowoduje, że będzie to odbywało się o wiele sprawniej i skuteczniej. Mając na uwadze podstawowe cele, jakie przyświecają projektowi ustawy, należy pamiętać, że szybsze dopuszczenie cudzoziemców do polskiego rynku pracy może nastąpić tylko w przypadku wzmocnienia służb konsularnych na wschodzie Europy, tj. na Białorusi i na Ukrainie. Tak jak mówiłem, Koalicja Polska popiera ten projekt. Dziękuję, panie pośle, panie ministrze. Zapraszam pana posła Dobromira Sośnierza, koło Konfederacja.

Są więc płatnikami netto do naszego budżetu, ale taki stan nie będzie trwał wiecznie.

Zamiast doraźnego zapychania dziury zajmijmy się więc tym, co działa w długiej perspektywie, czyli demontażem socjalizmu. Jeśli chodzi o doraźne rozwiązania, to trzeba też jednak podkreślić, że potrzebujemy imigrantów do pracy, ale nie wszystkich w takim samym stopniu. Emigracja emigracji nierówna. Należy to w końcu wyraźnie rozgraniczyć. Nie chcemy np. dziczy, która rzuca w naszych żołnierzy kamieniami. Nie chcemy ludzi, którzy, jak pokazują doświadczenia innych krajów, sprawiają potem problemy. Nie chcemy ludzi, którzy się nie asymilują, tylko budują islamskie dzielnice. Boimy się islamistów, nawet jeśli przychodzą z darami. Ułatwienia należy adresować do europejskiej imigracji bliskiej nam kulturowo. W przyszłości może będą to uciekinierzy z kalifatu nadreńskiego czy Australii zamieniającej się właśnie w groteskową despocję maseczkową. Uczmy się na cudzych błędach. Wysoka Izbo! W ostatnich latach bez żadnej debaty politycznej, bez żadnej fundamentalnej debaty w tym parlamencie de facto zmienia się strukturę społeczną, narodowościową Polski.

Wy oczywiście robicie - nieudolnie - wszystko, żeby powstrzymać tych na granicy, ale z drugiej strony fundujecie nam dokładnie tę samą perspektywę jak w Europie Zachodniej. Dlaczego?

Dziękuję serdecznie, panie pośle. Pan poseł Tomasz Zimoch, koło Polska 2050. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Polska 2050 lubi usprawnienia, dlatego popieramy usprawnienie postepowań dotyczących cudzoziemców, dlatego popieramy tę potrzebną ustawę. Uważamy, że można by procedować nad nią w trybie mini-max, czyli minimum słów, maksimum dobrego, koniecznego prawa. W uzasadnieniu czytamy: składanych jest coraz więcej wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych na terytorium Polski, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, dlatego że istnieje potrzeba dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, jak również ułatwienie pozyskiwania przez inwestorów strategicznych pracowników z zagranicy. Cytat z uzasadnienia. Cieszy, że ustawa powstała też po to, by wdrożyć orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cieszy dlatego, bo instytucja ta jest ostatnio przez obóz rządzący bardzo często lekceważona. To świadczy o pośpiechu i niestety o prawniczym niechlujstwie. Wydaje mi się, że ta ustawa przechodzi niezauważona, bo o cudzoziemcach mówi się ostatnio z zupełnie innego powodu. Wysoki Sejmie! Składam podziękowania z tej sali plenarnej dla polskich żołnierzy, policjantów, Straży Granicznej. Chcę wyrazić też słowa wielkiego uznania dla Grupy Granica i wchodzących w jej skład stowarzyszeń.

Ratunek przynosili również medycy na granicy. Przed wami także, drodzy ratownicy, lekarze, czapki z głów.

Dziękuję serdecznie. Do pytań zgłosiło się 11 osób. Ustalam czas na pytanie - 1 minuta. Zapraszam pana Jana Szopińskiego, posła z klubu parlamentarnego Lewica. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z dużym zadowoleniem należy przyjąć proponowane zmiany. Krajowy rynek pracy został umiędzynarodowiony, podobnie jak dzieje się to we wszystkich krajach rozwiniętych na całym świecie. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie polskiej gospodarki bez pracowników pochodzących z innych krajów. Dobrze, że rząd widzi konieczność dostosowania prawa do realiów gospodarczych. Czy faktycznie system administracyjny w naszym kraju, który podobno jest jednym z najlepiej funkcjonujących w Europie, potrzebuje aż 60 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku cudzoziemca o pobyt czasowy? Czy przepisy muszą wymuszać na pracodawcach stosowanie rotacji wśród zatrudnianych cudzoziemców? To ostatnie pytanie jest szczególnie ważne w przypadku pracowników przechodzących często kosztowne szkolenie. No i wreszcie czy urzędy nie muszą pomiędzy sobą wymieniać dokumentów w formie elektronicznej, a tylko mogą? Ja uważam, że powinny i muszą. Dziękuję bardzo. Poproszę, panie ministrze, o odpowiedź na piśmie. Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt dotyczy usprawnienia postępowań w sprawie udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce. Bardzo bym prosił o informację: Czy jest pan przekonany co do tego, że termin rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwoleń na ten pobyt będzie dotrzymany przez poszczególne instytucje? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Cudzoziemcy, którym kończy się pozwolenie na pracę, muszą na nowo o nie występować lub występować o jego przedłużenie. A więc mam pytanie: Czy rozważacie państwo automatyczne przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca, gdy pracodawca nie zmienił umowy o pracę i warunków, a cudzoziemiec nie ulega żadnym pokusom i pracuje bardzo dobrze? Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Chciałem zapytać o branżę transportową. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której brak osób wykonujących zawód kierowcy jest miejscami potężną barierą dla rozwoju i funkcjonowania tej branży. Chciałem zapytać, czy przedmiotowe przepisy poprawią sytuację i o ile może wzrosnąć ilość osób z zagranicy, które będą mogły wykonywać pracę kierowcy w naszych, polskich firmach. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Franciszek Sterczewski. Nie ma pana posła. Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska.

Trzeba przyznać, że branża, szczególnie gospodarka czekała na tę ustawę, bo brakuje w Polsce rąk do pracy i głów do pracy, i to prawie 2 czy ponad 2,5 mln.

I bardzo dobrze, że ta ustawa jest, bardzo dobrze, że daje możliwości, żeby ci ludzie przyjeżdżali. Zauważyłem, że ta ustawa troszeczkę przechyliła szalę. Ona daje możliwości pracownikom, którzy przyjeżdżają, daje im podstawową pensję, niezależnie od tego, kto przyjedzie - może się okazać, że przyjedzie leser, który nic nie umie, i trzeba mu płacić podstawową pensję - daje możliwość przyjechania, wyboru pracodawcy, daje możliwość niepodawania adresu, gdzie jadą. Ale panowie rządzący, my tworzymy prawo dla obywateli polskich, dla przedsiębiorców polskich, dla tych, którzy tutaj tworzą PKB. A więc proszę, żebyście o tym pamiętali, tworząc takie przepisy, i żeby w tych przepisach też ulżyć przedsiębiorcom polskim. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Szanowny Panie Ministrze! Same rozwiązania ustawy idą w dobrym kierunku, bo polski rynek pracy potrzebuje również cudzoziemców, a skrócenie tych wszystkich procedur administracyjnych zapewne poprawi sytuację, w szczególności w newralgicznych miesiącach, kiedy potrzeba rąk do pracy w rolnictwie. Ale chciałbym zapytać o jedną sprawę, mianowicie o przeszkodę w źle działającym systemie informatycznym.

Mimo że pracodawcy zapewniają, że mają stosowne zezwolenie, i zapewniają stanowiska pracy, to tam trzeba czekać w kolejce prawie 8 miesięcy. Czy braki kadrowe, czy inne przeszkody (Dzwonek), które powodują taki długi okres oczekiwania? Dziękuję. Pani poseł Katarzyna Maria Piekarska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Niewątpliwie to jest ustawa, która była od dawna oczekiwana przez polskich przedsiębiorców.

Mam zatem dwa pytania, które się z tym wiążą.

Bo jeżeli ten pracownik ma być dłużej i ma być dobrym pracownikiem, to na pewno będzie lepszym pracownikiem, jeśli będzie miał przy sobie rodzinę. Czy szkoły są na to przygotowane?

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cóż, rozmawiamy o ustawie, która ma po raz kolejny uprościć też życie cudzoziemcom w Polsce. Nie mówię o tym, że mamy jakoś specjalnie je utrudniać, ale chociaż zachowajmy pewne standardy. Rezygnacja z wymogu dotyczącego zamieszkania, jeśli ktoś ma mieć przedłużony pobyt, to nie jest rzecz, która prowadzi do stabilniej i odpowiedzialnej migracji. Państwa partia wygrała wybory w 2015 r. m.in. dlatego, że mówiliście o tym, że będziecie prowadzić odpowiedzialną politykę migracyjną, a ja mam wrażenie, że upraszczanie tych przepisów w tym momencie to jest takie zamykanie oczu, wpuszczanie wszystkich jak leci i zero odpowiedzialności za to, co może się wydarzyć w przyszłości. Na to nie będzie naszej zgodny. Nie przekonuje mnie także fakt mówiący o problemie (Dzwonek) dotyczącym emerytur, ponieważ już dziś mamy sytuację, w której np. Ukraińcy mogą pobierać emerytury, mają prawo do emerytury nawet po przepracowaniu bardzo krótkiego czasu, więc mogą zarabiać tutaj i wyjechać. Nie ma na to naszej zgody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałem zapytać o osoby, które przyjeżdżają do pracy do rolników.

Obecnie duża część pracowników, którzy przyjeżdżają do tego typu pracy, w ogóle u rolnika się nie pojawia.

Oni przechodzą do innych branż. Czy w związku z tymi zmianami ta sytuacja przypadkiem się nie pogorszy?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana ministra Bartosza Grodeckiego o odpowiedź na pytania.

Bardzo dziękuję, pani marszałek. Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Może spróbuję odpowiedzieć na nie po kolei. Pytanie pana posła Adamczyka, jeśli chodzi o terminy. Według nas poprawka dotycząca terminów jest poprawką, która te terminy przede wszystkim urealnia. Pamiętajcie państwo, że to jest do 60 dni, to nie jest tak, że w 60. dniu wojewoda taką decyzję podejmuje.

A więc ten termin urealniliśmy, natomiast to nie jest tak, że to będzie trwało 60 dni. Dziękuję za nie. Nie, nie rozważamy takiej zmiany, ponieważ to by zakładało, że musielibyśmy przyjmować, że każda osoba, która pracuje np. 2 lata u danego pracodawcy, dalej będzie u tego pracodawcy pracowała. Tego nie wiemy, bo być może zmieni pracę na lepszą albo w ogóle wyjedzie z Polski.

To tak jak z wizą. Wizę też się dostaje na określony czas i ona nie zostaje automatycznie przedłużona. bo musielibyśmy taką wiedzą skądś powziąć, a to wymagałoby poinformowania urzędu, czyli wydania tak czy owak jakiegoś zaświadczenia w tym zakresie.

Pytanie pana posła Tomaszewskiego, jeśli chodzi o Indie. MSZ pracował z nami przy tej ustawie.

Jeżeli szkoła przyjmuje do siebie na studia studentów z Indii, przeprowadza wywiady na Skypie, niejednokrotnie nie wiedząc, z kim ma do czynienia, bo ta osoba z drugiej strony legitymuje się jakimś dokumentem, którego dobrze na Skypie nie widać, i podaje się za jakąś osobę, a później ta osoba składa wniosek w konsulacie, przychodzi i nie jest w stanie powiedzieć słowa po angielsku, a jedzie na studia, które będą prowadzone w języku angielskim, to konsul musi poświęcić czas na weryfikację wniosku. To powoduje ustawianie się dużych kolejek przed konsulatami, bo musimy te procedury wizowe przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu weryfikować. Natomiast oczywiście z tego, co wiem, kierunek indyjski będzie, mam nadzieję, wzmacniany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jeśli chodzi o komponent konsularny. Pytanie pani poseł Piekarskiej, ale nie ma jej. Jeśli chodzi o wsparcie kadrowe urzędów wojewódzkich, to już się wydarzyło. To znaczy, że my możemy dać pieniądze na etaty, ale musimy zatrudnić też ludzi. Ci ludzie muszą być chętni do pracy w warunkach przedstawianych przez wojewodów przy obsłudze cudzoziemców, co nie jest pracą prostą. Ale to już się wydarzyło i kadry urzędów wojewódzkich są wzmocnione na tyle, żeby w naszej ocenie w sposób sprawny poradzić sobie z procedowaniem nad sprawami dotyczącymi legalizacji pobytu.

To znaczy, że nie mamy informacji i zresztą nie widać tego, żeby nasze polskie szkoły miały jakieś problemy absorpcyjne, jeśli chodzi o przyjmowanie dzieci obcokrajowców do szkół. To się po prostu dzieje. Natomiast, tak jak powiedziałem na wstępie, nie przewidujemy żadnej nagłej fali napływu osób chcących pracować na polskim rynku pracy. To jest raczej zmiana usprawniająca te procedury tu i teraz i dla tych osób, które już właściwie są na polskim rynku. Pan poseł Urbaniak z Konfederacji pytał o kwestię bezpieczeństwa i podniósł kwestię adresu we wniosku. We wniosku cudzoziemiec i tak podaje adres, bo przecież gdzieś tę decyzję musimy wysłać. Natomiast nie chcemy, żeby to był warunek konieczny, żeby on pokazywał, jaki ma tytuł prawny, jeśli chodzi o posiadanie tej nieruchomości. Proszę też wziąć pod uwagę fakt, że każdy cudzoziemiec starający się o jakąkolwiek formę legalizacji pobytu jest sprawdzany przez odpowiednie służby: ABW, Policję i Straż Graniczną. Takie sprawdzenie trwa 30 dni i w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone do 60 dni.

Pytanie pana posła Wojciechowskiego. Musielibyśmy wprowadzić system, który niemalże przypisuje pracownika do pracodawcy. To znaczy, że jeżeli pracownik przyjeżdża do pracodawcy, a znajdzie pracę lepszą, to jego prawem jest tego pracodawcę zmienić. Aczkolwiek słyszeliśmy rzeczywiście, że dochodziło do takich sytuacji, przede wszystkim w sektorze rolnictwa, że pracownicy przepływali od gospodarstwa rolnego do gospodarstwa rolnego, bo tam mieli więcej zapłacone.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druki nr 1677 i 1688) Bardzo proszę pana posła Roberta Telusa o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Państwo Ministrowie! Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, druk nr 1677. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 i art. 40 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 26 października 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania.

Holdingu, który jest oczekiwany przez rolników, holdingu, który ma pomóc w całym łańcuchu spożywczym, holdingu, który ma być akumulatorem, jeżeli chodzi o ceny.

Bo gdyby to były koncerny polskie, to myślę, że byłoby o wiele łatwiej, ale zazwyczaj są to koncerny zagraniczne i koncerny, które bardzo mocno wykorzystują rolnika i swoją pozycję, bo są silnymi koncernami w tym całym łańcuchu spożywczym, wykorzystują w ten sposób, że rolnikom płacą ceny bardzo niskie przede wszystkim za owoce miękkie, ale chodzi tu nie tylko o owoce miękkie, lecz także o wszystkie produkty rolne. Bywa tak, że rolnik przywozi swoje produkty do skupu i tak naprawdę nawet jak rozładuje swoje produkty, to nie wie, w jakiej cenie koncerny zapłacą. Dobrze by było, żeby to była państwowa firma, która będzie miała wpływ na ceny, będzie miała wpływ na skup. Holding jest tworzony w Ministerstwie Aktywów Państwowych i na bazie spółki Skarbu Państwa, spółki cukrowej. Żeby ten holding stworzyć, jest potrzeba, aby przekazać również inne spółki, które w tej chwili są we władaniu albo w zarządzaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który jest pod ministrem rolnictwa. Powstała pewna wątpliwość, wątpliwość prawna, czy na bazie tego prawa, które w tym momencie mamy, jest możliwe przekazanie aktywów tych spółek do Ministerstwa Aktywów Państwowych, do innego resortu, pod zarządzanie innego resortu. Żeby właśnie tę wątpliwość rozwiać, jest wniesiony ten projekt ustawy, poselski projekt ustawy, który ma tak naprawdę tylko dwa artykuły, który tak naprawdę prawnie rozwija te wątpliwości, że KOWR, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, będzie mógł te aktywa tych spółek, które są potrzebne, które są niezbędne do stworzenia tego holdingu, przekazać zgodnie z prawem.

Tutaj ubolewamy nad tym faktem, dlatego że z jednej strony posłowie opozycji mówią, że holding jest bardzo potrzebny, że ten holding powinien już być, dlaczego go jeszcze nie ma, a jak przychodzi co do czego, jak przechodzimy już do takiego konkretnego: sprawdzam, głosowania, to albo są posłowie przeciw, albo są wstrzymujący się. W tej sprawie to były głosy wstrzymujące się. Mimo że rozmawia się z posłami, którzy wiedzą o tym, że ten holding jest bardzo potrzebny i że ten holding pomoże polskiemu rolnikowi, to w głosowaniu widzimy, że jest inaczej. Dlatego, pani marszałek, Wysoka Izbo, proszę w imieniu komisji o to, aby - tak jak już przeczytałem na wstępie - ten projekt uchwalić.

Przez te zaniedbania, które były przez wiele lat, bo to, że polskie przetwórnie, które były kiedyś polskie, zostały sprzedane w ręce koncernów zagranicznych, to oczywiście jest wina. tych, którzy na to pozwolili w Polsce do tej pory, którzy odpowiadali za polskie rolnictwo w kilku rządach, bo to nie tylko jeden rząd, ale kilka rządów do tej pory.

Takim przykładem na to, że to jednak jest, skutkuje, była sprawa tzw. Eskimosa. Myślę, że posłowie z komisji rolnictwa wiedzą, o czym mówię. Wtedy właśnie minister Ardanowski podjął taką bardzo daleko idącą decyzję, decyzję, która była bardzo potrzebna. i zobaczcie, drodzy państwo, co się wtedy stało. firma zaczęła skupować na zlecenie pana ministra Ardanowskiego, wtedy ceny jabłek wzrosły do 30, a nawet w niektórych miejscach trzydziestu paru groszy.

Jeszcze raz chcę to podkreślić, bo tutaj pani poseł tak mocno krzyczy: Nieprawda, nieprawda.

I tak naprawdę dzisiaj decyduje o cenie produktów rolnych u rolnika nie rolnik, tylko decydują właśnie te koncerny, na które wy pozwoliliście.

Od 6 lat, ma pani poseł rację, 6 lat. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Bardzo proszę, pan poseł Kazimierz Gołojuch, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, druki sejmowe nr 1677 i 1688. Ustawa ta ma na celu umożliwienie przekazania na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych przez krajowy ośrodek temu ministrowi akcji lub udziałów, z których prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Trzeba dodać, że ten projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczno-gospodarcze, nie generuje skutków finansowych zarówno dla budżetu państwa, jak i dla samorządów terytorialnych. Klub Prawo i Sprawiedliwość wnosi od Wysokiego Sejmu o uchwalenie procedowanego projektu ustawy zawartego w druku nr 1688. Bardzo proszę, pani poseł Dorota Niedziela, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę słuchać, panie pośle. Te obietnice złożył publicznie Krzysztof Jurgiel. Po 2 latach jego następca Krzysztof Ardanowski tę obietnicę powtórzył. A więc 16 listopada 2018 r. powołano pełnomocnika ds. utworzenia narodowego holdingu spożywczego. Przez kilka miesięcy specjalnie zatrudniony pracownik otrzymywał wynagrodzenie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo 20 listopada 2018 r. został powołany Zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej, czytaj: holding. Za kilkadziesiąt tysięcy złotych wynajęto firmę, która miała znaleźć kolejną, która stworzyłaby biznes plan dla krajowej grupy spożywczej. Na te wszystkie działania Skarb Państwa wydał setki tysięcy złotych. Działania ministra Ardanowskiego w kwestii holdingu najlepiej podsumował europoseł Krzysztof Jurgiel, cytuję: Uprawianie polityki słów, a nie czynów, publicznego zapowiadania działań, które w większości nie były realizowane. Sztandarowym przykładem jest wielokrotna zapowiedź utworzenia holdingu spożywczego, później grupy spożywczej, które nigdy nie zostały zrealizowane. Nic dziwnego, że misję holdingu przeniesiono do Ministerstwa Aktywów Państwowych i zabawa, oczywiście za pieniądze podatników, zaczęła się od nowa. Od lutego 2020 r. działają kolejne zespoły, doradcy, prezesi, a jakże, za pieniądze podatników.

Odpowiedź jest bardzo prosta, Wysoka Izbo. Ta ustawa to kolejny skok Zjednoczonej Prawicy na państwową kasę. Pomysł jest następujący. Niech pan dobrze słucha, panie pośle.

Ta ustawa to prosta droga do wyprowadzenia majątku, który trafi pod zarząd tłustych kotów politycznych Porozumienia i Bóg wie kogo. Mało wam? Najpierw wymieniliście wszystkich członków zarządów tych spółek, kilkadziesiąt osób, a teraz sięgacie po majątek tych spółek? Wartość nominalna udziałów spółek, na których Zjednoczona Prawica chce położyć łapy, to prawie 700 mln zł.

Na tym majątku, na tych miliardach za chwilę położą ręce kolejni Misiewicze i działacze PiS-owscy. Twierdzicie, że majątek tych spółek ma zabezpieczyć działania rynkowe holdingu. Holding ma waszym zdaniem łamać zmowy cenowe. Wy już łamaliście zmowy cenowe w 2018 r. Wtedy interwencję na rynku jabłek prowadził minister Ardanowski. Wiecie, ile Skarb Państwa stracił na tej interwencji? Prezesem był senator PiS-u, wiceminister rolnictwa w waszym rządzie, który obecnie siedzi w areszcie. Wiecie, ile stracił Skarb Państwa na tej pomocy? Nie ma naszej zgody na takie uprawianie polityki.

Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę, pan poseł Marcin Kulasek, Lewica. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość ma wiele ikonicznych osiągnięć. Miliony samochodów elektrycznych, budowa promów przez stocznię w Szczecinie, elektrownia węglowa w Ostrołęce. Wszystkie te wielkie inwestycje łączy jedna cecha: nigdy nie zostały zrealizowane. Zapowiadaliście wielkie projekty, tworzyliście piękne slajdy i nie zrealizowaliście tych tematów. Do tego dochodzi jeszcze jeden projekt: narodowy holding spożywczy. Ile było zapowiedzi, ile zespołów roboczych, ilu konsultantów, ile to wszystko kosztowało pieniędzy nas wszystkich, podatników, ilu ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu brało w tym projekcie udział, brało się z tym projektem za bary. Efekt jest i był taki sam: zerowy. Teraz posłowie PiS przedstawili Wysokiej Izbie projekt ustawy, którego celem jest przeniesienie odpowiedzialności za utworzenie narodowego holdingu spożywczego na barki ministra aktywów. Czy to się uda? Jak mówi stare powiedzenie, na słowie Sasina polegaj jak na Zawiszy. Żadnemu z trzech PiS-owskich ministrów rolnictwa nie udało się utworzyć holdingu. To logiczny wniosek, że misje z kategorii: mission impossible powierzycie swojej strategicznej rezerwie kadrowej - premierowi Sasinowi. Za ideą utworzenia narodowego holdingu spożywczego wokół Krajowej Spółki Cukrowej stoją racjonalne przesłanki. Czy takie przesłanki stoją za powierzeniem tej misji premierowi Sasinowi? Mam tylko jedną prośbę: bądźcie oszczędni. Nie wyrzucajcie milionów na zachodnie firmy doradcze, nie twórzcie nowych synekur. Pamiętajcie, że gospodarujecie publicznym groszem i że 70 mln to bardzo dużo pieniędzy. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Klub Lewicy zagłosuje przeciwko poselskiemu przedłożeniu. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle.

Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, druki nr 1677 i 1688. Wydaje się, że opozycja nie powinna być przeciwna. Nie naszą rolą jest znajdowanie narzędzi, w oparciu o jakie powinien być zbudowany holding, bo to rząd bierze za to odpowiedzialność, tylko obserwując to już przez te 6 lat, kiedy były pierwsze zapewnienia o tym, że holding powstanie, że on będzie wspierał rolników, że będzie zbierał nadwyżkę z rynku, że będzie kształtował ceny. Tylko, panie ministrze, pytanie już na początek: Ile procent rynku musielibyście skupić w swoich rękach, żeby taką cenę móc kształtować? Co zrobiliście po drodze? To przejęcie chociażby Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek za długi wobec Skarbu Państwa. To już powinien być zakład, spółka holdingu spożywczego.

Tak wspieracie. Po drodze padł Ozorków, padł Rypin. Dalej wiele prywatnych firm, które dawały miejsca pracy, skupowały produkty z rynku. Ich nie ma. Ziarno to przecież też przyjaciele przedstawicieli rządu i posłów właśnie Zjednoczonej Prawicy, które oszukało wielu rolników. Nikt ich do odpowiedzialności karnej nie wezwał. Niestety to się nie zadziało. Tak jak powiedziałem z tej mównicy, że CPK to centralna pralnia Kaczyńskiego, bo nic nie powstało, ale pełnomocnicy, firmy, wasze firmy zarabiają na tym ogromne pieniądze, tak znowu to będzie państwowa dojarnia - dojarnia spółek, dojarnia rolników. Bo o co chodzi z przejmowaniem tych udziałów, akcji? Piękne gospodarstwo w województwie zachodniopomorskim, Nowielice. Zostało to wszystko przez waszego dyrektora sprzedane. Dzisiaj jest prowadzona uprawa roślinna, jakieś łąki, które tak naprawdę powinny być jako baza paszowa dla bydła, ale dzisiaj dopłaty wpływają na konto, a za chwilę, żeby nie było widać, jak wasz kolejny fachowiec położył kolejną spółkę, przekaże się ją do Ministerstwa Aktywów Państwowych, do Sasina. I tak się żongluje tymi pieniędzmi, żeby ukryć faktyczny stan zadłużenia, stan finansów, i tak przerzuca się. Teraz może trzeba będzie którąś spółkę szybko przekazać. Gospodarstwo, które było wzorcowe, ośrodek doradztwa rolniczego, miejsce słynne z wielu wystaw, z wielu dużych wydarzeń dla wszystkich, którzy się interesują rolnictwem, pracują w tej branży, w tej otoczce rolnictwa. Za chwilę może też trzeba będzie przekazać, powiedzieć: budujemy holding, jest to niezbędne, konieczne, szybko przekażcie, a my sobie poradzimy. Chcieliście budować holding? Dziś powinno być przynajmniej tyle, ile starych województw, sklepów skupionych w rękach właśnie tego już sławetnego, obiecanego holdingu.

To powinno się dziać. Jeśli przychodzi do działania, to przekręt przekrętem przekręt pogania. Ale będziemy patrzeć wam na ręce i oczywiście za chwilę pewnie będziemy przedstawiać tutaj informację, że mieliśmy rację. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Paulina Hennig-Kloska, Polska 2050. Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Ale ponieważ tak naprawdę ma on kupić jeszcze trochę głosów poparcia na wsi, to powołujecie go teraz, kiedy spada wam poparcie, a wy szykujecie się do kolejnych wyborów. Hortex był sprywatyzowany za czasów AWS-u, jak pamiętam, a to było ugrupowanie współtworzone przez wielu polityków PiS.

Tak ją napisaliście, że mamy dużą kolizję prawną i minister aktywów państwowych nie może mieć nawet z KOWR-u przekazanej ziemi będącej w zasobach własności rolnej Skarbu Państwa, bo okazuje się, że w praktyce dokonanie tej czynności jest kwestionowane, jest niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Sytuacja przeciętnego polskiego rolnika jest coraz trudniejsza. Od 6 lat mamicie rolnika, że coś się zmieni. Krzyczycie, że jesteście głównym reprezentantem wsi w parlamencie, a sytuacja rolnika się pogarsza. Taka jest sytuacja.

Pan poseł Michał Urbaniak, Konfederacja. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam dylemat, ponieważ to jest ustawa, która z jednej strony, można by powiedzieć, jest ustawą techniczną, ale z racji swojej prostoty też jasno wskazuje pewien kierunek polityczny. Szanowni Państwo! Daliście premierowi Sasinowi wybory kopertowe. Wiemy, jak to się skończyło. Daliście premierowi Sasinowi spór z Czechami o Turów. Wiemy, jak to się skończyło. Daliście państwo premierowi Sasinowi także Ostrołękę i wiemy, jak to się skończyło. Myślę, że dzisiaj, jak już premier Sasin dostał sasinadę, czyli igrzyska europejskie, nie podejmujmy już tej decyzji politycznej. Róbcie państwo, co chcecie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce zgłosić się jeszcze do zadania pytania? Jako pierwszy pan poseł Jan Szopiński, Lewica. 1 minuta na zadanie pytania. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgodnie z treścią uzasadnienia właścicielem gruntów opisanym w projekcie pozostaje Skarb Państwa, a zmienia się jedynie podmiot, który go reprezentuje. Wbrew pozorom jest to jednak bardzo istotna zmiana, gdy zmienia się przeznaczenie gruntów z rolnych na bliżej nieokreślone, ważne z punktu widzenia strategicznego grunty przemysłowe, wojskowe lub inne. Czy wystąpienie ministra o zmianę kwalifikacji gruntów nie powinno być poprzedzone ustawowo zapisanym obowiązkiem wcześniejszego uzyskania akceptacji służb geologicznych, ochrony środowiska oraz wszystkich innych, których zgody i opinie mogą być istotne z punktu widzenia przyszłego przeznaczenia gruntów? Wszyscy wiemy, że niektóre inwestycje planowane są na wyrost, w związku z czym mogą mieć znaczący wpływ na polską gospodarkę żywieniową, którą powinno się mimo wszystko pozostawiać na czele problemów strategicznych naszego kraju. Uprzejmie poproszę pana ministra o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. Wysoka Izbo!

Ust. 8 brzmi: „W przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji polityki gospodarczej państwa, w tym ochrony interesów Skarbu Państwa, na wniosek ministra właściwego do spraw aktywów państwowych Krajowy Ośrodek, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych akcje lub udziały, o których mowa w ust. 5” Panie Ministrze! Czy, a jeżeli tak, to kiedy, minister do spraw aktywów państwowych zamierza zbywać otrzymany majątek? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pytam o to, dlatego że ten proces trwa już wiele lat, środki finansowe z budżetu wypływają, nie widać efektów. W związku z tym istnieje podejrzenie, że o to właśnie chodzi, żeby to trwało, żeby przypominać o tym w trudnych momentach, kiedy sondaże nie stoją najlepiej, i powodować krótkotrwałe wzmożenie, które pomaga przełamać tę niemoc sondażową. Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że w tym bardzo długim procesie, który być może nigdy się nie skończy, dojdzie do wielu różnych nieprawidłowości, pytam: Czy ten proces zostanie objęty tarczą antykorupcyjną, nadzorem odpowiednich służb, tak żeby przy tej okazji nie wypływały poza budżet te środki finansowe? Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Mam pytanie do pana posła przedstawiciela wnioskodawców, a dotyczy ono uzasadnienia tego projektu. Otóż w treści uzasadnienia dokumentu, nad którym procedujemy, regulującego moim zdaniem kwestie kompetencyjne i mającego na celu usunięcie rozbieżności w dwóch ustawach - ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - wskazujecie państwo, że projekt tej ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczne i gospodarcze. Proszę zatem o wskazanie tych korzyści oraz ewentualne uszczegółowienie zasad, na jakich korzyści te zostały wyliczone. Bardzo dziękuję. Pani poseł Henryka Krzywonos-Strycharska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jakie środki z Krajowego Planu Odbudowy trafią do holdingu? Ilu nowych Misiewiczów i ile tłustych kotów wchłonie holding spożywczy? I czy już sporządziliście państwo listy działaczy PiS i członków ich rodzin, którzy znajdą zatrudnienie w narodowym holdingu spożywczym? Dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł Dorota Niedziela, Koalicja Obywatelska. Jakie są gwarancje, że Skarb Państwa nie straci kontroli nad spółkami strategicznymi, w tym ziemią państwową, jaką dysponują?

Cała pana interwencja, czyli 250 tys. t, nie miała żadnego wpływu na rynek.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałem spytać: Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zamierza uwłaszczyć spółki Skarbu Państwa nadzorowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? Przypomnę, że te spółki dzierżawią od Skarbu Państwa ok. 100 tys. ha gruntów rolnych.

Czy te kredyty mogą być kierowane na działalność operacyjną holdingu, czy na inne cele? Bo z praktyki wiemy, że pieniądze bardzo szybko się rozchodzą. A my coraz bardziej zastanawiamy się, kiedy ten proces (Dzwonek) się oddala, gdzie jest interes polskiego rolnika. Pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tak budujecie, że nie dalej jak rok temu procedowaliśmy tutaj nad ustawą antyrolniczą, piątką Kaczyńskiego, za co rolnicy was nazwali po imieniu: zdrajcy polskiej wsi. Dzisiaj mówicie, że to odbudujecie.

Dziękuję, panie pośle. To było ostatnie pytanie. Bardzo proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Szymona Giżyńskiego o odpowiedź na pytania.

Wysoki Sejmie! Jeżeliby porównać dzisiejsze obrady, rozpoczętą przez państwa dyskusję.

Takich głosów było kilka.

Ale przeważały głosy, które w ogóle abstrahowały od materii ustawy. Ustawa była gdzieś kompletnie na boku, za tą salą, ponad i poza rzeczywistością, ponieważ chodziło o coś zupełne innego. Państwo doskonale wiedzą, po co ten holding pojawi się na rynku któregoś, mam nadzieję, że już bliskiego dnia. Pojawi się jako interwent, i to zwycięski interwent, na rzecz polskiego rolnictwa i polskich rolników. Z kim się zmierzy? Zmierzy się z obcym kapitałem, z właścicielami wielkich przetwórni, takimi, którzy od lat 90. przechwycili sprzedawane za bezcen poszczególne składniki polskiego państwowego majątku i rządzą nim do dzisiaj. Wbrew temu, co powiedział jeden z przedmówców, pan Stefan Krajewski, nie jest tak, że trzeba zbudować jakąś gigantyczną machinę np. równoważną kapitałowo, żeby zwycięsko toczyć bój z obcą przewagą kapitałową. Jak w 2018 r. małymi sposobami udało się zachwiać, o czym mówił bardzo sensownie i bardzo konkretnie na tym przykładzie pan przewodniczący Robert Telus. Stosunkowo małe zaangażowanie kapitałowe wystarczyło, żeby do bardzo rzeczywistych, sensownych, opłacalnych dla polskich sadowników, dla polskich przetwórców. Wtedy oczywiście chodziło o jabłka.

Zarabiali utylizatorzy, zarabiali wielcy przemysłowcy, którzy weszli cudownie i płynnie w przemysł bioasekuracyjny, zarabiały sieci, bo w te wszystkie patologie się kapitalnie wmontowały, zarabiał oczywiście tucz nakładczy, bo też się w patologie i nierównowagi niekorzystne dla polskich rolników znakomicie wmontował. Więc to jest kwestia interesów. Specjalnie pewnym kontekstem wtrąciłem się, po to żeby też podać następny przykład, że właśnie wystarczyło krótkie anonsowanie przez parę dni, ale wiarygodne, rzetelne, że będziemy się wtrącać jako państwo w przemysł utylizacyjny.

Proszę państwa, niemieccy analitycy, bo tutaj przemysł niemiecki miał wtedy bardzo dużą przewagę - czy też: obcy, a nie polski - wieścili najpierw, że ASF ma w Polsce takie perspektywy i tak się będzie świetnie spisywał pod ich zarządem - tych wielkich firm i wielkich finansistów - że należy na najbliższe lata przewidzieć, że to będzie ok. 30 mld zł obrotu. Trzeba w tę branżę inwestować. Lekkie anonse ze strony państwa polskiego, ministerstwa rolnictwa, że my w to wejdziemy, spowodowały, że w takiej wielkiej masie kapitał inwestujący, jeszcze bardziej podtrzymujący branżę utylizacyjną się nie pojawił. Więc liczą się skutki, ale skutki, których źródłem jest wola i konsekwencja, a nie jakieś mityczne pieniądze. Proszę państwa, to, co się stało w tej chwili na tej sali, oczywiście nie dotyczy ustawy, bo ona jest prościutka, oczywista, ma charakter formalny, intencje są oczywiste; całkowita zgodność z prawem, tak żeby uniemożliwić jakiekolwiek kwestionowanie, żeby nie było żadnej luki na jakiś woluntaryzm czy inną podejrzliwość. Część przyznała to oficjalnie, a ta druga część, potężniejsza poszła już zupełnie w zaparte.

Dlaczego? Dlatego że holding pojawi się na rynku jako interwent w obronie polskich interesów, w obronie interesów polskich rolników, polskich przetwórców. To was najbardziej państwo drodzy boli. Dlaczego? Dlatego że to wy w swoich dobrych czasach byliście instalatorami tego przemysłu i później ASF-owego, właśnie takiego, który do tej pory dominuje w polskim przetwórstwie i tym samym w polskim rolnictwie.

Jesteście w dalszym ciągu, bo wasze umocowanie się nie zmieniło, po tamtej stronie, przeciwnej do polskich interesów.

Są prokuratorzy, jest prokuratura, są sądy, czekają na to, żeby te insynuacje znalazły się tam, gdzie ich miejsce. Ale niech ta konfrontacja będzie miała charakter formalny, bo go nie ma.

Jeszcze raz powtarzam: holding jest na polskim rynku i będzie projektowany jako silny interwent. I taka jest filozofia tego pomysłu i taka będzie jego skuteczność.

Proszę państwa, były również takie pytania, które doczekają się, i to szybko, odpowiedzi na piśmie, tym bardziej że z absolutnie formalnych powodów zdecydowanie istotna część, być może nawet przeważająca, tych pytań była kierowana do Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Większościowy udział Skarbu Państwa jest na dzisiaj w tym wyjściowym procesie zapewniony i będzie poprzez ten mechanizm, który pokazałem, tylko wzmacniany.

Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Roberta Telusa. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Co się stało?

Pani marszałek, jako sprawozdawca komisji już zabierałem głos, a teraz odpowiadam na pytania, które zostały zadane. Tak, jako sprawozdawca komisji odpowiadam na pytania, które zadali posłowie na sali.

Zjednoczona Prawica, rząd polski chce położyć łapę, a nie tak jak do tej pory wy wysprzedawaliście wszystko. Chcę przypomnieć, że wy sprzedaliście wszystko: i przetwórnie, i horteksy, i firmy, które zajmowały się skupem.

Nie, no nie ma to nic wspólnego, pani poseł, że sprzedawaliście wszystko, co się rusza. A my chcemy. Panie pośle, bardzo przepraszam.

Pani marszałek, jako sprawozdawca komisji odpowiadam na pytania, które zadali posłowie. No tak, zgadzam się z tym, waszej zgody na to, żeby to było polskie i żeby było w polskich rękach, żeby było państwowe, nie ma. My to wiemy i myślę, że Polacy też to wiedzą. W jakiś sposób bardzo zaskoczył mnie też głos posła PSL, który to samo mówił: że to będzie państwowa dojarnia.

Panie pośle, wiem, że ma pan poglądy narodowe. To jest człowiek, który dba o interes narodowy. Dba o interes narodowy. Przecież pan wie o tym, panie pośle, że panu premierowi Sasinowi zależy na tym, żeby to było polskie.

Pani poseł Iwony Marii. Przepraszam, że zapomniałem.

Potrzebna jest interwencja na rynku skupu, dlatego że w tej chwili całe przetwórstwo, handel w Polsce mają koncerny zagraniczne.

Mam świadomość, że nie wszyscy to rozumieją, bo nie wszyscy zajmują się polskim rolnictwem. Dlatego bardzo dziękuję pani poseł za to naprawdę merytoryczne i sensowne pytanie.

Jeszcze raz: 1200 mln euro z Polskiego Ładu na polskie przetwórstwo. Nigdy tak nie było. Tak nie było, bo wy robiliście wszystko, żeby sprzedać polskie przetwórstwo, i to wam się udało. Słyszałem, że rządziła w Polsce. Polacy pamiętają o tym i będą pamiętać, bo wy doprowadziliście do tego, że sprzedano wiele polskiego majątku.

I naprawdę nie przeszkadzajcie, nie krytykujcie, nie głosujcie przeciw. bo ten holding jest potrzebny.

A jeżeli zależy wam na tym. Pani Marszałek! Drodzy Państwo!

Ale my wam udowodnimy, że nawet jak będziecie przeciw, nawet jak będziecie tak mocno krzyczeć, zrobimy to, bo to jest dla polskiego rolnictwa, a my jesteśmy gotowi zrobić wszystko. Dlatego jeszcze raz dziękuję, panie ministrze, za tę ustawę, że przygotowaliśmy ją wspólnie, mimo że to jest ustawa poselska, ale w uzgodnieniu z ministerstwem. Wiem o tym, że ona jest bardzo potrzebna.

Dlatego, drodzy państwo, jeszcze raz jako sprawozdawca w imieniu posłów komisji rolnictwa, bo tam naprawdę była ta dyskusja merytoryczna, proszę państwa o to, żebyśmy poparli tę ustawę, bo ona jest naprawdę potrzebna dla polskiego rolnictwa. Dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projekt ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (druki nr 1676 i 1744) Bardzo proszę pana posła Tomasza Ławniczaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, zawartym w druku nr 1676. Powyższy projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 22 października 2021 r., zaś marszałek Sejmu skierowała go 26 października br. do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do pierwszego czytania. W dniu 15 listopada ww. komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły projekt.

Powyższy wyrok dotyczył zbadania konstytucyjności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wywołał skutek retroakcji, czyli cechy norm prawnych mających moc wsteczną, zwłaszcza w zakresie nowelizacji definicji budowli oraz definicji elektrowni wiatrowej. W wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność art. 17 pkt 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie, w jakim narusza zasadę nieretroakcji, i zobowiązał ustawodawcę do podjęcia prac legislacyjnych mających na celu opracowanie regulacji rekompensującej gminom straty poniesione w wyniku wprowadzenia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii. W wyniku analizy ww. wyroku Rada Ministrów podjęła decyzję o przygotowaniu projektu ustawy dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego pierwszego szczebla, bowiem obecnie nie istnieją przepisy, na podstawie których byłaby możliwa realizacja wypłat gminom rekompensat wskazanych przez trybunał. W związku z powyższym realizację wyroku trybunału można wdrożyć w życie wyłącznie poprzez uchwalenie stosownego projektu uchwały. W trakcie dyskusji było kilka pytań, ale nikt nie wniósł poprawek do przedłożonego projektu. Dziękuję. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Jako pierwszy głos zabierze pan poseł Tomasz Ławniczak, Prawo i Sprawiedliwość. Chciałem tylko dodać do tego, bo nie będę już tutaj powielał tego, o czym mówiłem, że mianowicie nie jest to, jak niektórzy myślą, ustawa wiatrakowa, która wprowadzała zasadę 10H, tylko jest to zmiana tej ustawy z czerwca 2018 r., która wprowadzała zmiany w ustawie o budownictwie - tutaj chodzi o definicję budowli - oraz w ustawie właśnie o elektrowniach wiatrowych w zakresie definicji elektrowni wiatrowych. To powodowało zmiany podatkowe.

Jest to po prostu realizacja tego wyroku.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Poncyljusz, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Tą ustawą zajmujemy się dlatego, że klub Prawo i Sprawiedliwość w maju 2016 r. w tej Izbie przegłosował ustawę, która tak naprawdę zabiła energetykę wiatrową na lądzie. Zabito rozwój energetyki wiatrowej.

Tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy o ustawie, która nie budzi kontrowersji, bo wiadomo, że gminom trzeba zrekompensować straty, ale rekompensowane są straty tylko za rok 2018, w którym Prawo i Sprawiedliwość przeforsowało kolejną ustawę, tzw. nowelę OZE.

Ostatnia rzecz. Namawiam pana ministra, żeby tak samo szybko procedować nad ustawą odblokowującą budowę wiatraków w Polsce.

Pół miliarda złotych to kolejny koszt głupiej, nieprzemyślanej, pozbawionej rozsądku polityki energetycznej polskiego państwa, polityki państwa, na której tracą wszyscy. Tracą samorządy, tracą przedsiębiorcy, tracą lokalne społeczności i traci też nasz budżet. Tak naprawdę to my, podatnicy, zapłacimy za błędy rządu. Nie rząd, nie ministrowie, nie ci, którzy uchwalali szkodliwe, niezgodne z konstytucją prawo. Tym kosztem zostają obciążone kieszenie Polek i Polaków, a te 0,5 mld zł to i tak jest za mało, dlatego że nie jest w nich uwzględniona ani inflacja, ani koszty kredytów, które gminy musiały wziąć.

Ale premier Morawiecki mówi dzisiaj, że pieniędzy mamy w bród. Co więc za problem, żeby wyrzucać je w błoto?

Nic dziwnego, że galopują ceny energii. Nic dziwnego, że walka z ubóstwem energetycznym stała się totalną klapą w Polsce. Za butę i głupotę rządu płacą dzisiaj ludzie wysokimi rachunkami i samorządowcy dodatkowymi kosztami i problemami. Polityka energetyczna to obszar rekordowych strat, rekordowej niekompetencji, codzienny chleb polskiego rządu. Niezwykle drogo kosztuje nas głupota PiS-u. Niezwykle droga jest walka polskiego rządu z wiatrakami. Symbolem głupiej, wyniszczającej polityki pozostanie wypowiedź minister Zalewskiej, posłanki symbolu walczącej z wiatrakami, która doprowadziła w zasadzie do zamrożenia branży wiatrakowej.

Skutki polityki opartej na strachu przed śmigłem wielkości autobusu spadającym na głowę odczuwamy codziennie i będziemy odczuwać przez długie lata. Jako Lewica popieramy ten projekt, dlatego że uznajemy zasadność wypłacenia rekompensat za prawo, które było niezgodne z konstytucją, ale nie popieramy wyrzucania pieniędzy w błoto, głupiej, bezmyślnej polityki opartej na uprzedzeniach, braku skoordynowanych działań, obarczaniu kieszeni podatników nieodpowiedzialnością rządzących. Dziękuję bardzo, pani poseł.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Koalicji Polskiej - PSL, Unii Europejskich Demokratów, Konserwatystów, Marka Biernackiego przedstawić stanowisko klubu w sprawie projektu ustawy z druku nr 1676 o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Ustawa, nad którą dzisiaj procedujemy, jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., a dokładnie z 22 lipca, do którego wniesione zostały protesty, wnioski rady gminy Świecie nad Osą oraz rady gminy Kobylnica o zbadanie zgodności z konstytucją regulacji przewidującej wejście w życie z mocą wsteczną przepisów nadających nowe brzmienie definicjom budowli i elektrowni wiatrowej. Ale wracam do historii. Ustawa odległościowa, bo tak ją nazywano, z 2016 r. podniosła opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości stanowiącym wyłączny dochód gmin. Wcześniej podatek ten był płacony jedynie od części budowlanej i stanowił 30% wartości turbiny. Od 2017 r. podatkiem od nieruchomości obłożono również część techniczną. Rozwiązanie to zostało w 2018 r. zniesione wstecznie - od początku 2018 r. - jako niezgodne ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski. Tymczasem gminy uwzględniły już zwiększone wpływy w swoich budżetach i w związku z tym zaplanowały odpowiednio wyższe wydatki. W związku z tym zostały pozbawione spodziewanych wpływów, dlatego że musiały zwrócić nienależnie pobrany podatek za 2018 r. To z kolei spowodowało, że nie mogły zrealizować wielu założonych wcześniej inwestycji i nie mogły skorzystać np. z różnych projektów realizowanych z Unii Europejskiej. W wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niekonstytucyjność art. 17 pkt 2 noweli ustawy o OZE, ustawodawca musi dzisiaj dokonać rekompensaty na rzecz samorządów. Ta rekompensata dotyczy ok. 200 gmin, na obszarze których zlokalizowane są elektrownie wiatrowe. Środki te po złożeniu stosownych wniosków do wojewody w ramach rezerwy celowej budżetu państwa w 2022 r. zostaną wypłacone samorządom. Wysoka Izbo! Po zapoznaniu się z tym projektem ustawy, wiedząc, że w dzisiejszych czasach każdy grosz i każda złotówka dla samorządu są ważne, będziemy popierać ten projekt ustawy. Bardzo dziękuję.

Panie Ministrze! Ta ustawa jest najlepszym przykładem tego, jak rząd PiS potrafi marnować pieniądze obywateli, przepalając je w zasadzie, bo inaczej tego nazwać nie można. To mechanizm złego stanowienia prawa od początku do końca, z nieposzanowaniem praktyk zwykłych, gospodarczych czy w zakresie legislacji, za który dzisiaj z budżetu państwa trzeba zapłacić 0,5 mld zł, a w gruncie rzeczy jeśli z budżetu państwa, to tak naprawdę z kieszeni obywateli, bo przecież nasz budżet w ponad 90% to podatki, na które składają się właśnie obywatele. O czym on mówi? O tym, że oddamy samorządom utracone dochody wynikające z podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 r. Było to już tutaj tłumaczone. Najpierw rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł opodatkowanie turbin wiatrowych, zwiększając zakres tego opodatkowania. Potem międzynarodowe koncerny wniosły do sądów arbitrażowych wnioski, bo nie godziły się na wsteczne działanie takiego prawa. Było to potraktowane jako zmiana zasad w trakcie gry. W związku z tym, że rząd nie chciał płacić ogromnych odszkodowań z budżetu państwa, prawo wstecznie zmienił. Samorządy, mimo że miały to zaplanowane w budżetach, pieniędzy nie dostały, a tak jak tu mówiła pani poseł, mogły już je wydać, mogły to zaplanować, bo podstawa prawna ku temu była. Dzisiaj mamy to oddać. Mam nadzieję, że środki te będą dobrze spożytkowane, na ważne inwestycje czy też realizację zadań własnych przez te samorządy. Dwa pytania. Od 2018 r. te pieniądze straciły na wartości. TK w wyroku o tym nie mówił, ale też nie wiedział, kiedy i w jakich warunkach gospodarczych, tudzież inflacyjnych, ten wyrok zrealizujecie.

Oczywiście sam projekt poprzemy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Korwin-Mikke, Konfederacja.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z przyjemnością zauważam, że gminy dbają o swój interes i pozwały państwo polskie o odszkodowanie. Konfederacja stawia jednak pytanie: Kiedy państwo polskie zadba o swój interes i pozwie Unię Europejską o straty, jakie ponieśliśmy, montując te elektrownie wiatrowe? Koszt prądu z elektrowni wiatrowych jest znacznie wyższy, nawet po doliczeniu, że od węgla pobieramy dodatkowe podatki. Co więcej, prąd z elektrowni wiatrowych to jest, krótko mówiąc, śmieć energetyczny.

Jest to zakłócenie systemu, a nie pomoc. Powinniśmy od Unii Europejskiej wyciągnąć o wiele, wiele większe pieniądze niż gminy od państwa polskiego.

I, proszę państwa ten, kto najtaniej i najlepiej produkuje, ten wygrywa. Państwo się do tego w ogóle nie miesza. Wtedy gminy nie miałyby od kogo brać pieniędzy, od kogo żądać, bo po prostu sobie kapitalista założył, albo zamknął - to jest ich problem. Natomiast tutaj to roszczenie gmin powstaje stąd, że to państwo się wzięło za politykę energetyczną, a nie zostawiło jej po prostu rynkowi. Bo działanie rynku, proszę państwa, oznacza spełnianie życzeń ludzi: nie przemysłowców, nie biurokratów, tylko konsumentów.

Bo celem produkcji jest konsumpcja. O tym się zapomina, bo my realizujemy postulaty ludzi pracy, kapitalistów, a zapominamy o podstawowym elemencie gospodarki - o odbiorcy. Tak że proszę jeszcze na zakończenie, żeby rząd łaskawie zechciał rozważyć wystąpienie do Unii Europejskiej o gigantyczne odszkodowanie za te pomysły z wiatrakami i innymi odnawialnymi źródłami energii. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Bardzo proszę.

Pani Marszałek! Realizując tę tradycję, chciałbym zapytać o kwestię dotyczącą tej ustawy. Mianowicie, moim zdaniem ta ustawa to brak spójności tworzonego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości prawa.

Jednak pomimo licznych wniosków płynących ze strony samorządów pominięto wtedy kwestię utraconych z tego tytułu przychodów. Pominę kwestię, w jaki sposób samorządy mają realizować powierzone im zadanie, jeśli rząd z takim opóźnieniem reaguje na ich problemy. Chciałbym natomiast zapytać z tego miejsca, czy kwestie te zostały odpowiednio uregulowane w bliźniaczych projektach dotyczących zwolnień podatkowych w odniesieniu do budowli związanych z infrastrukturą lotniczą czy kolejową.

Bardzo proszę, pan poseł Rafał Adamczyk, Lewica. To pani poseł Henryka Krzywonos-Strycharska, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Niektóre samorządy, aby pokryć stratę dochodu w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, musiały zaciągnąć zobowiązania. Zobowiązania wiążą się z odsetkami. Podczas konsultacji publicznych związek gmin wielkopolskich zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości poszerzenia rekompensaty o koszt odsetek. Odpisaliście państwo, że nie można tego pokryć i zrealizować, i tu cytuję: z powodu złożonej sytuacji budżetu państwa. A teraz mam pytanie: Dlaczego nie chcecie państwo poszerzyć rekompensaty o koszt odsetek? Przecież pan premier wszędzie wygłasza, że nasz budżet ma nadwyżki.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zapominamy, skąd się wziął problem farm wiatrowych w Polsce. Wziął się stąd, że dużo szmelcu z Europy Zachodniej w czasie boomu wiatrakowego przyjechało do Polski. Tak, widziałem ten szmelc. Wielokrotnie.

W tej chwili gminy już się nauczyły stawiać wiatraki, tak jak i przedsiębiorcy się nauczyli, że na wiatrakach można rzeczywiście zarobić.

Nie ma pana posła. Pan poseł Tomasz Olichwer, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiaj chcemy zrekompensować jedynie straty gmin za połowę 2018 r., ale przy tej okazji, przy tej ustawie chciałbym przypomnieć, że gminy nadal czekają na projekt ustawy w sprawie zmiany ustawy o elektrowniach wiatrowych, który tak szumnie był zapowiadany jeszcze przez panią minister Emilewicz, a wciąż nie został przez Radę Ministrów przedstawiony Sejmowi. A dotyczył rozwoju budownictwa mieszkaniowego, czyli rozwoju tych miejscowości. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Ponad 500 mln zł zostanie zwrócone gminom.

Na pewno rząd nie ma takich informacji, będą to grube miliardy. Przy okazji powiem - bo jest tutaj przewodniczący komisji samorządu terytorialnego - że jest taka gmina Dobrzyń Wielki, która została podzielona, odebrano jej tereny miasta Opole i ta gmina nie może się rozwijać.

Dziękuję bardzo. Nie ma pana posła. Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zabiliście w 2016 r. całkowicie elektrownie wiatrowe, mimo że to jest najtańsza energia odnawialna.

Podnosiłam wówczas argument, że tak wysokie opodatkowanie spowoduje ich całkowitą likwidację. W 2018 r. przyznaliście mi rację i wycofaliście się z opodatkowania całej elektrowni wiatrowej, czyli podstawy, wieża i łopaty, tylko oczywiście zrobiliście to źle. Przyjęliście ustawę, która działa wstecz, co jest sprzeczne z konstytucją. Teraz przez bezmyślność rządu Polacy będą musieli wydać ponad 524 mln zł na rekompensaty dla gmin (Dzwonek) za nieumiejętne wprowadzenie prawa przez ten rząd. Kiedy wreszcie przedstawicie projekt ustawy przywracającej możliwość budowy nowych elektrowni wiatrowych w Polsce? Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wszyscy widzimy i oceniamy: chaos, bałagan, niekompetencja, procedowanie i dociskanie ustaw w nocy.

To efekt działalności Prawa i Sprawiedliwości.

Stało się. Samorządom zlikwidowaliście dochody z podatków, mało tego, samorządy na co dzień tracą pieniądze, bo na ich terenie nie wybudowano kolejnych wiatraków. Panie Ministrze!

Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 524 mln zł to pieniądze, które tym samorządom się należą. Szkoda tylko, że tak długo musieliście myśleć nad tym, żeby to przywrócić. Nie interesowaliście się tym. Szanowni Państwo! Zlikwidowaliście 5 tys. miejsc pracy.

Naprawdę tym ludziom, tym gminom należy się powrót do normalności, dlatego będziemy za tym, żeby głosować za tą ustawą, ale również za tym, żeby jak najszybciej to odblokować. Proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Ta ustawa pokazuje w pigułce, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość traktuje samorządy, czyli wszystkich mieszkańców mniejszych i większych gmin w całej Polsce, przyjmując wiele ustaw, które w sposób oczywisty ograniczają dochody samorządów.

Takie uderzenia były w wielu ustawach, niestety niezbyt wiele później trafia do parlamentu ponownie, żeby tę sytuację pokazać i naświetlić. Takich ustaw było wiele i tak być nie powinno.

Bardzo proszę, pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Podobne pytanie.

Nie pierwsze, nie ostatnie, kolejne, jedno z nich. Zatem, po pierwsze, inflacja. Zatem to tylko częściowa rekompensata. Pierwsze pytanie: Jak zamierzacie wyrównać tę stratę? Bo ona jest i jeśli pokryje ją samorząd, to pokryjemy ją my, pokryję ja, pokryją pan poseł i pani poseł, po prostu my, mieszkańcy. Więc jak będzie wyglądała pełna rekompensata? I pytanie drugie dotyczące pewnej filozofii rozwoju (Dzwonek) farm i pozyskiwania w ten sposób energii.

Pani Marszałek!

Widzę w ostatnim czasie, że nie ma tego poszanowania dla władzy samorządowej, bo tam często nie są nasi, bo często ktoś inny rządzi, a przecież system się sprawdza. Konstytucyjnie jeżeli ustawa wprowadza zmiany finansowe i traci na tym samorząd, powinna być kompensata z automatu. Nie poprzez trybunał, nie przez jakąś instytucję państwową, tylko z automatu. Czy nie możemy wypracować takiego systemu, że gdy wchodzi ustawa, która zabiera jakąś część przychodów czy dochodów samorządu, to od razu jest w niej ujęte, że państwo kompensuje tę stratę? Są komisje rządowa i samorządowa, można tam to regulować.

Dziękuję.

Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! Skutkiem wprowadzenia rozwiązań ideologicznych do ustawy, która reguluje prawne funkcjonowanie energii wiatrowej, jest to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Będzie częściowa rekompensata gminom za utracone dochody z podatku od nieruchomości. Ale m.in. w powiecie średzkim w Wielkopolsce, gdy mam dyżury poselskie w Dominowie, w Środzie Wielkopolskiej, samorządowcy pytają, kiedy wreszcie rząd przedstawi nowelę tych rozwiązań, bo to, co funkcjonuje, zaburza ład przestrzenny. To wszystko powoduje bardzo trudną (Dzwonek) sytuację, również dochodową, samorządów. Wobec powyższego chciałbym zapytać, kiedy rząd przedstawi nowelę tej ustawy i co jest powodem czy jakie są przyczyny tego, że ta ustawa tak długo jest w rządzie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Polski węgiel, polskie ciepłownictwo i polska elektroenergetyka są w sposób sztuczny opodatkowane przez Unię Europejską, bo najtańsza energia elektryczna produkowana jest w Bełchatowie. I my, szanowni państwo, popełniamy samobójstwo, podcinamy sobie skrzydła. Tego chcecie? Niestety PSL cały czas mówi głosem (Dzwonek) Waldemara Pawlaka, broniąc rosyjskiego gazu, a Lewica zapomniała o OPZZ, zapomniała o ludziach pracy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, pani poseł Monika Falej, Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rozwiązania proponowane w ustawie o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych to goła rekompensata. Nie uwzględnia się tu kosztów, jakie gminy musiały ponieść, nie uwzględnia się również rosnącej inflacji czy kosztów kredytów, kosztów związanych ze zmianą opodatkowania.

Bo to, co proponujecie, jest po prostu niesprawiedliwe. Przez to, że gminy tych pieniędzy nie mają, mieszkańcy nie mają usług, które powinni otrzymać w ramach pieniędzy, które akurat samorządy miałyby do dyspozycji. Bardzo proszę, pan poseł Stefan Krajewski, Koalicja Polska. Wysoki Sejmie!

Grabicie te samorządy ciągle.

Ile jeszcze takich pieniędzy wydacie bez sensu i kto za to weźmie odpowiedzialność? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie Pośle!

Pan doskonale to wie, a mimo to próbuje pan niestety oszukiwać Polaków w tym względzie. A Niemcy nie chcą nałożyć embarga na rosyjski węgiel, bo są największym eksporterem. Natomiast wracając do tej ustawy, do tej bardzo dobrej ustawy z roku 2016, [[Oklaski]] pragnę przypomnieć, że była to odpowiedź na ogromne żądania Polaków skupionych w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, które sprzeciwiały się dzikiej zabudowie Polski właśnie przez farmy [[Dzwonek]] wiatrowe. Proszę państwa, dzisiaj ta ustawa też ma swoje pozytywy. Natomiast prawda jest taka, że zielona energia to nie tylko farmy wiatrowe.

I ostatnie pytanie zadaje pan poseł Grzegorz Wojciechowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

I budowało się bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na warunkach zabudowy, ludziom zupełnie pod domem, tam gdzie mieszkają.

Proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pana ministra Ireneusza Zyskę o odpowiedź na pytania.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Parlamentarzyści! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować przewodniczącym Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, ale także panu przewodniczącemu komisji samorządu terytorialnego i wszystkim państwu członkom tych komisji za merytoryczną pracę nad projektem ustawy. Dziękuję wszystkim partiom politycznym skupionym w klubach, kołach poselskich za wyrażenie pozytywnej opinii na temat tego projektu. Oczywiście opozycja ma prawo krytykować rząd, realizację projektów podjętych chociażby kilka lat temu.

Dzisiaj w pytaniach większości państwa posłów też ten temat wybrzmiewał. Otóż liberalizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dotycząca warunków odległościowych to jeden z gorących tematów poruszanych od dawna w debacie publicznej. Zmiany w tym obszarze z pewnością korzystnie wpłyną na rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Obecnie trwają prace, które są na ukończeniu, w zakresie licznych wniosków, które wpłynęły w ramach konsultacji publicznych projektu ustawy. To jest minister właściwy do spraw budownictwa, czyli dział budownictwa znajduje się jako właściwy w ministerstwie rozwoju i tutaj bezpośrednio, jeśli chodzi o interpelacje, które do nas wpływają, do mnie osobiście, bo one dotyczą rozwoju odnawialnych źródeł energii, muszę konsultować odpowiedzi albo uzupełniać je o stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Trudno mi składać deklaracje, drodzy państwo, w zakresie terminu, ale powiem w ten sposób, że największe spółki energetyczne, spółki Skarbu Państwa, w tym PKN Orlen czy Polska Grupa Energetyczna, w swoich strategiach rozwoju, realizacji projektów energetycznych zakładają również rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Stąd też myślę, że ta energetyka jest potrzebna. Niestety muszę się nie zgodzić z głosem jednego z parlamentarzystów, który twierdził, że energia wiatrowa jest najdroższa, jest nieekonomiczna. Tak nie jest. Otóż, Wysoki Sejmie, szanowni państwo, w całym życiu.

Świadczą o tym m.in. zakontraktowane na aukcjach OZE projekty. Kontrakt różnicowy, który został przyjęty jako model wsparcia pomocy publicznej notyfikowany przez Komisję Europejską i który od wielu lat funkcjonuje na polskim rynku energii, świadczy o tym, że koszt energii wytworzonej w energetyce wiatrowej na lądzie to ok. 230 zł za 1 MWh, a dzisiejsza cena energii na giełdzie to 576 zł za 1 MWh.

Stąd też trzeba powiedzieć, że energetyka wiatrowa na lądzie mogłaby jeszcze skupić kilka gigawatów mocy pracujących na rzecz polskiego krajowego systemu elektroenergetycznego, wzbogacając polski miks energetyczny. W tej chwili trwa, zaczyna się dyskusja nad pakietem Fit for 55, ale to odrębny temat, którego nie chciałbym w tej chwili poruszać, nie dotyczy on tej ustawy. Niemniej jednak podam kilka informacji, które, myślę, są też ważne dla państwa, którzy się interesują energetyką, którzy przede wszystkim pracują w komisji do spraw energii, ale także w komisji samorządu terytorialnego. Otóż, proszę państwa, nie jest tak, jak niektórzy z państwa, szczególnie z opozycji, sugerowali, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował - nawet bardzo ekstremalne określenia tutaj padały: zabił -energetykę wiatrową na lądzie. Absolutnie jest to nieprawda.

Dzisiaj jest to 6,8, nawet więcej, ponad 6,8, czyli 1 GW mocy został zainstalowany.

Mamy opóźnienie związane z COVID-em, też wprowadziliśmy zmianę w jednej z ustaw COVID-owych, aby umożliwić realizację projektów ze względu na przerwane łańcuchy dostaw, więc w ciągu najbliższych 3 lat na lądzie w Polsce będziemy mieć zainstalowane ok. 11 GW mocy.

Przechodzę do odpowiedzi na pytania.

Otóż tak nie jest. W ostatnich 3, a szczególnie w ostatnich 2 latach, pomimo pandemii koronawirusa w Polsce nastąpił bum inwestycyjny związany z rozwojem fotowoltaiki.

Jedno wyjaśnienie dla Wysokiej Izby, dla szanownych państwa posłów - otóż rząd realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby literalnie trzymać się tego orzeczenia, również pełnego uzasadnienia, to z tego wyroku nie wynika, że ma być to rekompensata za cały rok 2018. Właściwie moglibyśmy poprzestać na połowie roku, czyli byłoby to 6 miesięcy z kilkunastoma dniami.

Po wielogodzinnych rozmowach, nie tylko po samych konsultacjach, ale też później, w trakcie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przyjęliśmy, że chcemy, aby było to obliczone za cały rok.

Ale żeby nie było tak, bo państwo utożsamiają to z tym, że samorządy tracą, że za to płacą mieszkańcy, że ktoś na tym cierpi. Otóż, proszę państwa, z pewnością samorządy utraciły dochody, a teraz naprawiamy tę sytuację. Ale proszę mieć na uwadze, że po drugiej stronie tej samej sprawy był interes inwestorów realizujących inwestycje wiatrowe, właściwie już funkcjonujące farmy wiatrowe, a co za tym idzie - byli tam odbiorcy końcowi energii elektrycznej, czyli de facto byliśmy my wszyscy, całe społeczeństwo.

Uważamy, że tamta decyzja była słuszna, jedyna właściwa w tamtym czasie, w tamtej sytuacji. Otóż, proszę państwa, pan poseł Jan Szopiński pytał o bliźniaczą infrastrukturę kolejową i lotniczą, podobne zależności. Najmocniej przepraszam pana posła, ale to jest pytanie do ministra infrastruktury. Z przyjemnością przekażę panu ministrowi sugestie pana posła.

Ale też - tak jak wcześniej powiedziałem - rekompensata jest za cały rok 2018, a nie za 6 miesięcy, jak wskazywałaby treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Takie sytuacje już w tej chwili się nie zdarzają. Chcę powiedzieć, że dzisiaj ta grupa zawodowa, ta grupa biznesowa energetyki wiatrowej na lądzie to jest elitarny klub. W większości są to przedsiębiorcy, którzy są skupieni w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, które wprowadziło kodeks dobrych praktyk. Dzisiaj jest to partner w dyskusji dla rządu, dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska nad nowymi regulacjami w tym zakresie. Kończąc, chciałbym jeszcze raz podziękować za merytoryczną, rzeczową dyskusję. Wierzę, że ta ustawa zostanie jak najszybciej przyjęta, abyśmy mogli wypłacić rekompensaty gminom w terminie przed 5 lutego 2022 r. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Tak jak podczas posiedzenia komisji, tak i dziś na sali plenarnej rysem charakterystycznym było to, że jeżeli toczyła się dyskusja, to nie nad samą treścią tej ustawy, ona akurat nie wzbudza kontrowersji, tylko wokół ustawy 10H, tak to nazwę, ustawy wiatrakowej.

Szanowne Panie i Panowie Posłowie!

Chociażby drogi lokalne, na których nam zależy, drogi kategorii, gminnej oraz powiatowej.

To rzeczywiście nawet niektórzy z posłów opozycji podczas innych debat, ale też nad tą debatą przyznawali, że wprowadzano wiatraki na zasadzie wolnej amerykanki.

Wracam do polityki samorządowej i do ustawodawstwa samorządowego.

Jeszcze raz: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie polityki samorządowej są kluczem. Teraz zgodzę się z głosami z opozycji.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druki nr 1730 i 1747) Bardzo proszę panią poseł Urszulę Rusecką o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przedkładam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, druk nr 1730, a druk sprawozdania to druk nr 1747. Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 8 listopada 2021 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na wczorajszym posiedzeniu przeprowadziła pierwsze czytanie oraz rozpatrzenie powyższego projektu ustawy. Procedowany projekt ustawy to kolejny krok, to cenna inicjatywa w kierunku zadośćuczynienia prawnego, finansowego i moralnego ludziom, którzy walczyli o naszą wolność. Procedowany projekt, tj. ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym przysługującym działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych, określa warunki nabywania prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zasady wypłaty tego świadczenia. Celem jednorazowego świadczenia jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Prawem do przedmiotowego świadczenia będą objęte osoby, które status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych uzyskały na podstawie decyzji szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych do 31 grudnia 2021 r. Osobie o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie będzie wypłacane z urzędu przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w kwocie 3000 zł i będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego będzie wydawał szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Decyzja przyznająca jednorazowe świadczenie pieniężne nie wymaga uzasadnienia i nadaje się jej rygor natychmiastowej wykonalności. W procedowanej ustawie proponuje się, by świadczenie było wolne od egzekucji i nie podlegało wliczeniu do dochodu uprawniającego do świadczenia i dodatków przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, oraz by było wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt to kolejny projekt ustawy w trwającym od 6 lat procesie przywracania godności działaczom opozycji antykomunistycznej. Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie nowelizował ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, a jej zmiany szły w kierunku rozszerzenia wsparcia udzielanego ww. grupie. Warto wspomnieć, że od 15 października 2020 r. przyznano prawo do świadczenia wyrównawczego, jeżeli osoba o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w kwocie niższej niż 2 501,76 zł brutto miesięcznie. W tej sytuacji osobie tej przysługuje wyrównanie pobieranego świadczenia do tej kwoty. Również w br. weszły w życie nowe regulacje pozwalające na zwiększenie dostępności pomocy pieniężnej.

Wprowadzono również nowy sposób ustalania podstawy wymiaru kapitału początkowego, uznając za okresy składkowe okresy represji politycznych z jednoczesnym przyjęciem kwoty przeciętnego wynagrodzenia za podstawę wymiaru składek w tym okresie. Oznacza to, że emerytury tych osób będą wyższe. Wprowadzono również istotne uprawnienia pracownicze: działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pozostającym w zatrudnieniu przysługuje dodatkowy, 5-dniowy urlop w roku kalendarzowym.

To sposób naprawiania krzywd, jakich doznało wiele osób. Żeby porównać wsparcie - a najbardziej przemawiają do państwa i do osób, które nas słuchają, liczby - powiem tak. Jeżeli chodzi o fundusze, jakie były przeznaczane dla kombatantów i dla działaczy opozycji antykomunistycznej w 2015 r., to była liczba 9 mln. W tej chwili ta liczba wynosi 130 mln. To jest duże wsparcie dla tych osób. Wszystkie działania prowadzą do tego, żeby zadośćuczynić osobom, które w tamtym czasie, w czasie stanu wojennego, w zasadzie od 1956 r. ponosiły ogromne straty moralne, finansowe. W związku z powyższym, zgodnie z ustaleniami komisji, która jednogłośnie o to wniosła, proponuję, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić procedowany projekt ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół.

Osoby o potwierdzonym statusie działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych będą miały prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł.

Dodać można, że działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych mogą skorzystać z innych działań pomocowych wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Szerzej mówiła o tym poseł sprawozdawca, przewodnicząca komisji pani Urszula Rusecka. Powyższe wskazuje, że jesteśmy formacją wiarygodną, konsekwentnie realizującą głoszone deklaracje, w tym przypadku - zwiększenia pomocy dla osób szczególnie zasłużonych dla Polski. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób możemy zrekompensować krzywdy i prześladowania wobec osób, które walczyły o wolną Polskę. Osoby te, podejmując walkę z systemem zła, jakim był komunizm, sprzeciwiały się różnego rodzaju formom nacisku i ucisku, nie bacząc na negatywne konsekwencje, jakie ta walka mogła przynieść i niestety przynosiła, w postaci aresztowań, prześladowań, utraty pracy itp. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Śp. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński był gorącym orędownikiem działań ze strony państwa, które gwarantowałyby opiekę nad członkami PRL-owskiej opozycji. Lech Kaczyński zawsze podkreślał, że Polska musi szanować swoich bohaterów, że jest to obowiązek, który wynika z uczciwości wobec tych osób. Poselski projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, jak również przytoczone rozwiązania prawne, które przedstawiła pan poseł Urszula Rusecka, korzystne dla działaczy PRL-owskiej opozycji, wpisują się w słowa śp. prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, jak również nawiązują do jego koncepcji, wizji niesienia pomocy osobom, które walczyły o wolną i suwerenną Polskę. Jak czytam w uzasadnieniu do projektu ustawy, wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego rozpocznie się w grudniu 2021 r., tj. w miesiącu, w którym przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W przypadku osoby uprawnionej zamieszkałej za granicą jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone byłoby w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą, a wypłata dokonywana byłaby w walucie wymienialnej. Jest to istotne zwłaszcza dla tych, którzy musieli opuścić ojczyznę w wyniku działań represyjnych systemu komunistycznego. W projekcie zapisano też, że świadczenie wraz z kosztami jego obsługi byłoby finansowane w ramach środków budżetu państwa, zaś skutki finansowe proponowanej regulacji są szacowane na ok. 42 mln zł.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, druk nr 1730. Wysoka Izbo! Poselski projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych zakłada przyznanie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł wcześniej wymienionym osobom.

Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska popiera przedmiotowy projekt ustawy, jednak chciałabym zwrócić uwagę, iż środowisko działaczy podziemia antykomunistycznego od kilku miesięcy walczy o włączenie do dyskusji parlamentarnej złożonego 9 lipca br. apelu 258 opozycjonistów i osób represjonowanych, zawierającego przygotowany dokument o nazwie: projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Apel ten został zainicjowany przez pana Jarosława Macieja Goliszewskiego, pana Leszka Stalla oraz dr. Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa i poparty 258 podpisami byłych opozycjonistów i osób represjonowanych. 15 lipca apel wraz z załączonym projektem ustawy został skierowany przez panią marszałek Sejmu do procedowania w komisji. Niestety apel ten utknął w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w czasie procedowania nad przedmiotową ustawą wnioskowałam o rozszerzenie porządku obrad i rozpoczęcie prac nad apelem opozycjonistów. Pan minister Kasprzyk podniósł na wczorajszych obradach komisji konieczność przygotowania przez Instytut Pamięci Narodowej opinii dotyczącej postulatów opozycjonistów zapisanych w przedłożonym apelu. Opinia taka jest w posiadaniu inicjatorów apelu i podpisana została przez prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego w sierpniu br. Przypomnę również, że 14 października wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz wystąpiła z pismem o podjęcie prac nad przekazanym przez opozycjonistów apelem i z propozycją zmian przepisów. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że zarówno apel środowisk działaczy antykomunistycznych, jak i pismo pani poseł zostały zignorowane. Od wielu miesięcy inicjatorzy apelu prowadzili działania mające na celu wprowadzenie przez Sejm zmian do obecnego prawa i włączenie do procedowania przez komisję złożonego przez nich apelu wraz z projektem ustawy, tak aby w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego móc przełamać passę złych wspomnień związanych z tym szczególnym dniem. To oni najlepiej znają problemy swoich kolegów i koleżanek opozycjonistów. To oni są najbliżej środowiska osób represjonowanych. Z prawdziwą pasją poświęcają się słusznej sprawie. Projekt ustawy, który przedstawili wnioskodawcy, zawiera rozwiązania porządkujące zaszłości prawne, godnościowe i bytowe, dotykające byłych opozycjonistów antykomunistycznych i osoby represjonowane. Propozycje zawarte w tym dokumencie zakładają m.in. uhonorowanie i upamiętnienie osób z potwierdzonym statusem działacza opozycji lub osoby represjonowanej, rozszerzenie kręgu uprawnionych do występowania o pośmiertne potwierdzenie statusu działacza represjonowanego o organizacje środowiskowe, samorządy terytorialne i wojewodów czy objęcie przez ZUS miesięcznym świadczeniem zastępczym osób, które mają potwierdzony status działacza lub represjonowanego, ale które wskutek wykluczenia w czasach PRL nie zgromadziły stażu pracy wymaganego do wypłaty emerytury lub renty. Wysoka Izbo! Procedowany dziś projekt ustawy (Dzwonek) zasługuje na poparcie. Zwracam jednocześnie uwagę, że jest to najlepszy czas na zajęcie się również postulatami zawartymi w apelu działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych. W związku z tym, wsłuchując się w głos działaczy opozycji antykomunistycznej, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska składam poprawki do przedmiotowego projektu ustawy i proszę o ich uwzględnienie. Bardzo proszę, pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze! To ważny projekt, w którym Wysoka Izba potwierdza dziś art. 19 naszej konstytucji, który mówi, że Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych. Dziś rozpatrujemy projekt poselski o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Te rozwiązania, o których była mowa już dzisiaj w czasie debaty, dotyczące poprawy warunków życia i funkcjonowania osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej, rzeczywiście w naszym ustawodawstwie w ostatnich latach są powiększane, rozszerzane. Najistotniejszą kwestią z punktu widzenia klubu parlamentarnego Lewicy jest kwestia pewnej równowagi między działaczami opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych a kombatantami okresu powojennego i wojennego. Jak wynikało również z informacji pana ministra, ta grupa osób, kombatantów okresu powojennego, jest objęta pomocą jednorazową, jeśli chodzi o świadczenia z powodu niewystarczających środków do życia.

Powstaje więc pytanie, czy tych środków finansowych mamy wystarczająco dużo, jeśli chodzi o pomoc dla kombatantów okresu powojennego i działaczy opozycji antykomunistycznej. Tak, ta ustawa o jednorazowym świadczeniu mówi o tym, że koszt wdrożenia tego ważnego elementu wsparcia tej grupy osób to kwota 42 mln zł. Szkoda tylko, że nie są to środki w konkretnym miejscu, u pana ministra. One dopiero mają się pojawić w wyniku decyzji prezesa Rady Ministrów.

Zjada trzynastkę i jednorazowe świadczenie, które jest wypłacane. Szanowni Państwo!

Trzykrotnie wyższe koszty utrzymania.

Dlatego też w trakcie prac nad projektem budżetu państwa będziemy wnioskować o zwiększenie tej kwoty, która byłaby w dyspozycji szefa urzędu, na pomoc dla kombatantów oraz działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Klub parlamentarny Lewicy udzieli poparcia temu ważnemu projektowi, dotyczącemu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 tys. zł. Dziękuję. Bardzo proszę, pani poseł Bożena Żelazowska, Koalicja Polska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu dotyczące ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych z druku nr 1730. W tym roku, 13 grudnia, mija 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Pamiętamy - a ci z nas, którzy są młodsi, znają z kart historii i z opowieści - jak trudny dla naszego kraju był to czas, kiedy w Polsce panował komunizm.

Wiele z tych osób było represjonowanych, wielu straciło życie. Po latach ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej osobom tym przyznano status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoby te otrzymały również świadczenie pieniężne i szereg innych przywilejów, takich jak status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej, mogły uzyskać legitymację i tytuł do odznaki honorowej.

Osobie uprawnionej przysługuje również prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej. Samorząd terytorialny może udzielić pomocy działaczom opozycji w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych. Powstał na podstawie propozycji środowiska opozycjonistów, którzy czuli się niesprawiedliwie potraktowani przez obowiązujące przepisy. Ten projekt nie był jednak procedowany. Były to propozycje opozycjonistów i Senatu. Projekt zawierający te same rozwiązania, które proponowało środowisko opozycjonistów i Senat, plus nowe przepisy pojawił się w Sejmie w styczniu br. Dodatkowe przepisy dotyczyły podniesienia progów dochodowych uprawniających do jednorazowej pomocy pieniężnej, okresowej pomocy pieniężnej, zwiększenia kwot świadczeń oraz umożliwienia przyznania pomocy pieniężnej dwa razy w roku, a nie, jak dotychczas, raz na 12 miesięcy. Ta ustawa zapewniła też działaczom opozycji dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego i zwolnienie całkowite lub częściowe z opłat za pobyt w domu opieki społecznej. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej głosował za przyjęciem tej ustawy. Jak wspomniałam, 13 grudnia br. minie 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Z tej okazji przygotowany został projekt ustawy, na mocy której działaczom opozycji antykomunistycznej zostanie przyznane jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3 tys. zł.

Myślę, że jest to dobry moment, abyśmy w ramach solidarności społecznej pamiętali o tych, którzy w tym czasie jako nauczyciele kształtowali serca i umysły młodego pokolenia. Pamiętajmy o rolnikach, których emerytury są dzisiaj rażąco niskie, nie wiem, czy nie najniższe w hierarchii emerytur, którzy również wspierali działania opozycyjne w naszym kraju. Pamiętajmy także o druhach ochotniczych straży pożarnych, którym wciąż obiecywany jest dodatek emerytalny za wieloletnią pracę na rzecz drugiego człowieka, a do tej pory taki dodatek nie został im przyznany i wypłacony. Bardzo proszę, pan poseł Robert Winnicki, Konfederacja. Wysoka Izbo!

Dlatego ta drobna rekompensata, ten drobny jednorazowy gest dla tych kilkunastu tysięcy osób, które z reżimem komunistycznym w imię naszej wolności, suwerenności, w imię tego, żeby Polska była Polską, walczyły, jest rzeczą oczywistą. To jest gest, który im się po prostu należy. Natomiast warto przy tej okazji powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, wydaje mi się, że ciągle w przestrzeni publicznej naszego kraju przykłady heroizmu życiowego nie takiego wielkiego, nie takiego spektakularnego, jaki niektóre legendy mają na koncie, ale takiego heroizmu, który oznaczał lata życia w upokorzeniu, w niedostatku oraz cierpienie prześladowań, jak również głos tych ludzi są mało słyszalne.

Ważne, żeby ta wizja i ich świadectwo, ich przestrzeganie przed tym, czym jest czerwona utopia, czym jest w ogóle utopia realizowana w życiu społecznym, narodowym, ta utopia, która dzisiaj również manifestuje się w postaci sali Spinellego, komunisty, w Parlamencie Europejskim i ma swoją jawną ekspozyturę w bardzo wielu agendach tego nowego projektu po części socjalistycznego, jak również ta pamięć nie zaginęły. Bo utopie czy są czerwone, brunatne, zielone czy jakiekolwiek inne, czy tęczowe, zawsze kończą się fatalnie. Bardzo proszę, pan poseł Paweł Zalewski, Polska 2050. Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy! Trochę nawiązując do mojego przedmówcy, chcę powiedzieć, że również utopia nacjonalistyczna ma taki charakter. Ale nie o tym chciałbym mówić. Pamiętam okres po stanie wojennym, okres wielkiego rozczarowania, kiedy olbrzymia maszyna państwowa zniszczyła marzenia wielu. Okazało się, że nie wszystkich. Nie zniszczyła marzeń, determinacji tych, którzy wtedy podjęli działania, ten wielki mit solidarności, tę wielką ideę solidarności i nieutopijną tym razem, ale praktyczną, prawdziwą ideę, która tak naprawdę sprowadzała się do tego, że chcieliśmy być wolni, chcieliśmy być demokratyczni, rządzić się demokratycznie, chcieliśmy żyć w suwerennym państwie. Otóż byli tacy, którzy tę ideę podjęli. Nie liczyli na żadne uposażenia, żadne apanaże, uważali po prostu, że tak muszą robić. Kontynuowali pracę tych, którzy w latach 70., wcześniej 60. i jeszcze powojennych walczyli o wolność. I mimo że nawiązywali czasami do różnych nurtów polskiej tradycji niepodległościowej, politycznej, mieli bardzo wiele wspólnego, a to, co było wspólne, ukształtowała w nich solidarność.

Powtarzam, tak mało jest tego, co nas łączy, tak bardzo jesteśmy podzieleni, że dzisiaj złożenie wyrazów uznania, hołdu także w ten sposób, także przez jednorazową wypłatę, jest wyrazem jakiegoś instynktu narodowego, chęci obrony tożsamości narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czy ktoś z pań i panów posłów chce jeszcze zgłosić się do zadania pytania? Jeżeli nie, zamykam listę. Bardzo proszę, pan poseł Szopiński, Lewica. Wysoka Izbo!

Duża część bohaterów tamtego okresu nigdy nie występowała o zaświadczenie, że walczyła o wolność ojczyzny. Proszę też o odniesienie się do informacji, że przedmiotowe zaświadczenie przysługuje z urzędu oraz zapisanej kilka linii niżej informacji, że przyznaje je szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Który z tych zapisów jest prawdziwy? Dlaczego projekt w tym zakresie jest niespójny?

Pan poseł Rafał Adamczyk, klub Lewica. Nie ma. Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowny Panie Ministrze!

Chodzi mi o małoletnie ofiary wojny.

Ta sprawa nie jest nowa.

Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Uprzejmie dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Chciałem zapytać o przepis, który znajdziemy w art. 4 ust. 2 pkt 2, który zmierza do tego, aby osobie niepobierającej świadczenia pieniężnego zamieszkałej w kraju przekazywać to świadczenie przekazem pieniężnym na ostatni znany adres używany w korespondencji z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych! Mam zaszczyt i honor mieć status działacza opozycji antykomunistycznej. Traktuję to jako olbrzymie wyróżnienie i jestem z tego dumny.

Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na pewien problem.

Proszę o 15 sekund, pani marszałek.

Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dlaczego apel, o którym tak szeroko mówiła moja koleżanka, pani poseł Joanna Frydrych, podpisany przez 258 działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych utknął w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny pomimo wielu prób, które podejmowaliśmy w celu rozpoczęcia nad nim dyskusji i podjęcia merytorycznej pracy? Z niewiadomych, niezrozumiałych dla nas powodów leży on w zamrażarce komisji. Przecież opozycjoniści wiedzą najlepiej, z jakimi problemami i procedurami administracyjnymi zderzają się na co dzień. Czy dzisiaj, w przeddzień 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, nie należy wreszcie wsłuchać się w ich głos i rozwiązać sygnalizowane przez nich problemy? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przypomnę, że w strefie państw komunistycznych znaleźliśmy się w wyniku decyzji mocarstw.

Całe pokolenia Polaków walczyły o tę wolność i o tym trzeba pamiętać. To nie jest tylko ostatni okres i okrągły stół, który był ważny dla Polski. Mam tu inne zdanie - że drogą pokojową doszliśmy do tej wolności.

Dlatego pytam się.

Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wiele lat działacze opozycji antykomunistycznej czekali na wsparcie ze strony państwa polskiego. Dobrze, że taka ustawa pojawiła się w roku 2015.

Pan poseł Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jako osoba posiadająca status osoby represjonowanej za działalność antykomunistyczną nie zgadzam się z niektórymi wypowiedziami przedstawicieli klubów parlamentarnych opozycji, którzy mówili - tak to wybrzmiało, tak to zrozumiałem, więc przepraszam, być może źle zrozumiałem, ale raczej nie sądzę - że niewiele zrobiliśmy od 2015 r. do chwili obecnej dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych za działalność polityczną. Mam pytanie do pana ministra Kasprzyka, jeżeli dysponuje takimi danymi.

Pani poseł Zofia Czernow, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Chciałam zapytać szefa urzędu do spraw kombatantów, jaki procent żyjących działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych korzysta z pomocy, a jaki procent z tej pomocy nie korzysta ze względu na to, że nie ma takiej wiedzy.

Dlaczego o tym mówię?

Pan poseł Dariusz Bąk, Prawo i Sprawiedliwość.

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Jestem w takiej sytuacji, że znam zarówno z opowieści, jak i bezpośrednio z walki czynnej osoby, które zasłużyły się dla niepodległości Polski, działając w opozycji antykomunistycznej.

Szanowni Państwo! Dzisiaj był wspomniany przez przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Ale aktualny rząd Prawa i Sprawiedliwości robi, proszę państwa, dużo. działacze opozycji antykomunistycznej mają godność i honor i jest im przyjemnie z tego powodu, że jest taki rząd w Polsce, który o nich dba. Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Chciałem zabrać głos, wypowiadając się z perspektywy pełnomocnika szeregu opozycjonistów w rozumieniu ustawy o IPN-ie, i to takich z ważnymi nazwiskami. Otóż należałoby zwrócić uwagę na pewną charakterystyczną sytuację, która dotyczy małżeństw opozycjonistów.

Dlatego też jest prośba, panie ministrze, żeby w porozumieniu z Prezesem IPN-u przeanalizować status tych osób, które będąc w związku małżeńskim, formalnym czy nieformalnym, wspólnie prowadziły działalność opozycyjną, bo niejednokrotnie z takimi sytuacjami się spotykałem. Natomiast zupełnie innym problemem jest to, co powiem w tej chwili.

Dziękuję, panie pośle. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O udzielenie odpowiedzi na pytania pań i panów posłów uprzejmie proszę szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję uprzejmie. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Zacznę od liczb, bo one są ważne, aby uporządkować sprawy związane z tym, kto otrzyma to jednorazowe wsparcie, które w projekcie poselskim związane jest, jak rozumiem, ze zbliżającą się rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Otóż osób, które otrzymały status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, jest 15 218, z czego żyje 13 731. Po potwierdzeniu statusu w ciągu tych 6 lat funkcjonowania ustawy zmarło już 1199 osób. Szanowni Państwo! Tak jak mówili tu parlamentarzyści, nastąpiła istotna zmiana, jeżeli chodzi o opiekę nad działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów politycznych. Ustawa, którą Wysoki Sejm przyjął w 2015 r., wyłoniła z tej grupy zasłużonych w walce o wolność Polski kolejną grupę podopiecznych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Chodzi o to, że w istocie swojej przyznanie statusu miało charakter czysto honorowy i dopiero trzy nowelizacje: z 2017 r., 2020 r. i 2021 r. uczyniły z tej grupy kilkunastu tysięcy osób grupę, która ma takie same uprawnienia jak kombatanci okresu wojennego, czyli ci, którzy objęci są ustawą kombatancką, którzy walczyli z bronią w ręku.

mają wreszcie możliwość korzystania, już teraz dwa razy w roku, z pomocy jednorazowej bądź okresowej, jeżeli np. muszą dostosować mieszkanie do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. Mają też prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Mają oni prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Podwójnie uwzględnia się okres ich działalności, internowania lub podlegania represjom przy ustalaniu kapitału początkowego.

Mają również prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, które opłaca bezpośrednio szef urzędu, jeżeli jest taka potrzeba. I to się niezwykle dobrze sprawdziło w czasie pandemii, kiedy również działacze opozycyjni, oprócz kombatantów, objęci zostali akcją pomocową chociażby dostarczania posiłków, obiadów do domu, aby minimalizować ich kontakt ze światem zewnętrznym. Wreszcie bardzo ważna nowelizacja z ubiegłego roku. Działacze opozycji mają prawo do świadczenia wyrównawczego. Jeżeli posiadają emeryturę lub rentę niższą niż obecnie 2501 zł, a takich osób jest wiele w tym gronie 13 tys., mają oni prawo do świadczenia wyrównawczego, które wypłacają organy emerytalno-rentowe.

Wreszcie w tym roku działacze uzyskali prawo do korzystania z nowego sposobu ustalania kapitału podstawowego w odniesieniu do okresów uznawanych za składkowe. Chociażby dofinansowujemy działaczom opozycji antykomunistycznej pobyt w uzdrowiskach i sanatoriach. Wybierają sanatorium, a urząd, na postawie faktury wystawionej przez uzdrowisko, w kwocie określonej w regulaminie, dopłaca im do pobytu i leczenia uzdrowiskowego. Tak samo objęci są programem dofinansowania zakupu aparatów słuchowych, w ramach którego urząd dofinansowuje taki aparat do kwoty 10 tys. zł na oba uszy, i ten program cieszy się, podobnie jak w przypadku kombatantów wojennych, ogromnym zainteresowaniem. Odpowiadając na pytania pań i panów posłów i porządkując pewne sprawy, w odniesieniu do pytania pana posła Jana Szopińskiego chcę powiedzieć, że status działacza opozycji antykomunistycznej potwierdza szef urzędu do spraw kombatantów na wniosek osoby, która taki status chce posiadać. Przede wszystkim zaczyna się ono od procesu autolustracji, to znaczy osoba, która ubiega się o status działacza, musi przedłożyć decyzję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o tym, że nie współpracowała z organami bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Zazwyczaj - to w odpowiedzi na pytania kolejne - ten proces potwierdzania statusu, jeżeli sprawa jest bardzo prosta i potwierdzona dowodami, dokumentami, zeznaniami świadków, trwa 30 dni. Jeżeli sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo brak dowodów w Instytucie Pamięci Narodowej, brak zeznań świadków, to zgodnie z ustawą takie przypadki rozpatrywane są przez wojewódzkie rady do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej. Ich rekomendacja dla urzędu nie jest wiążąca, ale jest bardzo pomocna. Jeżeli chodzi o środki, jakie na ten cel są przyznawane, na działaczy opozycji antykomunistycznej - to w odniesieniu do pytań pani poseł Anny Kwiecień i pana posła Jana Mosińskiego. Proszę państwa, w 2015 r. na pomoc i dla kombatantów wojennych, i dla działaczy opozycji antykomunistycznej urząd do spraw kombatantów miał zapisaną w budżecie kwotę 9 mln zł w skali roku. A zważą państwo, iż szczególnie w środowisku kombatanckim niestety z uwagi na nieubłagane prawa biologii odpływ naszych podopiecznych jest znaczący i średnia wieku kombatantów wojennych to obecnie 94 lata. To są te dwie wartości: 9 mln w 2015 r. i 130 mln w roku bieżącym. Pani poseł Zofia Czernow pytała, jaki procent działaczy korzysta z pomocy, a jaki nie korzysta. Kiedy ustawa była procedowana w 2015 r., wieszczono, że status otrzyma docelowo 200 tys. osób, ale badacze z Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie redaktorzy Encyklopedii Solidarności, uspokajali, że grupa docelowa, która objęta będzie zapisami ustawy, nie będzie większa niż 30 tys. osób, i po 6 latach funkcjonowania ustawy należy im przyznać rację. Jeżeli osiągniemy w ogóle wynik 30 tys. osób, to będzie to wynik bardzo dobry, biorąc pod uwagę, że po 6 latach status ma, łącznie z nieżyjącymi osobami, 15 tys. osób. My jako urząd - też odpowiadam pani poseł - nie posiadamy przedstawicielstw w terenie. Przy wojewodach działają rady do spraw działaczy. Chodzi o to, aby w państwa biurach, jeżeli przychodzą zainteresowani, pomóc - wszystkie materiały są czytelne, dostępne na stronie urzędu i nie tylko - w wypełnieniu wniosku i złożeniu go do urzędu.

Takich małżeństw mamy sporo, małżeństw, które są nadal czy też były wtedy małżeństwami. Każda z tych osób ma indywidualne prawo ubiegania się o status działacza czy osoby represjonowanej z powodów politycznych. Chciałbym się też odnieść do pytania pana posła Tadeusza Tomaszewskiego dotyczącego dzieci wojny, choć nie jest to przedmiotem tego projektu, który jest procedowany. To też wybrzmiało w wystąpieniu pana posła Marka Dyducha. Szanowni państwo, małoletnie ofiary wojny, które z różnych powodów były represjonowane czy to przez narodowych socjalistów niemieckich, czy to przez bolszewików, czyli były więźniami obozów koncentracyjnych, były zesłane na roboty przymusowe w głąb III Rzeszy czy były zesłane na nieludzką ziemię, w głąb Związku Sowieckiego, posiadają od 30 lat uprawnienia kombatanckie.

A co z dziećmi, które się urodziły w latach 30. i przeżywały wojnę jako ośmiolatki?

Natomiast powtórzę: dzieci, które, tak jak i dorośli, były poddane represjom czy to ze strony Niemców, czy Sowietów, uprawnienia kombatanckie posiadają. Mamy przecież przypadki dzieci narodzonych np. w Auschwitz - i one mają uprawnienia kombatanckie, czy też przypadki dzieci zesłanych na niewolniczą pracę w głąb III Rzeszy czy w głąb Związku Sowieckiego. Szanowni Państwo! Raz jeszcze, kończąc, chciałem podziękować za ten projekt. To jest też projekt, który - raz jeszcze powtórzyć warto - ma charakter jednorazowej wypłaty dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, jednorazowej, bo związanej z rocznicą.

O możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania postawione Wysokiej Izbie prosiła również sprawozdawca komisji pani poseł Urszula Rusecka. Bardzo proszę, pani poseł. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! Ja chciałabym z tego miejsca bardzo podziękować wszystkim klubom parlamentarnym, członkom Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za pozytywne opinie w sprawie ww. projektu ustawy, podziękować posłom wnioskodawcom tego projektu, posłom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Natomiast muszę odnieść się jednym zdaniem do słów, które tutaj przytoczyła pani poseł Koalicji Obywatelskiej, dotyczących przygotowanego przez grupę opozycjonistów, a tak naprawdę będącego inicjatywą trzech osób projektu ustawy, który wpłynął do komisji. Tak, faktycznie, takie propozycje projektu ustawy do komisji wpłynęły.

Natomiast jeżeli chodzi konkretnie o projekt i inicjatywę, która wpłynęła ostatnio do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, to pragnę zapewnić osoby, które złożyły te propozycje, że pochyliliśmy się szczegółowo nad zapisami i propozycjami zawartymi w projekcie przesłanym do komisji, jednak nie mogliśmy nadać im biegu, ponieważ zawarte tam rozwiązania nie uzyskały pozytywnych opinii merytorycznych urzędów. Przykładem jest chociażby propozycja zmiany definicji współpracy z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa czy wprowadzenie rozwiązania, na podstawie którego publikowane byłyby w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, listy osób, którym nadano Krzyż Wolności i Solidarności, zawierających imię, nazwisko tej osoby oraz datę potwierdzenia statusu.

Bardzo dziękuję panu ministrowi i reprezentującemu przez niego Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wsparcie i pomoc w przygotowaniu ustawy, jak również pani minister Annie Schmidt, reprezentującej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, która pochylała się i nad propozycjami, i nad przygotowanym projektem ustawy. Jeszcze raz z tego miejsca bardzo dziękuję.

W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny celem przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druki nr 1729, 919 i 1736) Uprzejmie proszę pana posła Szymona Pogodę o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia wysokich komisji. Na podstawie art. 39 ust. 2 regulaminu Sejmu Sejm na 42. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r. po przeprowadzeniu pierwszego czytania skierował do wspólnego rozpatrzenia przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisję Infrastruktury rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 1729, oraz senacki projekt ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 919. Komisja na wspólnym posiedzeniu uznała za wiodący rządowy projekt o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 1729, i poddała go szczegółowemu rozpatrzeniu. Jedną z najistotniejszych zmian procedowanej ustawy jest doprecyzowanie zakresu zwolnienia gruntów z infrastrukturą kolejową z podatku od nieruchomości zajętych przez podmioty, które nie prowadzą działalności kolejowej. Obecnie regulacje w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zwalniają z podatku od nieruchomości grunty, na których znajduje się infrastruktura kolejowa. Powyższy przepis jest wykorzystywany do unikania opodatkowania gruntów, na których znajduje się infrastruktura kolejowa, przez podmioty nieprowadzące działalności kolejowej. Interpretacja przepisów pozwalała unikać opodatkowania od podatku od nieruchomości m.in. przez kopalnie czy galerie handlowe, czego skutkiem jest utrata części dochodów przez gminy. W procedowanej ustawie zaproponowano zmiany w art. 7, które uszczelniają system zwolnień oraz wykluczają możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku gruntów lub ich części zajętych na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności innej niż związana z wykonywaniem zadań zarządcy infrastruktury kolejowej lub świadczeniem usług przez operatora obiektu infrastruktury usługowej w rozumieniu załącznika nr 2 ust. 2 i 3 do ustawy o transporcie kolejowym. Pierwsza o charakterze redakcyjno-technicznym, druga wprowadzająca istotne zmiany merytoryczne.

Wykorzystywanie zwolnienia od podatku przez podmioty nieuprawnione motywuje do jak najszybszego wprowadzenia przepisów w życie. Poprawka wprowadziła również zapis w zakresie dotyczącym zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład obiektu infrastruktury usługowej, mowa o terminalach towarowych.

Wszystkie zgłoszone poprawki oraz cały projekt ustawy uzyskały pozytywną rekomendację wysokich komisji. Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy wnoszą o przyjęcie przez Wysoką Izbę ustawy wraz ze zgłoszonymi poprawkami.

Bardzo się cieszę, że wspólnie ponad podziałami mogliśmy tę zmianę przeprowadzić. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowych oświadczeń w imieniu kół. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi pan poseł Mariusz Trepka. Zapraszam.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Omawiany projekt dotyczy doprecyzowania zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości, jeśli chodzi o grunty kolejowe, w szczególności grunty zajęte na prowadzenie działalności przez zarządców infrastruktury kolejowej i operatorów. Projektowany przepis pozwoli na obciążenie podatkiem części gruntów, budynków lub budowli wykorzystywanych do działalności komercyjnej, tj. np. dzierżawionych, wynajmowanych przez podmioty prowadzące inną działalność niż przewoźnika kolejowego albo operatora stacji pasażerskich. Wejście w życie powyższych regulacji powinno skutkować zwiększeniem wpływów podatkowych do części budżetu gmin w związku z uszczelnieniem korzystania ze zwolnień z opodatkowania w obszarze kolejnictwa. Zaproponowane rozwiązania zmierzają do eliminacji zgłaszanego przez jednostki samorządu terytorialnego problemu unikania opodatkowania przez podmioty prowadzące inną niż kolejowa działalność gospodarczą.

Wysoka Izbo!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 Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska przedstawi pani poseł Zofia Czernow. Zapraszam. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska wobec sprawozdania Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej dotyczącego senackiego i rządowego projektów ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, druk nr 1736. W trakcie prac połączonych komisji udało się wiele spraw wyjaśnić, doprecyzować i uzyskać częściowy kompromis, co z satysfakcją stwierdzam.

To wielka ulga i radość w samorządach. 200 mln zł wpłynie do samorządów i będzie wykorzystane do finansowania pilnych zadań mieszkańców, bo najczęściej dotyczyło to biednych gmin. Po drugie, udało się uzyskać kompromis dotyczący terminu wejścia w życie ustawy.

To pozwoli na to, żeby konstytucyjna zasada polegająca na unikaniu.

Podatki to jest domena Komisji Finansów Publicznych.

Tego do tej pory nie wiemy. Dlatego zgłaszam poprawkę w imieniu klubu Koalicja Obywatelska, aby zwolnienie z obowiązku płacenia podatku trwało nie dłużej niż przez okres 5 lat. Chodzi o to, aby był to instrument mobilizujący do większej dbałości o majątek i jego wykorzystanie. Pozostałe ulgi wymagać będą monitoringu w ciągu roku podatkowego i sądzę, że w przyszłości można będzie określić skutki ich obowiązywania. Klub Koalicji Obywatelskiej, mając na uwadze cały ten projekt i to, jakie skutki on powoduje, poprze ten projekt, oczywiście licząc, że ta poprawka zostanie przyjęta.

Dziękuję, pani poseł. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W drugim czytaniu ustawy mamy dużą szansę, graniczącą z pewnością, że zainteresowane samorządy od 1 stycznia 2022 r. otrzymają należne podatki i będą mogły budować i remontować drogi, szkoły czy przedszkola. Praca nad ustawą o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przebiega ponad podziałami, to ważne. Jest to ustawa długo wyczekiwana szczególnie przez te gminy, które spotykały się z nadużywaniem obecnie obowiązujących zapisów ustawy przez część przedsiębiorców nieprowadzących działalności zarządcy na rynku kolejowym, wykorzystujących przepisy do unikania opodatkowania. Problem ten miał ogromny wpływ na uszczuplenie przychodów z podatku od nieruchomości do budżetów gmin i był on znany rządowi od momentu wejścia w życie niefortunnych dla samorządu terytorialnego, znowelizowanych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nomen omen, z dnia 16 listopada 2016 r. W konsekwencji wiele z planowanych przez samorządy terytorialne inwestycji nie zostało zrealizowanych lub ich realizacja uległa opóźnieniu. Przykładem w regionie legnicko-jeleniogórskim może być Osiecznica czy Nowogrodziec. Zwrot takiej kwoty dla tak małej gminy niesie za sobą skrajnie niebezpieczne konsekwencje finansowe. Praca nad zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych pokazuje podwójne standardy w pracy legislacyjnej prowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość. Jedne ustawy procedowane są błyskawicznie, a prace nad innymi przedłużają się, co oznacza ryzyko dla stabilności finansowej samorządu terytorialnego. To, co pokazuje pewną iskrę optymizmu, to przede wszystkim dzisiejsze prace nad niniejszą ustawą w sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Mimo pewnych wątpliwości wszystkie siły polityczne w duchu przekonania o konieczności zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej i rozwoju gmin w Polsce poparły propozycje zawarte w prezentowanej ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Biorąc pod uwagę pozytywne opinie gmin w zakresie przepisów, które znalazły się w niniejszej ustawie, i konieczność jak najszybszego rozwiązania zaistniałej sytuacji prawnej, klub Lewicy będzie głosował za przedstawioną przez Ministerstwo Infrastruktury ustawą. Liczymy też na ponadpartyjne dalsze działanie i przeprocedowanie tejże ustawy na najbliższym posiedzeniu Senatu oraz bezzwłoczne - bez względu na to, jak groteskowo to zabrzmi - podpisanie ustawy przez pana prezydenta. Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Panie i Panowie. Posłowie! Panie Ministrze!

Po pierwsze, to jest w ogóle coś niezwykle rzadko spotykanego - mówili o tym przedmówcy - że jesteśmy w stanie w Izbie sejmowej doprowadzić do takiego ponadpartyjnego, ponadklubowego, wspólnego sposobu myślenia nad rozwiązaniami problemów, które są przed nami.

I tu jesteśmy też na dobrej drodze, żeby to rozwiązać, żeby nie było równych i równiejszych przedsiębiorców.

Bardzo proszę. Uprzejmie dziękuję. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Koła Parlamentarnego Polska 2050 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przedstawiony projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Tak jak tutaj już wielokrotnie zostało wspomniane, zasadniczym celem tego projektu jest likwidacja pewnej luki w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Na skutek tej luki zwolnienie podatkowe jest stosowane do różnego rodzaju działalności, pod warunkiem że jest ona prowadzona na gruntach kolejowych. To jest oczywiście niedopuszczalne, dlatego że to zwolnienie powinno przysługiwać wyłącznie tym, którzy na tych gruntach kolejowych prowadzą działalność kolejową, czyli np. w zakresie infrastruktury kolejowej czy też przewozów kolejowych. I ten projekt ustawy tę sytuację normuje.

Wydaje się, że to jest dobre rozwiązanie również dlatego, że począwszy od dnia 1 stycznia, to uprzywilejowanie podatkowe, które nie powinno mieć miejsca, zostanie zakończone, a z drugiej strony wspólnoty samorządowe, czyli mieszkańcy tych miejscowości, które posiadają tego rodzaju grunty, które są zwolnione z podatku od nieruchomości, będą mogli dysponować większą kwotą, np. na wydatki inwestycyjne, na remonty czy też na prowadzenie edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Jako pierwszy pytanie zada pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Bardzo proszę. Powszechnie wiadomo, że utrzymanie dworców kolejowych w małych miastach i miejscowościach nie jest rentowne. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w dużych miastach, gdzie obiekty takie pełnią rolę centrów handlowych z licznymi sklepami, punktami gastronomicznymi czy usługowymi.

Mam jednak pytanie na przykładzie dworca kolejowego w Bydgoszczy, w którego bryle bardzo dużą powierzchnię zajmuje taras widokowy, wprawdzie nigdy nie oddany do użytku i niepełniący swojej roli, ale istniejący. Nie jest on związany ani z infrastrukturą kolejową, ani z działalnością gospodarczą. Gdybym mógł otrzymać odpowiedź na piśmie, byłbym wielce zobowiązany? Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Rozmawiamy tutaj o zwolnieniach z podatku, rozmawiamy o różnych nieruchomościach, które są z podatku zwalniane. Przez to samorządy nie mają odpowiednich dochodów. Panie Ministrze! Kolejne rzeczy i kolejne tematy czekają. Mam nadzieję, że ta ustawa, nad którą dzisiaj procedujemy, będzie szybko wprowadzona w życie i samorządy nie będą już traciły swoich dochodów. Dziękuję. Wysoka Izbo! Dlaczego Ministerstwo Infrastruktury, posiadając informację od organizacji samorządowych działających w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz zespołu ds. infrastruktury rozwoju lokalnego, polityki regionalnej, a także wiedząc, że grupa senatorów wystąpiła z inicjatywą legislacyjną, a nawet przedłożyła projekt marszałkowi Senatu w tej sprawie, nie kwapiło się z wprowadzeniem tych niezwykle ważnych dla samorządu terytorialnego zmian? Skala problemu, który stara się naprawić procedowana ustawa, jest ogromna. Wpłynęło to negatywnie na budżety tych gmin, nieraz paraliżując bądź opóźniając planowane inwestycje. Czy ministerstwo planuje wypłacenie rekompensat tym gminom, które w wyniku wadliwych przepisów najbardziej ucierpiały finansowo? Dziękuję. Pan poseł Robert Obaz, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu: Osiecznica - 1 mln zł rocznie. Mam takie pytanie: Czy państwo policzyli, ile straciły samorządy w całej Polsce i czy planujecie jakikolwiek zwrot w formie subwencji na inwestycje, przesunięcia pieniędzy na budowę dróg czy też odnowienia infrastruktury kolejowej akurat w tychże gminach? Dziękuję bardzo. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.

Wysoka Izbo! Panie ministrze, chciałem wrócić do tematu, który już sygnalizowałem, i bardzo bym prosił o to, aby pan minister był uprzejmy odpowiedzieć na piśmie na to moje pytanie. Ono dotyczy terenu kolejowego, a konkretnie bocznicy w Bielsku Podlaskim, która to bocznica ma zostać z końcem roku zlikwidowana. Tam jest taka sytuacja, że chyba nieuczciwy deweloper wybudował budynki mieszkalne i w związku z pewnym poziomem hałasu pojawił się problem wśród mieszkańców.

Natomiast bardzo bym prosił, żeby ministerstwo było uprzejme odpowiedzieć (Dzwonek), czy zamierza ten problem rozwiązać, czy będzie dążyło do likwidacji tej bocznicy? Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Dyduch, klub Lewica. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Jest taki konkretny przypadek. Były kamieniołomy, polski inwestor je kupił.

Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub Lewica. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Wysoka Izbo!

Kilkuset milionów złotych, które utracą gminy województwa kujawsko-pomorskiego, nie zrekompensują na pewno Program Inwestycji Strategicznych ani ta ustawa. Bydgoszcz - strata w podatkach lokalnych 140 mln zł, prawie 20 mln - Inowrocław, 10 mln - Świecie, 7 mln - Nakło, 4 mln - Tuchola, prawie 5 mln - Żnin. To są tylko nieliczne miasta w województwie kujawsko-pomorskim, a tak duże straty. Apeluję o to, aby ministerstwo finansów za zadaniami, które deleguje, przekierowało również środki, a utracone pieniądze rekompensowało, bo samorządy bez tych pieniędzy sobie nie poradzą. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Koalicja Polska. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję.

Czy właściciel galerii, który funkcjonuje na gruntach nienależących do kolei i ten, który wybudował galerie na gruntach należących do kolei, będą funkcjonować na podobnych warunkach?

Czy będą funkcjonowali na tych samych warunkach czy nie? Lista posłów zapisanych od głosu została wyczerpana. Uprzejmie proszę sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana ministra Andrzeja Bittela o udzielenie odpowiedzi na postawione pytania. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Ja się też bardzo cieszę z tej dyskusji, która odbyła się na sali plenarnej. Tam można było rzeczywiście więcej kwestii poruszyć, powiedzieć bardziej szczegółowo i dlatego też myślę, że lista pytających jest krótsza. W tej procedurze wiele spraw zostało wyjaśnionych. Jeśli chodzi o pytania dotyczące galerii handlowych, to według mojej wiedzy, jeśli galeria handlowa została wybudowana na terenie kolejowym, to już dawno z tego terenu kolejowego została wyłączona i z całą pewnością jest opodatkowana podatkiem od działalności gospodarczej, podatkiem od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Również te przypadki zbadamy, mam zweryfikowany jeden, podczas prac nad tym projektem w Senacie będę miał zweryfikowane wszystkie galerie wybudowane nad torami, przy torach, jest kilka takich obiektów w Krakowie, w Warszawie. Na pewno Galeria Krakowska, panie pośle, to do pana, płaci podatki od nieruchomości. Chciałbym więc tę galerię zostawić już lekko na boku, bo w tym porządku prawnym, który obowiązuje, i w tym, który jest projektowany, te części budynków, obiektów lub gruntów, które służą działalności komercyjnej, powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Znaczy sprzedaż w galerii handlowej nie służy bezpośrednio obsłudze podróży. W związku z tym nie powinno być wątpliwości co do zakresu opodatkowania. Organ podatkowy, samorząd ma prawo to kontrolować, powinien takie sprawy pilnować, kontrolować.

Efektem tej rozmowy, również tej ostatniej dyskusji, jest ten projekt ustawy. On był pierwotnie odrobinę szerszy, po dyskusji z samorządami, z korporacjami samorządowymi jest odrobinę krótszy. Uznaliśmy, że to już jest temat, który należało zamknąć. Punkt trzeci. W mojej ocenie przepisy obowiązujące nie uzasadniają zwalniania z opodatkowania tych przedsiębiorców, o których była mowa, którzy korzystają z luki.

Dziękuję bardzo. Jestem rad, że jeszcze się spotkamy w komisji w ramach prac nad poprawką, tylko wydaje mi się, że ona dotyczy nie tego tekstu ustawy, który został przyjęty w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej celem przedstawienia sprawozdania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 13. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druki nr 1728 i 1739) Uprzejmie proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, pani poseł. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawiam sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Projekt jest zawarty w druku nr 1728, a sprawozdanie komisji jest w druku nr 1739. Wysoka Izbo!

Wysoka Izbo! Oczywiście rząd nie chce tego sporu z Komisją Europejską eskalować i stąd przygotowany jest projekt ustawy, o którym mówimy. Zmiany zawarte w tej ustawie obejmują: po pierwsze, uchylenie w ustawie o lasach przepisów, które dotyczą wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej oraz zmianę przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących tychże wymagań dobrej praktyki; po drugie, dodanie w ustawie o ochronie przyrody art. 52b zobowiązującego właścicieli lasów do stosowania wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej i to zarówno na etapie przygotowywania, jak i na etapie realizacji działań z zakresu gospodarki leśnej oraz przepisu zawierającego delegację ustawową dla ministra właściwego ds. środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej z uwzględnieniem zapewnienia ochrony gatunków, celów, zasad gospodarki leśnej oraz wymogów gospodarczych, społecznych i kulturowych - tenże kodeks dobrych praktyk będzie przeciwdziałać występowaniu potencjalnych kolizji działań w zakresie gospodarki leśnej z elementami środowiska; po trzecie, doprecyzowanie w omawianym projekcie art. 52 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody w oparciu o art. 12 i art. 13 dyrektywy siedliskowej poprzez wskazanie, że odstępstwa nie dotyczą gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy dyrektyw. Wysoka Izbo!